Szanowny Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata, świata po koronawirusie. Wiemy doskonale, że to, co dzieje się dzisiaj, będzie miało wpływ na Polskę, na Europę za 5, za 10 lat. Polska potrzebuje podejścia, które będzie najbardziej właściwe dla realizacji jej interesów. Chciałbym zacząć od tego, żeby zadać takie jedno proste, a zarazem najważniejsze pytanie - właśnie czego potrzebują dzisiaj Polacy. Otóż Polacy potrzebują dzisiaj przede wszystkim skuteczności, sprawiedliwości, potrzebują tego, żeby nasze działania miały wpływ, [[Oklaski]] realny wpływ na rzeczywistość zdrowotną i rzeczywistość gospodarczą. I w takich okolicznościach, w jakich jesteśmy, Polacy nie potrzebują waszych awantur, nie potrzebują jałowych dyskusji. Nie potrzebują też Polacy waszego pieniactwa, nie potrzebują awantur. Polacy potrzebują stabilności i spokoju, potrzebują działania na rzecz dobra Rzeczypospolitej. Proszę państwa, proszę pozwolić na wypowiedź. Państwo będziecie mieć czas na zadawanie pytań, na wystąpienia. Polacy zadecydowali, żeby złożyć los Polski na kolejne 4 lata w ręce rządów Zjednoczonej Prawicy.

I to jest silny mandat, który my chcemy dzisiaj wykorzystać po to, żeby Polska była w taki sposób zbudowana po koronawirusie, żebyśmy skorzystali na tym, a nie żeby w tych trudnych okolicznościach, w których się znaleźliśmy, Polska była w ogonie Europy. rzeczywistości, która nas otacza, kiedy w Stanach Zjednoczonych sytuacja jest bardzo trudna i w obszarze pandemii, w obszarze służby zdrowia, i oczywiście również w gospodarce, i widzimy zamieszki polityczne. kiedy Europa powoli wychodzi z kryzysu zdrowotnego i wpada bardzo głęboko w kryzys gospodarczy, kiedy drży w posadach porządek i ład międzynarodowy na Dalekim Wschodzie - widzimy, co dzieje się wokół Chin - kiedy już nie miliony osób, ale miliardy osób na świecie drżą o swoje miejsca pracy, w takiej sytuacji potrzebujemy jedności. Jedności między władzą wykonawczą, władzą ustawodawczą, między Sejmem, Senatem, panem prezydentem, rządem i samorządami. Bardzo tego potrzebujemy. I dlatego w ostatnich kilku dniach rozmawiałem z panem prezydentem. Pan prezydent zaproponował, żeby przeciąć ten festiwal, który państwo próbujecie urządzać. Prezes. ...ten festiwal awantur, i żeby po prostu powiedzieć: sprawdzam. Jeżeli macie wystarczającą liczbę głosów, to odwołajcie nas albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić. przestańcie wymyślać tematy zastępcze: [[Oklaski]] raz odwoływanie pana premiera Sasina, dzisiaj ministra Szumowskiego, zapowiadacie odwoływanie pana ministra Ziobry, pana ministra Kamińskiego. To wszystko są polityczne sztuczki, które mają przykryć naszą rzeczywistość.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Kilka zdań chcę powiedzieć, ponieważ jest to prośba o wotum zaufania do mojego rządu, o naszych osiągnięciach, o tym, co udało się zrobić w ostatnich kilku latach. Otóż 5 lat temu doszło do fundamentalnej zmiany. Drzwi do tej dobrej zmiany otworzył pan prezydent Andrzej Duda. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. I ta zmiana potem była realizowana w ramach nowej polityki społecznej, nowej polityki gospodarczej, najpierw przez gabinet pani premier Beaty Szydło, którego miałem zaszczyt być członkiem, a później kontynuowany również przeze mnie i przez rząd, który tutaj z nami dzisiaj się znajduje. To zupełnie nowa polityka, polityka, która miała na celu przesunąć tę zwrotnicę rozwoju, zwrotnicę modernizacji w kierunku zwykłego człowieka. Dziękuję, panie prezydencie. Ale też ta polityka, ta zupełnie nowa polityka dla dobra ludzi nie byłaby możliwa, gdyby nie zjednoczenie sił patriotycznych wokół tego wspólnego celu, wspólnego dobra, jakim jest silna, sprawiedliwa, dostatnia Rzeczpospolita. Dlatego dziękuję bardzo zarówno Porozumieniu pana Jarosława Gowina, jak i Solidarnej Polsce pana Zbigniewa Ziobry, które przyłączyły się i które są z nami przy tym dziele naprawy Rzeczypospolitej. Pan minister Zbigniew Ziobro bardzo zdecydowanie stara się naprawić coś, co jest jedną z najpotężniejszych pięt achillesowych III Rzeczypospolitej: wymiar sprawiedliwości. I tutaj, szanowni państwo, dla tych z państwa, którzy choćbyście mieli np. jakieś wątpliwości czy zastanawiali się, to mam tylko jedną taką bardzo drobną sugestię: sięgnijcie sobie tak raz na miesiąc, raz na 2 miesiące do ostatnich wyroków wydawanych przez polskie sądy w zwyczajnych sprawach, kryminalnych, cywilnych, takich czy innych, jak niedawno sąd w Zamościu, który skazał przestępców na 4 i 5 lat więzienia, przestępców, którzy tępym narzędziem zamordowali na oczach matki i jej dzieci mężczyznę z premedytacją i w wyjątkowo bestialski sposób, albo sąd w Elblągu, który w zawieszeniu skazał mężczyzn za gwałt, a później jeszcze sąd bodaj wyższej instancji nałożył karę grzywny za niestawienie się dla tej kobiety przed oblicze sądu, bo nie chciała oglądać twarzy swoich oprawców. To są wyroki sądów Rzeczypospolitej. Z tym walczy pan Zbigniew Ziobro, pan minister Zbigniew Ziobro. I bardzo dziękuję panu ministrowi za to. Walczymy również o jak najlepsze środowisko dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo one są solą ziemi. Dziękuję bardzo panu premierowi Jarosławowi Gowinowi i partii Porozumienie za reformy, za dbanie o małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanowni Państwo! które próbujecie zakrzyczeć, próbujecie przez swoje awanturnictwo zamazać, ale podkreślam: to są liczby, które bardzo łatwo sprawdzić i które przemawiają na rzecz skutecznych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, po pierwsze, bezrobocie spadło do poziomu drugiego najniższego w Unii Europejskiej.

Po drugie, wzrost PKB - 4,2 średnio w ostatnich kilku latach, dwa razy szybciej niż w Unii Europejskiej, trzy razy szybciej niż w państwach strefy euro. Tego się nie da zakrzyczeć, tego się nie da przykryć. Pensje. Pensja minimalna - z 1750 zł do 2600 zł, wzrost o blisko 50%. Nigdy wcześniej, w poprzednich czterolatkach, nie było tak szybkiego wzrostu realnych wynagrodzeń Polaków jak w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Obniżenie podatków, podatku CIT - z 19 do 9%, podatku PIT - o 6%, o 1 punkt procentowy, czyli 6% mniej więcej, z 18 na 17, i to dla 24 mln naszych rodaków. Poprzez matrycę VAT obniżenie również podatku VAT dla bardzo wielu towarów. Wreszcie to wszystko, te wszystkie wielkie programy społeczne, które zmieniły życie milionów Polaków, dziesiątków milionów Polaków: 500+, „Emerytura+”, obniżenie wieku emerytalnego czy wreszcie zerowy podatek dla młodych, po to żeby tu zostawali. wykorzystywali swoje talenty, swoją kreatywność, [[Oklaski]] a nie oferta, którą wy mieliście: weź kredyt, zmień pracę albo wyjedź sobie za granicę. Wszyscy Polacy muszą tu mieć miejsce, muszą tu mieć swój dom i dlatego te nasze działania zmierzały ku temu, żeby stworzyć jak największą liczbę miejsc pracy. Ponad 2 mln nowych osób pracujących, osób, które budowały polski dobrobyt, polskie PKB. Wyprzedzaliśmy również wzrostem gospodarczym średnio państwa Grupy Wyszehradzkiej. I to jest miara naszego sukcesu, realna miara gospodarcza, którą poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez usprawnienie instytucji. W komunie trudno mówić o instytucjach podatkowych, a przez 30 lat, przez 25 lat były praktycznie traktowane jak piąte koło u wozu. Bez sprawiedliwie płaconych podatków nie ma sprawiedliwego państwa. Tak, jeszcze przed nami daleka droga, [[Oklaski]] ale idziemy ku coraz bardziej sprawnym instytucjom i jestem przekonany, że to w kolejnych latach również przełoży się na zwiększenie dobrobytu całego państwa polskiego. Tymczasem dzisiaj wszyscy, cały świat rozmawia o koronawirusie, więc ja też chcę teraz przejść do części dotyczącej epidemii, dotyczącej pandemii. Otóż w momencie, kiedy cały świat zaczął się zmagać z koronawirusem, nie było żadnych podręczników walki z taką pandemią, nie było żadnych dobrych doradców, nie było kogoś, kto dałby jedyną dobrą radę. I właśnie w tym czasie my musieliśmy podejmować decyzje, czasami z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Przy waszym trybie podejmowania decyzji w poprzednich latach, jestem przekonany. Zresztą zaraz spróbuję wykonać taki eksperyment, jeśli ktoś chciałby usłyszeć, jak by to wyglądało, bo za waszych czasów też była epidemia, dużo mniej groźna. Przypomnę, jak reagowali wasi ministrowie zdrowia i wasi premierzy. Jak najszybciej zamknęliśmy granice celem dokonywania kontroli sanitarnych. Zamknęliśmy imprezy masowe 6 dni po pojawieniu się pierwszego przypadku w Polsce. W Niemczech, Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii taka sama zasada została wdrożona po 40 dniach. I to jest właśnie sztuka: sztuka podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie. I nie damy sobie wmówić przez was, że dwa razy dwa jest pięć albo że prawo to lewo, a lewo to prawo. Prawda jest taka, że odnieśliśmy ogromny sukces w walce z koronawirusem, [[Oklaski]] sukces, który jest dostrzegany przez wszystkich na całym świecie. W waszych ławach pojawiały się głosy: model zachodni, model szwedzki. Przeczytajcie sobie wczorajszą wypowiedź głównego epidemiologa Szwecji, jak przyznaje się do błędów, przyznaje się do winy. Mówi: dzisiaj już wiem, że nasze działania powinny być szybsze, były spóźnione. To mówią Szwedzi o Szwecji. Zobaczcie, jaki jest poziom zgonów na 1 mln mieszkańców w państwach daleko bogatszych od nas. Popatrzcie na Hiszpanię i na Włochy, gdzie osoby były chowane w samotności, bez bliskich. Popatrzcie na Stany Zjednoczone, gdzie w Nowym Jorku niestety musiały być przygotowywane mogiły zbiorowe. W Brazylii podobnie. A są inne kraje świata, gdzie z braku trumien ludzi musiano chować w kartonach. I to, że nie doszło u nas do żadnej takiej tragedii, to, że u nas nie zabrakło respiratorów, nie zabrakło łóżek, mieliśmy zawsze ich nadmiar, to jest skuteczna polityka rządu Zjednoczonej Prawicy, [[Oklaski]] to jest skuteczna polityka ministra zdrowia Zjednoczonej Prawicy pana Łukasza Szumowskiego. Nawet w jednym z absolutnie najbogatszych krajów świata jak Szwajcaria jest osiem razy więcej zgonów. W Wielkiej Brytanii - ponad 20 razy więcej zgonów, w Belgii - 32 razy więcej zgonów niż w Polsce. Nawet w krajach środkowej Europy, jak Węgry, czy północnej Europy, jak Finlandia, jest dwa razy więcej zgonów niż w Polsce. To jest miara naszej skuteczności. I to jednocześnie oznacza, drodzy rodacy, że wszystkie te próby przykrycia prawdy, przykrycia prawdy o walce z epidemią są jedynie przygrywką polityczną, są jedynie próbą zamazania rzeczywistości takiej, jaką ona jest.

Nie dajmy sobie, rodacy, tego wmówić.

Pani marszałek Kidawa-Błońska mówiła o tym, że ukrywamy pierwszy przypadek koronawirusa. Dzisiaj, teraz nawet kiwa głową. Pan przewodniczący Budka mówił, że nie testujemy po to, żeby ukrywać prawdziwe dane. Szanowni Państwo! Te wszystkie rzeczy, które dzisiaj wyraźnie widać. W jaki sposób to przeprowadziliśmy? Skutecznie. I w rzeczywistości, tak jak pokazywałem nawet z tej mównicy, chcemy przesuwać ten szczyt zachorowań na koronawirusa, wypłaszczać krzywą. To wszystko zostało zrealizowane zgodnie z planem. Po co się wypłaszcza tak tę krzywą? Po to, żeby nigdy nie zabrakło łóżek, żeby nigdy nie trzeba było dokonywać selekcji, Wysoka Izbo, selekcji, jaka się odbywała w najbogatszych krajach świata. Tak było w tych bogatych krajach.

Żaden kraj nie zastosował takiej strategii, nigdzie nie było takiej strategii. Tylko że u nich zachorowania miały miejsce wcześniej. To właśnie tego typu rady były niewłaściwymi radami, były radami, które miały zakłócić porządek walki z koronawirusem. Najpierw mówiliście o tym, że koperty mogą być zabójcze, mogą być śmiercionośne, chodzi o koperty do głosowania, by potem, chwilę później żądać otwierania całej gospodarki, natychmiast, ażeby potem jednak, jak już otworzyliśmy pewne sektory, mówić, że to za wcześnie, by chwilę później, na początku maja jednak znowu domagać się, żeby wybory były w trybie tradycyjnym, a gospodarka natychmiast otwarta. Gdzie tu jest konsekwencja? Nie ma konsekwencji w Platformie Obywatelskiej. Nie było konsekwencji w walce z kryzysem 12 lat temu - o tym jeszcze za chwilę powiem - i nie ma konsekwencji w waszym podejściu dzisiaj. Jest tylko próba zamieszania, jest liczenie na to, że ludzie mają krótką pamięć. Ale nie bójcie się, nie obawiajcie się, Polacy mają dobrą pamięć. A teraz, szanowni państwo, Wysoka Izbo, taki eksperyment dla ludzi o stalowych nerwach. Jak wyglądałoby zarządzanie pandemią w czasach koronawirusa na przykładzie świńskiej grypy w 2009 r. I kiedy w Polsce zachorowań było już ponad 130 tys., to był listopad 2009 r., rada ówczesnej pani minister Kopacz była taka: nic nie róbcie, cieszcie się wiosną - mniej więcej w ten sposób - a ówczesny premier Tusk mówił o tym, że to globalna histeria.

Tak reagowali wówczas przywódcy, osoby odpowiedzialne za służbę zdrowia.

pan Janusz Lewandowski powiedział wówczas w następujący sposób: na szczęście byliśmy odporni na wołanie ze strony gospodarki, żeby wdrożyć pakiety stymulacyjne, tak jak w innych krajach. Szanowni Państwo! Drodzy Przedsiębiorcy! Drodzy Pracownicy! Platforma Obywatelska na pewno byłaby odporna na wasze wołanie o pomoc, o tarczę, o pakiety stymulacyjne.

Nawet teraz, parę dni temu, parę lat temu powołany został chyba u was gabinet cieni.

Ale ja się nie dziwię, bo praktycznie przez poprzednie 8 lat to był taki gabinet cieni. Szanowni Państwo! Warto bardzo mocno podkreślić, co się działo w czasach, kiedy na świat spadł kryzys finansowy z lat 2008 i 2009.

Już zamknijmy oczy czy spuśćmy kurtynę miłosierdzia na to, że ponad 1 mld zł to nie jest zbyt dużo pieniędzy na rosnące gwałtownie wówczas bezrobocie.

Na ubóstwo, na bezrobotnych nie było wówczas pieniędzy.

Nie było pieniędzy na 500+, nie było pieniędzy na politykę rodzinną, nie było planu dla rodzin. Nie było planu dla rodzin wtedy, ale jest plan dla rodzin teraz. To jest taki plan, nazwijmy go umownie, Rabieja i Trzaskowskiego. To jest plan ataku na rodziny. To jest plan, który grozi polskim rodzinom. Mówimy bardzo wyraźnie, mówimy bardzo jednoznacznie, że podniesienie ręki na dzieci, na dzieci w polskich rodzinach jest niedopuszczalne, że granica pomiędzy rodziną a ideologią, waszą ideologią, waszymi eksperymentami ideologicznymi, musi być postawiona twardo. Jesteśmy gwarantem, że nie będzie ingerencji, że w całej Polsce nie będzie takiej ingerencji, jaka już odbywa się w niektórych miastach rządzonych przez Platformę Obywatelską. do tego, że dzieci będą chronione, chronione przed waszymi różnymi ideologicznymi eksperymentami, przed różnymi światopoglądowymi fanaberiami, bo dzieci są świętością.

Tymczasem w przypadku Platformy Obywatelskiej nie było żadnego działania, które mogłoby pomóc wówczas polskim rodzinom.

Skuteczność nie polega na tym, że ktoś was klepie po plecach czy ktoś się ustawi do dobrego zdjęcia, tylko na twardym negocjowaniu. Skutecznie wynegocjowaliśmy dodatkowe blisko 300 mld zł, [[Oklaski]] oprócz budżetu na kolejną perspektywę. Podkreślam: oprócz budżetu na kolejną perspektywę. Po co to robimy? Po to, żeby polscy pracownicy mogli spać spokojniej. Nie spokojnie, bo dzisiaj cały świat jest w ogromnym rozedrganiu, żyje pod ogromnym pręgierzem ryzyka. Musimy proponować rozwiązania w klimacie ogromnej niepewności i robimy to, ale robimy to po setkach wideokonferencji z przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, pracownikami, bo na tym polega realne rządzenie. Po to się idzie do polityki, żeby pomagać ludziom, żeby służyć ludziom, służyć Polsce.

Bo kiedy Komisja Europejska albo EBOR lub inne instytucje finansowe z całego świata mówią o tym, że Polska również w tym roku zostanie najmniej dotknięta w Unii Europejskiej pandemią koronawirusa od strony gospodarczej, to jest to najlepszy dowód na to, że nasze odważne działania, przeznaczenie przez nas miliardów złotych na pomoc, na ratowanie miejsc pracy, jest właściwą strategią. My - repolonizacja. My - przekazanie środków dla polskich przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy. To jest różnica między Platformą Obywatelską, partią wyprzedaży, a Prawem i Sprawiedliwością, partią, która dba o polski kapitał, o polskich przedsiębiorców, o polską własność. Zapytajcie firmę Black Red White, jak szybko dostała pieniądze na swoje konto na ratowanie miejsc pracy.

Otóż kiedy pan przewodniczący Budka tu czy tu rozmawiał z panem przewodniczącym Kosiniakiem, po cichu, nie wiedząc, że kamery słuchają, nagrywają, to było powiedziane, że: ta tarcza jest dobra, co nie? Dobra jest. Drodzy Rodacy! Tacy oni są: po cichu przyznają, że to jest. Tak jak Galileusz, prawda? Ale wiecie co? Dziękujemy wam bardzo za to.

Powtarzał to za Leszkiem Balcerowiczem, który mówi to ostatnio chyba co kwartał, a może nawet co miesiąc, już nie pamiętam. Ale nie przejmujcie się tym. Nie było wtedy katastrofy, nie będzie teraz. Tylko pozwólcie nam rządzić. Nie przeszkadzajcie.

Tutaj chcę powiedzieć o wielkim programie wielu inwestycji. I chcę powiedzieć, że w tym momencie chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi. Dziękuję, panie prezydencie. Bo to z inspiracji pana prezydenta Andrzeja Dudy, tak, właśnie z jego inspiracji, ale nie tylko. To również z jego planów, z jego wizji rozwoju zrodził się wielki program inwestycyjny.

A może plan Junckera?

Kolejna niekonsekwencja.

To jest miara skuteczności i umiejętności negocjacyjnych rządu Prawa i Sprawiedliwości. Owszem, drodzy państwo, nasze inwestycje nie zakładają modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Nasze inwestycje to realne inwestycje dla mikro-, małych, średnich i dużych firm, dla małych gmin, dla większych gmin, dla powiatów i dla dużych miast. Każdy z 380 powiatów doświadczy planu inwestycyjnego, który przygotowuje rząd Zjednoczonej Prawicy razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą.

Niektórym się to nie będzie podobało, tak jak Centralny Port Komunikacyjny. Wiem, że dla niektórych z was byłoby lepiej, żeby lotnisko było w Berlinie, rozumiem, natomiast my chcemy jako suwerenne państwo, państwo z ambicjami mieć tutaj Centralny Port Komunikacyjny, który przełamie jeszcze pozaborowy układ komunikacyjny.

To jest repatriacja kapitału, a nie wyprzedaż majątku, tak jak w waszych czasach. Wysoka Izbo! Te inwestycje to nie jest żadne albo-albo: albo szkoły, albo drogi. Oni tak mówią. To kolejna niekonsekwencja. Te inwestycje to inwestycje zarówno w szkoły i żłobki, jak również w drogi, mosty i koleje. Spytajcie swoich samorządowców, dlaczego proszą o tę pomoc. Bo wiedzą, że sami nie będą w stanie tego sfinansować. I my dajemy tę pomoc, również wielkim miastom, dajemy małym powiatom, bo nasz model rozwoju gospodarczego to model zrównoważony, taki, na jaki umówiliśmy się z Polakami.

Te pieniądze będą dostępne na szereg projektów. Przekonacie się państwo o tym w ciągu kilku najbliższych dni. To jest ważne, żeby każdy wiedział, że ma szansę na wyjście z tego błędnego koła koronawirusa, w którą wpadł cały świat. Dzisiaj rano przeczytałem, że w Meksyku zmarło w ciągu jednego dnia więcej osób niż w ciągu 3 miesięcy w Polsce. To bardzo smutne, bo każda śmierć jest ogromną tragedią, ale to jednocześnie pokazuje pewne miary, pewne porównania. Powinniście z odwagą, patrząc w lustro, przyznać, że nasze zarządzanie tym kryzysem zarówno od strony zdrowia, służby zdrowia, zdrowia publicznego, jak i od strony gospodarczej jest skuteczne. Teraz kilka zdań na temat polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej.

I dużo udało nam się rzeczywiście załatwić, i pierwszemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości, i kolejnym, którym miałem zaszczyt przewodzić.

I dlatego właśnie my, mając taką siłę, jaką mamy, blisko rok temu doprowadziliśmy do tego, że na najważniejszą funkcję w Unii Europejskiej nie został wybrany człowiek, który szkodził Polsce. Pokazaliśmy, co znaczą skuteczne negocjacje.

Was to oczywiście boli, bo to był wasz ogromny sojusznik, ale niestety właśnie na tym polega realizacja interesów polskich, a nie realizacja interesów za granicą. Jak jeździcie za granicę, to dbajcie o interesy polskie, a nie walczcie z rządem polskim, bo to wielki błąd. Ja, Wysoka Izbo, do dzisiaj czasami nie mogę uwierzyć, że prominentni działacze Platformy Obywatelskiej nie chcieli środków z Unii Europejskiej.

Albo były przewodniczący pan Grzegorz Schetyna, który w podobnym tonie wypowiadał się na te tematy. Szanowni Państwo! To jest strzał do własnej bramki, to są gole, które strzelacie społeczeństwu polskiemu. Możemy się spierać we własnym gronie, spierać na wizje, jeśli będzie taka wizja z waszej strony, jeśli będzie taki program, chętnie się pospieramy na programy, ale nie szkodźcie naszym interesom za granicą. My kształtujemy politykę międzynarodową w duchu pewnej refleksji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powiedział o tym, że jeżeli ktoś chce być wielkim narodem, być traktowany jako wielki naród, to musi chcieć nim być. I jeśli ktoś chce, żeby inne państwa miały do nas szacunek, to sam musi mieć szacunek do samego siebie. Szanujemy Polskę, szanujemy Polaków, szanujemy polskie interesy, nawet jeżeli walka jest na nierównym polu. Bo walka w Brukseli jest na trudnym polu, jest walka na trudnym ringu, nie do końca nasze boisko. Ale nie boimy się, walczymy skutecznie o interesy Polski właśnie po to, żeby móc Polakom powiedzieć: wywalczyliśmy maksymalnie to wszystko, co się dało, albo może nawet trochę więcej. Dzięki tej polityce.

Z budżetu państwa polskiego dzięki uszczelnieniu, dzięki uszczelnieniu podatków. Mam też prośbę do waszych samorządowców, którzy nie radzą sobie z dystrybucją środków. Drodzy państwo - do wszystkich szanownych posłów - sprawdzajcie w waszych samorządach, kto ile środków rozdystrybuował przekazanych przez budżet państwa. Dajemy je mikroprzedsiębiorcom na uratowanie ich biznesów, żeby przetrwali ten trudny Schumpeteriański dołek w szoku podażowym, szoku popytowym, który nastąpił. Ale niektóre samorządy sobie z tym nie radzą. Ciekawe, jak to jest, że zwykle nie radzą sobie z tym samorządy z Platformy Obywatelskiej. No, bardzo ciekawe. Ale one sobie często nie radzą z wieloma rzeczami. Jakoś tak zwykle przychodzą po pomoc do państwa polskiego, kiedy sobie nie radzą.

W latach przed 2015 r. Polska chorowała na taką chorobę, którą pan prezes Jarosław Kaczyński określił imposybilizmem. No, to jest dobrze opisana już w literaturze choroba, myślę, że nawet po waszej stronie jest zrozumienie: nic się Jak bezrobotny, to znaczy, że chyba leniwy, więc niech on sobie tam gdzieś z tego lenistwa sam wychodzi. Rolnicy, jak cierpią biedę, no to najwyraźniej nie radzą sobie po prostu, nie potrafią stosować odpowiednich instrumentów. Dzięki krokom, dzięki drodze, którą utorował pan prezydent Andrzej Duda 5 lat temu, zaczęliśmy przełamywać ten imposybilizm i później dzięki rządom, które nastały, rządom dobrej zmiany, pokazaliśmy, czym jest droga polskiej pracy, droga polskiej nadziei, przełamany imposybilizm. Ale dzisiaj grozi nam inna choroba, dzisiaj grozi nam choroba, którą nazwałbym immobilizmem. Immobilizm, czyli groźba pewnego klinczu, pewnego paraliżu, paraliżu pomiędzy poszczególnymi głównymi władzami w państwie. Ten immobilizm w czasie koronawirusa może być niezwykle groźny, bo może doprowadzić do marazmu, do paraliżu instytucji państwa. Przez to te instytucje nie będą mogły realizować tej wizji rozwoju, którą zaproponował pan prezydent Andrzej Duda i którą rząd Zjednoczonej Prawicy chce realizować. Wiecie co? Żeby zmienić Polskę, żeby wzmocnić Polskę, bo to ludzie widzą, że nasza polityka jest inna, jest polityką dla ludzi. A więc wkrótce Polacy rzeczywiście będą wybierać pomiędzy polityką takiej dojutrkowości, polityką marazmu, polityką immobilizmu a polityką nadziei na przyszłość, polityką inwestycji dużych i małych... 1 mln mieszkań.

A więc, aby tak było, abyśmy w pensjach, w wynagrodzeniach, w jakości wzrostu gospodarczego, w innowacyjności, w modernizacji państwa polskiego byli sprawni, byli skuteczni - po to wszystko potrzebne są rządy zgody, rządy jedności, jedności w państwie polskim... Blok Jedności Narodowej.

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Z tej mównicy równo 28 lat temu pan premier Jan Olszewski zadał znamienne pytanie: Czyja ma być Polska? Nie, nie tylko ono jest jeszcze dzisiaj aktualne. Co więcej, ono dzisiaj się rozstrzyga, ono rozstrzyga się właśnie w tym czasie. które chcą po kompradorsku wysługiwać się zagranicy, czy Polską wszystkich Polaków, nawet tych, którzy byli zapomniani, byli na marginesie procesu transformacji?

Czy Polska ma być krajem ambitnym, czy krajem, który sobie dryfuje gdzieś tam na falach oceanu? Czy Polska ma być aktorem, czy widzem w tej europejskiej, a może z czasem nawet światowej grze? Tak, my mamy właśnie takie ambicje. żeby Polska była państwem coraz więcej znaczącym na świecie. I te wybory dzisiaj się rozstrzygają. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Przez ostatnie 3 miesiące doświadczyliśmy kryzysu, jakiego wcześniej nie widzieliśmy przez 30 lat, co najmniej 30 lat. Ale warto również podkreślić, że te ostatnie 3 miesiące to także zagrożenie dla pewnych postępów, dla korzyści, które społeczeństwo polskie odniosło w ostatnich 5 i w ostatnich 30 latach, bo przecież Polska się rozwijała, rzecz jasna. To wielkie zagrożenie. I w tym wielkim zagrożeniu nie potrzebujemy tego awanturnictwa, pieniactwa i niezgody.

Potrzebujemy jedności i potrzebujemy spokoju, po to żeby przezwyciężyć te wszystkie patologie, które wokół się szerzą. całe zło, które jest do wyplenienia. Wysoka Izbo! Warto to podkreślić, że poradziliśmy sobie całkiem nieźle z pandemią koronawirusa. Radzimy sobie nieźle, coraz lepiej z kryzysem od strony gospodarczej.

Wysoka Izbo! I chciałbym na koniec powiedzieć, trochę tak jak Stanisław Barańczak mówił o tym, żeby spojrzeć prawdzie w oczy, bo prawda was boli. Spójrzmy w oczy Polsce i Polakom. mimo kryzysu, mimo tych wszystkich kłamstw, które padają z tamtej strony, my będziemy dalej prowadzić Polskę ku ambitnym celom. ku lepszemu podziałowi dóbr, ku Polsce sprawiedliwej. Będziemy to robić, dopóki starczy sił.

Dziękuję, panie premierze.

Proszę państwa, ogłoszę teraz przerwę do godz. 13.20.

Rozpatrzenie wniosku Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów. Przypominam, że zgodnie z art. 117 ust. 2 regulaminu Sejmu debata nad wnioskiem obejmuje wyłącznie zadawanie pytań prezesowi Rady Ministrów i jego odpowiedzi na pytania. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Zamykam listę osób zgłoszonych do pytań. Pierwszy pytanie zadaje pan poseł Waldemar Andzel, klub Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Borys Budka, klub Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Nie dziwię się. Mamy dość tych kłamstw, mamy dość tej obłudy. To, co pan premier przed chwilą powiedział, to była farsa, próba przykrycia nieudolności tego rządu. Dlaczego pan premier nie wspomniał o stadninie w Janowie? Dlaczego pan premier nie wspomniał o tym, jak jego rząd dał zarobić kumplom z banków, odkupując Bank Pekao od Włochów za 123 zł, a teraz akcja jest warta 54 zł? Zniszczyliście Alior Bank, jak zabraliście się za ten bank. Za co się nie zabierzecie, to zepsujecie. Raz jeszcze, panie premierze, mamy dość obłudy i kłamstwa. Dzisiaj, gdyby pan był człowiekiem honoru, za Szumowskiego, za Banasia podałby się pan do dymisji, a nie błagał o wotum zaufania, przebłagując pana prezesa, [[Dzwonek]] który zresztą.

Wysoka Izbo! Panie Premierze!

Im więcej pan mówi, tym bardziej każdy widzi, że to wszystko jest pic, nieprawda i oszustwo. Podam tylko dwa przykłady. Czy pan uważa, że to jest naprawa państwa, o której pan mówi, że w Gliwicach studenci, że w Katowicach studenci są przesłuchiwani przez prokuraturę i policję z udziałem Ordo Iuris? To jest ta naprawa państwa, że fundamentaliści przejmują państwo? Druga sprawa również jest ze Śląska. Pan jest posłem ze Śląska.

Pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, klub PSL-Kukiz15. To było jedno z najbardziej bezczelnych wystąpień w historii tej Izby. Pan wiele o historii, jak zawsze, ale to nie było historyczne wystąpienie, tylko histeryczne, ustawka pod Andrzeja Dudę. Wasze PO-PiS-owe wojny, podział Polski. Zamiast czytać „Die Welt”, niech pan zacznie czytać listy od polskich przedsiębiorców, którzy musieli zlikwidować działalność albo ją zawiesić, od 600 tys. pracowników, którzy od grudnia stracili pracę, [[Oklaski]] od rolników, którzy nie dostali suszowego, od rodziców dzieci chorych na choroby rzadkie, którzy nie mogą się doprosić o pomoc państwa. Niech pan nie słucha oklasków klakierów, tylko niech pan usłyszy rodziców, którzy pragną, żeby ich dzieci miały implanty. Tego nie słyszycie, na to jesteście głusi. O leczeniu. Was trzeba uleczyć z ciężkiej choroby nienawiści. Jesteście wektorem tej choroby. Roznosicie ją po całej Polsce. W tej wojnie czujecie się dobrze. Macie jeden program: zabić PiS, [[Wesołość na sali]] zabić Platformę.

Szanowny Panie Premierze! Pytanie bardzo konkretne: Czy prawdą jest, że w ramach walki z pandemią dokonano zakupu większej ilości jeszcze nowszych, jeszcze lepszych niszczarek, które przez to półrocze, które pan sobie kupuje dzisiejszym wotum zaufania, będą mogły zamortyzować się w urzędach centralnych? Konkretne pytanie. Chciałbym również wiedzieć, czy pański rząd śledzi statystykę, tragiczną statystykę zgonów z przyczyn innych niż jedynie słuszny i modny w tym sezonie koronawirus. Czy państwo liczycie tych wszystkich ludzi, którzy odeszli na tamten świat, ponieważ nie dopuściliście do łóżek obłożnie chorych, tak, owszem, nie dopuściliście ich bliskich, najbliższych? Przy najwyższym oddaniu personelu niższego szpitalnego. Pan poseł Paweł Rychlik, klub Prawo i Sprawiedliwości. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Ja klaskałem jako przede wszystkim wielunianin, w którym siedzibę ma główny, największy producent naczep - firma Wielton. Dzięki tarczy antykryzysowej, którą on wymyślił i która działa dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, główny chlebodawca miasta i ziemi wieluńskiej funkcjonuje. I dzięki temu zostały zachowane miejsca pracy. Dlatego chciałem zadać pytanie: Ile miejsc pracy zostało zachowanych, zabezpieczonych dzięki tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej? Pani poseł Katarzyna Lubnauer, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Atak paniki, histeria i bezsilność wyzierały z tej wypowiedzi pana premiera Morawieckiego. Czujecie, że za sprawą Szumowskiego grunt pali się wam pod nogami, czujecie spadające sondaże Dudy i rosnące Rafała Trzaskowskiego. Tak, Polacy są oburzeni kręceniem lodów z okazji pandemii. Polacy tracili dochody, a w tym czasie krewni i znajomi ministrów z PiS zdobywali zamówienia na przepłacone maseczki, przyłbice i testy. Plan: rodzina Szumowskich na swoim. Gigantyczny konflikt interesów: minister, jego żona i brat, konflikt na setki milionów. Tak, zakłamujecie rzeczywistość, cieszycie się statystykami, ale mamy dość tej ściemy.

Pani poseł Monika Falej, klub Lewicy. Panie Marszałku! Panie Premierze! Krytykując pana rząd, niemal wszyscy pomijają pana, atakując tak naprawdę pana Kaczyńskiego, oskarżając go o nieudolność rządów PiS, i to jego postrzegają jako lidera tej ratalnej ekipy, zapewne słusznie. Dziś może pan jednak przejść do historii jako polityk, który bierze odpowiedzialność za rząd, którym kieruje. Czy poczuwa się pan do odpowiedzialności za afery i nadużycia w niemal w każdym ministerstwie, za nieudolność pana Sasina, za rodzinę na swoim pana Szumowskiego, chaos w wymiarze sprawiedliwości pana Ziobry, który dopuszcza fundamentalistów z Ordo Iuris do przesłuchiwania studentów? Jeśli rzeczywiście ma pan jakikolwiek wpływ na własny rząd, to może pan to dziś udowodnić - samemu podając się do dymisji. Będzie to najlepsze uczczenie rocznicy wyborów, wolnych wyborów, wolnej Polski, którą właśnie zniewalacie. Poseł Czesław Siekierski, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie Premierze! Dlaczego pana wystąpienie miało tak konfrontacyjny charakter? Zaczął pan mówić o pieniaczach opozycji, żeby za chwilę nawoływać do jedności. Jak się ma jedno do drugiego? Co pan chciał uzyskać? Czemu to ma służyć?

Mówi pan o dobrobycie. Jakie wskaźniki określają ten dobrobyt? Czy to, że dzieci nie mają komputerów, żeby móc zdalnie się uczyć? Mówi pan o polityce zagranicznej. Polska jest osamotniona w polityce zagranicznej, jesteśmy samotni. Gdzie mamy dobre relacje, z kim? Czy w Unii Europejskiej? Czy poprawiły się relacje z Rosją?

W swoim wystąpieniu wielokrotnie zachwalał pan stymulowanie gospodarki za pomocą publicznych pieniędzy. Wiem, że już o to pytałem, ale będę pytał i uświadamiał do skutku: Czy wie pan, skąd się biorą publiczne pieniądze? Publiczne pieniądze biorą się stąd, że rząd zabiera je najpierw z gospodarki, więc pomysł, że można stymulować gospodarkę za pomocą pieniędzy wyjętych z tej gospodarki, to jest taki sam pomysł jak to, że można się podnieść za włosy nad ziemię. To jest ta idea, tylko bardziej skomplikowana. Bo działacie według zasady, że jeśli coś nie działa, to rozbuduj i trudniej będzie zauważyć, że to nie działa. Jeśli coś nie działa w małej skali, to nie zadziała też w dużej skali. Drugie pytanie: Dlaczego pan o epidemii mówi w czasie przeszłym? Bo dane na to nie wskazują. Pan powołał się na przykłady innych krajów. U nas trzyma się cały czas na wysokim poziomie. Pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość.

Wysoka Izbo! Panie premierze, kilka dni temu kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta powiedział, że należy zawiesić, zamrozić, de facto zlikwidować istotne inwestycje prorozwojowe dla Polski.

Wiemy doskonale, że ta inwestycja to również tzw. dziewięć szprych dla kolei szybkich prędkości. Gdyby pójść tokiem myślenia pana Trzaskowskiego, to również miejscowości, gdzie ta kolej miałaby przebiegać, stracą na tym nie tylko miejsca pracy, ale również możliwość szybkiej komunikacji z wieloma miejscami w Polsce.

Panie Marszałku!

Nic, nic z takich rzeczy. Za to usłyszeliśmy kilkanaście razy: Platforma Obywatelska, Borys Budka, Donald Tusk, nawet słyszeliśmy nazwisko Rabiej, Balcerowicz i kilkanaście razy nazwisko Trzaskowski.

Czasy kryzysu to są zawsze czasy próby. Poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska, klub Lewicy.

Chwalił się pan wieloma rzeczami. Na szczęście nie pochwalił się pan tym, i słusznie, co robi minister Ardanowski. A robi on wszystko, żeby nikt nie mógł z rąk oprawców ratować maltretowanych zwierząt, zwierząt głodzonych, którym łańcuchy wrastają w szyje, które miesiącami stoją we własnych odchodach. Niestety nie udało się nawet pana koledze, najważniejszemu posłowi, Kaczyńskiemu powstrzymać tego łajdackiego interesu.

Wysoka Izbo! Panie Premierze! W których więzieniach siedzą osądzone osoby z mafii VAT-owskiej? Kto mieszka w tych 100 tys. mieszkań+? Kto jeździ tym milionem samochodów elektrycznych? Kto oddycha tym czystym powietrzem i w jakich miejscowościach? A może, panie premierze, odpowie mi pan na pytanie: Dokąd pływają te promy ze Szczecina? Gdzie one są, panie premierze? Bo jeżeli mówimy o wotum zaufania, to musimy też mówić o tym, co nam się nie udało. Panie premierze, takich słów nie uzyskałem od pana.

Pan poseł Jakub Kulesza, koło Konfederacji. Panie Premierze! Ciężko się odnieść do tej całej serenady manipulacji, kłamstw, pustosłowia. W dużej mierze skupił pan się na krytyce Platformy Obywatelskiej, i jest to, że Platforma, wzorem innych krajów, nie zmarnowała milionów złotych na szczepionkę, która była niepotrzebna. Państwo by zmarnowali, tak jak zmarnowali państwo 68 mln zł na druk kart wyborczych.

Państwo się boją tego, że obywatele zauważą, że niczym się państwo od Platformy nie różnią. 34 nowe podatki lub podniesione podatki - to jest właśnie clou państwa rządów.

Panie Premierze! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić się do pana premiera w ramach odpowiedzi na pytania o rozszerzenie informacji, dlatego że skupił się pan premier właściwie na sprawach krajowych, na tym, co się u nas dzieje, a przecież w tym czasie, w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, uzyskaliśmy bardzo duże sukcesy w sprawach międzynarodowych. Można wspomnieć choćby o takich rzeczach, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o wschodnią granicę, o ochronę naszej suwerenności, np. doprowadzenie do tego, że będzie synchronizacja energetyczna Litwy, Łotwy i Estonii dzięki działaniom Polaków, dzięki temu, że zostało w czerwcu 2019 r. podpisane porozumienie z tymi państwami. Ale przecież mamy jeszcze sukcesy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i szereg sukcesów, które uzyskaliśmy współpracując właśnie z Komisją Europejską i szerzej, także ze Stanami Zjednoczonymi.

Ja o formie, bo jednak estetyka dla naszego narodu jest rzeczą ważną. Panie Premierze! Nie ma obydwu panów, ale obydwaj panowie coraz głośniej krzyczycie i coraz szybciej mówicie. Chciałam zaapelować słowami poety, bo źle się kojarzy krzyk i szybkie mówienie, jako historyk, panie premierze, pan o tym wie: Wolno bardzo do nas mów, premierze, słodko bardzo do nas mów, premierze, nie krzycz, bo trzeba cenę swoją znać, premierze, trzeba trzeźwo życie brać, premierze, trzeba wyczuć, kiedy w szatni płaszcz pozostał przedostatni, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Ma pan szansę. Ja rozumiem, że to jest desperacja, bo wasze dni się kończą, ale ważne jest dla Polaków.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeden ze sztandarowych projektów - „Mieszkanie+” A jaka jest prawda? 867 mieszkań oddanych, 1900 w budowie. Pytam zatem: Ile spółek celowych powołał Krajowy Zasób Nieruchomości?

Bo dzisiaj wydaje się, panie premierze, że 100 tys. to wydaje decyzji i opóźnia o miesiąc sprzedaż nieruchomości przez różne podmioty, a nie kupuje tych nieruchomości. Ile z tych tysięcy decyzji, które wydaje na 1000 m na zakup lokalu, jest pozytywnych, a więc skorzystał z prawa pierwokupu? Ile nieruchomości posiada w swoich zasobach?

Panie Premierze! Trzeba mieć szacunek dla siebie.

Najczęściej słyszałem słowo „kłamca”, które się tutaj pojawiało, i to mnie trochę martwi. Obserwowałem też oklaski z sali. Pan poseł Artur Dziambor, koło Konfederacji. Jakoś nie widzę. Tymczasem pan poseł Arkadiusz Mularczyk, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ostatnie miesiące były niewątpliwie wstrząsem dla polskiego społeczeństwa, ale też społeczeństwa Europy i świata.

Udało się skutecznie walczyć, skutecznie leczyć te wszystkie osoby, które zachorowały na COVID-19. Także na tej Izbie przecież są parlamentarzyści czy członkowie rządu, samorządowcy, którzy korzystali z usług służby zdrowia. I niewątpliwie ta pomoc była wskazana i była skuteczna. Mam pytanie w związku z powyższym. Dziękuję bardzo. Koło Konfederacja.

Czy mamy połączenie z panem posłem? Pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! No to ja pana pytam: Jakiej skuteczności? Załogi wrocławskiego komisariatu, gdzie miał nieszczęście trafić Igor Stachowiaka? A może skuteczności w ściąganiu emerytom rzekomych zaległości w płaceniu abonamentu z tej trzynastej emerytury, którą pan im dał? Zabrali całą trzynastą, nawet zabierają już taką normalną. Więc jeżeli pan mówi o skuteczności, panie premierze, to proponuję odnieść to do siebie bezpośrednio. Otóż urządził pan nam tutaj bardzo piękny miniwiec wyborczy Andrzeja Dudy i wie pan co? Naprawdę jak tak będzie dalej, to na pewno przegracie niezależnie od tego, że i tak wygra Rafał Trzaskowski. Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Rząd PiS bardzo nie lubi samorządów. was, że władzę w terenie ma ktoś, kogo nie kontrolujecie. Samorządy dawały radę, bo Polską lokalną rządzą dobrzy gospodarze. Na walkę z pandemią samorządy z własnych środków dały 2 mld zł. Do końca roku kolejne 2 mld zł samorządy stracą z powodu mniejszych wpływów do budżetu, a to dane tylko z dużych miast. Oznacza to mniejsze nakłady na szkoły, na przedszkola, na komunikację publiczną. Stracą na tym ludzie, a nie prezydenci miast, których nie znosicie. Stąd moje pytanie: Co rząd zamierza zrobić, aby uratować samorządy przed budżetowymi skutkami pandemii? Czy poprzecie ustawę Lewicy o świadczeniu rekompensującym dla samorządów? Panie premierze, dość jazdy na gapę kosztem samorządów i ich mieszkańców.

Wysoka Izbo! Skoro pan premier mówi o skuteczności, to jestem bardzo ciekawy, dlaczego nie wspomniał o narodowym holdingu spożywczym.

O tym też pan premier w ramach skuteczności nie wspomniał. A może pan premier pochwaliłby się, dlaczego rokrocznie kilkadziesiąt miliardów złotych wynosi zadłużenie naszych szpitali? Dlaczego nie wspomniał pan o tym, że w ostatnim czasie, kiedy PiS rządzi, zniknęło z mapy polskich szpitali kilkadziesiąt oddziałów zakaźnych?

Miarą waszej skuteczności jest wjazd autem na cmentarz, kiedy on jest zamknięty.

Panie Premierze! To, że w Polsce panuje chaos, to wiemy, ale teraz mamy wielki atak paniki. Jak inaczej wytłumaczyć dzisiejsze wotum zaufania dla pana premiera? Myślałam, że pan premier ma nam coś do powiedzenia, że opowie nam o tym, jakie ma plany, pochwali się zasługami, a to był atak na Platformę, na koalicję, na naszych polityków. O tym, co wy zrobiliście, nie było ani słowa.

Boicie się prawdy. Tak, apelowałam o testy. Uważam, że tych testów było za mało, bo tam, gdzie są robione testy, wiemy naprawdę, ile osób jest zarażonych i bezobjawowo przechodzi tę chorobę. Nawet wyborów nie potrafiliście przeprowadzić i dobrze zorganizować. Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub Lewicy. Panie Premierze! Okazuje się, że dzięki panu prezydentowi Dudzie mamy te wszystkie wielkie sukcesy, o których pan premier mówił. Ewidentnie jest to jakiś element kampanii wyborczej. Zupełnie bez sensu, że na tej sali w taki sposób to robimy, ale to jest wasza odpowiedzialność, pewnie w wyborach za to odpowiedzialność poniesiecie. Natomiast moje pytanie jest konkretne. Co z Polską Żeglugą Morską, która notuje dziesiątki milionów strat w ostatnim czasie? Nic w tej sprawie do tej pory nie zrobiliście. Pan poseł Artur Dziambor. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Pan premier Morawiecki zaserwował nam tutaj przemówienie, które momentami niestety wyglądało tak, jakby pan premier żył jeszcze w poprzednim ustroju. Mówienie do opozycji, że ona nie powinna zabierać głosu, nie powinna przeszkadzać, jeżeli nie ma możliwości wpłynięcia na wynik, jest troszkę słabe i powinno zostać odnotowane przez wyborców, przez wszystkich Polaków. Natomiast inna sprawa jest taka, że pan premier bardzo chętnie chwali się sukcesami, ale nie mówi o konsekwencjach. Mowa była o tym, jak to wzrosły zarobki Polaków. Niestety powiedziane zostało znowu to, że Polacy coraz więcej zarabiają, natomiast nie powinno umknąć, że przy okazji więcej płacą. Wielokrotnie czytaliśmy taki przykład z zapiekanką, która dzisiaj kosztuje 15 zł przy najniższej krajowej wynoszącej 2600, a przy 4 tys., które było zapowiadane przez Jarosława Kaczyńskiego, kosztowałaby trochę więcej.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Premierze! Za obszar rolnictwa i obszarów wiejskich, panie premierze, w pańskim rządzie odpowiedzialność konstytucyjną ponosi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Obraził on w nieodległym czasie nauczycieli, odsyłając ich do zbioru truskawek. Widzimy, jak radzi sobie jeśli chodzi o nadzór nad stadniną koni w Janowie Podlaskim, natomiast całkowicie zaniedbuje swoje powinności i zobowiązania, które ogłosił, chociażby jeśli chodzi o rolników w temacie: wypłata świadczeń suszowych. Mamy początek czerwca 2020 r. i wielu rolników z Wielkopolski, z której pochodzę, i w całym kraju tych świadczeń suszowych do dzisiaj nie zauważyło. Jak to jest, panie premierze? Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke.

nadal będzie przewidziane wsparcie dla ośrodków regionalnych i mniejszych miejscowości, po to żeby dawać im szanse rozwojowe? Przykładem tego jest np. inwestycja w Radomiu w lotnisko komplementarne dla lotniska Okęcie. Mam nadzieję, że rząd będzie nadal prezentował ten sposób widzenia: pozbawiony kompleksów i takiego wyłącznie wielkomiejskiego spojrzenia, a dający szansę rozwoju mniejszym ośrodkom. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Spróbujemy się połączyć. Jestem połączony. Chciałbym zacząć od pytania retorycznego: Dlaczego rząd widzi tylko lewicową opozycję, a nie widzi prawicowej? Dlatego że opozycja mówi to samo, co mówi rząd, niczym się od niego nie różni.

Wysoka Izbo!

Jest pan premierem, ale jest pan także posłem wybranym na Śląsku, posłem z Katowic, a to Śląsk jest niemal codziennie wytykany przez was palcami, kiedy mówicie: epidemia się skończyła, tylko ten Śląsk. To Ślązakom, mieszkańcom województwa, odmawia się wynajmu kwater, przebija się opony. Jak będą traktowane, kiedy stygmatyzowany jest Śląsk, kiedy pana posłanka z PiS-u przy mnie zakłada maseczkę, mówiąc: pani jest Śląska, to zakładam maseczkę?

Pani poseł Karolina Pawliczak, klub Lewicy. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mamy tutaj pokaz jakiejś bufonady w wykonaniu premiera. To, o czym pan mówi, to wierutne kłamstwa. Jest pan premierem na papierze, wyjętym z rzeczywistości. Opowiada pan bajki. Proszę wyjść na ulicę i zobaczyć, jak Polki i Polacy tracą pracę i upadają walczące z codziennością firmy. To jest życie, panie premierze, to rzeczywistość - nie taka, jak pan ją przedstawia. Siedzi pan w swoim wygodnym gabinecie pod sufitem, bo tyle ma pan spraw zamiecionych pod dywan. Zatem moje pytanie: Kto odpowiada za błędne decyzje wydania kart wyborczych za 70 mln zł? To jest szczyt bufonady i hipokryzji. Kiedy wreszcie poznamy prawdę dotyczącą rodziny państwa Szumowskich? Co z ujawnieniem przez pana i przez pana żonę majątku? Przecież obiecał pan to Polkom i Polakom.

Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Chciałem zapytać, dlaczego pan i pański rząd blokujecie polskim rolnikom dostęp do unijnych pieniędzy.

Ponad 30 mld leży w bankach w Brukseli. Pan prezydent na spotkaniu z rolnikami mówił, że rolnicy chcą modernizować, inwestować, rozwijać swoje gospodarstwa. Czy panu nie wstyd? Pan minister Gróbarczyk oferował nam poszerzanie i pogłębianie koryt rzecznych. Pani poseł Barbara Bartuś, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Tak boicie się tego, że powołujemy się na pana prezydenta Andrzeja Dudę, ale tak, to właśnie od wygranej pana prezydenta Andrzeja Dudy i tego, co powiedział w swojej kampanii wyborczej, zaczęła się dobra zmiana, zaczęło się od przywrócenia wieku emerytalnego, który państwo podnieśliście. Po wygranych Andrzeja Dudy przyszły kolejne programy, m.in. program 500+, który można było dzięki prezydentowi zrealizować. Dzisiaj zadzwoniłam do mojej córki, matki trójki dzieci mieszkającej na osiedlu, gdzie takich rodzin jak jej jest dużo, i pytam: Beatko, o co mam zapytać pana premiera, bo są pytania? Usłyszałam: proszę podziękować za pieniądze, które idą na inwestycje drogowe. A państwo kłamiecie i. Dziękuję, pani poseł. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Premierze! Wysoka Izbo! Ja się bardzo cieszę, że rząd podejmuje tematy związane np. z transportem zbiorowym, rozpoczęty jest temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, lecz dlaczego to wszystko powstaje ponad głowami mieszkańców Baranowa, Łodzi, Warszawy? Dlaczego to wszystko nie jest konsultowane? Dlaczego program „Kolej+” jest tylko wirtualnym, propagandowym projektem tylko na potrzeby kampanii? Szanowni Państwo! Ile mieszkań powstało z programu „Mieszkanie+” Ile samochodów z miliona elektrycznych powstało? Dlaczego państwo, zamiast rządzić, walczycie z ostrym cieniem mgły? Dlaczego po prostu zajmujecie się propagandą w telewizji, zamiast po prostu zajmować się problemami Polek i Polaków, które są naprawdę ważne? To jest trudny rok, ekstremalnie trudny, jest pandemia, susza, kryzys ekonomiczny, a państwo bawicie się po prostu w jakieś wojenki. To jest wszystko skandal.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! To jest dobry dzień dla Polski, bo to jest dzień, w którym widać, że wam spada, że spada PiS-owi, [[Oklaski]] że spada Dudzie, że mimo że TVP robi wam cały czas kampanię wyborczą, to wam ciągle w sondażach spada. Opowiadacie jakieś farmazony o wielkich inwestycjach, a nie znacie życia, panie premierze, pan życia nie zna. Czy pan wie, że 14 mln ludzi w Polsce nie ma dostępu do transportu publicznego? Czy pan wie, że 45% ludzi do 34. roku życia mieszka z rodzicami, bo nie stać ich na mieszkanie? Pan wie coś o tym? Pani poseł Małgorzata Tracz, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciał nas pan dzisiaj przekonać, jak świetnie pana rząd radzi sobie z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym. Chciał nas pan przekonać, że w środku pola wybuduje nową metropolię, a przekopem Mierzei Wiślanej odmieni gospodarkę regionu. Panie Premierze! Czas skończyć z tym mydleniem oczu. Pana rząd nie szanuje prawa polskiego i europejskiego, marnotrawi publiczne pieniądze w imię własnych politycznych celów lub prywatnych interesów kacyków. Nie umiecie sobie dalej poradzić z suszą. Wasza metoda walki z ASF poniosła totalną klęskę. Pana rząd z dumą wyłączył Polskę z europejskiego zielonego ładu, pozbawiając nas szansy na udział w prawdziwej tarczy antykryzysowej - dla zielonych miejsc pracy. Pani poseł Katarzyna Ueberhan, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Dzisiaj wszyscy zastanawiamy się, co jest przyczyną tego wniosku o wotum zaufania dla rządu: czy jest to próba przykrycia afery Szumowskiego, afery Sasina. A właśnie, a propos kart wyborczych: zgodnie z odpowiedzią szefa kancelarii premiera koszty wydruku tych kart ponosi resort spraw wewnętrznych i administracji, a w praktyce faktury na 68 mln, jak dowiadujemy się z doniesień medialnych, zostały wystawione na Pocztę Polską. Poczta Polska opłaciła już 24 mln z tej kwoty. Moje pytanie: Co zrobił rząd, by zabezpieczyć Pocztę Polską, by zabezpieczyć środki na te wydatki?

Pan poseł Marek Suski, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!

Takie były wasze rządy. Szanowny Panie Premierze! Chciałem zapytać, czy możliwe byłoby obniżenie wieku emerytalnego podniesionego przez Platformę i PSL, czy możliwe byłoby znalezienie pieniędzy, których za ich czasów nie było, na program 500+, czy możliwe byłoby sprawne wprowadzenie tarczy antykryzysowej, gdyby nie dobra współpraca rządu z prezydentem Andrzejem Dudą. Dziękuję bardzo.

Szeregowy Pośle Kaczyński! Panie Marszałku! Panie Premierze! Jak kraj potrzebuje maseczek, to wiecie, że trzeba zwrócić się do instruktora narciarstwa. SMS i powstaje wianuszek zaprzyjaźnionych firm. Tak działa państwowa mafia, nawet podczas pandemii: cicho, sprawnie i niestety bardzo drogo dla podatnika. Wiadomo, że jak ktoś szuka roboty, nie ma kwalifikacji, ale należy do PiS-u, to spółki Skarbu Państwa stoją przed nim otworem, byle tylko umiał się przeżegnać. Przyznajcie: jesteście bezradni wobec kryzysu, bo was ten kryzys po prostu nie dotyczy. Opływacie w dostatki, a obywatele bez pomocy mądrego rządu cierpią. Prosi pan o zaufanie, ale podczas kryzysu, zamiast zjednoczyć naród, to go dzielicie. Kiedy ujawnicie majątki żon? Wasz ból jest lepszy niż mój. Niszczycie sądy, bo chcecie pozostać bezkarnymi. Blokujecie informację.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Brazylia, Rumunia, Szkocja, Izrael, Holandia, Ukraina, Nowa Zelandia, Ekwador, Ruanda i Bahamy - w tych wszystkich krajach ministrowie zdrowia zostali zdymisjonowani lub w poczuciu honoru podali się do dymisji, m.in. za sprowadzenie maseczek, które nie spełniały certyfikatów, czy złamanie zasad dystansu społecznego. W żadnych z tych krajów nie było przypadku kontraktu rządowego dla zaprzyjaźnionego instruktora narciarstwa.

Moje pytanie brzmi: Kiedy i czy rząd zamierza wprowadzić w swoich szeregach program honor+? Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie premierze, dlaczego jest pan tak nieudolny? Dlaczego nie radzi pan sobie, trwoniąc pieniądze podatników, z kuriozum, którym jest podkomisja Antoniego Macierewicza, grupa, której jedynym osiągnięciem było wysadzenie w powietrze blaszanego garażu i zepsucie ostatniego sprawnego tupolewa? Dlaczego miliony podatków zamiast na pomoc przedsiębiorcom idą na to bezsensowne działanie? Panie Premierze! Minister obrony narodowej rozkłada bezradnie ręce. Dlaczego? Ale Polacy mają dość i słusznie się tego boicie.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Pan prezydent, widzę, już poszedł. Chciałam wziąć udział w tym wiecu wyborczym i pochwalić rząd za 4 już lata niedziałania programu „Mieszkanie+” Dziękuję w imieniu połowy młodych ludzi w Polsce, którzy nadal mieszkają z rodzicami, za te 2 mln obiecanych i nieistniejących mieszkań. W imieniu drugiej połowy dziękuję za pętlę kredytową, którą mają na szyi, bo pan prezydent, nieobecny już, obiecał frankowiczom pomoc już 5 lat temu, ale swoich obietnic niestety nie dotrzymał.

Dziękuję, bo to pokazuje wasze priorytety. Macie ludzi, macie zasoby, macie nawet dobre pomysły, ale wolicie niestety robić własną rodzinę na swoim. Może też: panie prezesie, bo może pan prezes wysłucha, co się dzieje w ministerstwie rolnictwa. Od jesieni problemy na wsi narastają. Pozwoli pan premier, że przeczytam. 3% PKB na rolnictwo z budżetu krajowego. To podstawowa obietnica, której pan nie zrealizował. Średnia unijna: 50%. Upadek gospodarstw rodzinnych. To wy tak dbacie o gospodarstwa rodzinne. Zniknęło 100 tys. stad trzody chlewnej, głównie przydomowych. 40% rolników nie dostało odszkodowania za zlikwidowanie trzody chlewnej. Panie premierze, czy pan tam był? Bo ja tam byłam. Pan minister kłamie. Poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Szanowny panie premierze, czy pana rząd nie ma własnych osiągnięć, że musi pan 80% swojego wystąpienia poświęcać poprzednikom? A przecież tym poprzednikom pan doradzał.

Był na tej sali pan prezydent. Szkoda, że go nie ma. Z honorem go tutaj powitaliśmy. Z honorem byśmy go pożegnali, ale byśmy też zapytali: Panie prezydencie, gdzie są pańskie obietnice wyborcze? Mówił o nich pan poseł Suski. Może pan, panie premierze, rozwinie tę tezę i powie polskim rolnikom, gdzie jest zrównanie dopłat dla polskich rolników. Ja bym chciał. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Wysoka Izbo! Panie premierze, tymi krzykami i jarmarcznym dowcipem degraduje pan urząd premiera. Też z bardzo dużą uwagą czekałam na ten wielki sukces, jakim są prace podkomisji Antoniego Macierewicza. Na własną rękę próbowałam się dowiedzieć, jaki jest wynik tych prac, ale tajemnicza pani Zofia przekazała mi informację, że raportu mi nie pokaże, bo go po prostu nie ma. Ministerstwo Obrony Narodowej na pytanie, czy wiecie państwo, na co Antoni Macierewicz wydaje te ponad 2 mln rocznie, znacząco milczało. A więc nie sądzę, żeby pan do swoich sukcesów mógł zapisać nawet informacje na temat tego, na co Antoni Macierewicz wydaje publiczne w końcu pieniądze. Pani poseł Magdalena Biejat, klub Lewicy. Panie Premierze! Chwali się pan dziś z tej mównicy, jak to uważnie pan nadstawia ucha i wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym. Mam więc pytanie, kto panu szepcze do tego ucha, bo na pewno nie słucha pan głosu polskich obywateli, pracowników i pracowniczek, zwykłych ludzi i ich rodzin. Lewica ten głos przekazywała w postaci poprawek do kolejnych tarcz. Ile ich przyjęliście? W czasie 3 miesięcy kryzysu pan i pana gabinet zostawiacie zwykłych ludzi bez środków do życia, ze zmniejszonymi o połowę pensjami, na przymusowych urlopach, bez praw pracowniczych. W tym samym czasie przekazuje pan w ramach tarczy 70 mld rynkowi finansowemu. Na razie, jak widać, jedyne głosy, w jakie się pan wsłuchuje, to finansiści, banki i największe korporacje. Dla nich i dla pana kolegów bankierów, a nawet kolegów pana kolegów ministrów, pieniędzy nie brakuje. Brakuje ich za to zwykłym Polakom. Pan premier chce, byśmy przestali jako opozycja zadawać niewygodne pytania i nie przeszkadzali w wykuwaniu nowego ładu. Ja jednak zapytam: Dlaczego wymienia pan w swoim przemówieniu wielkie firmy, a ani razu nie wspomniał pan o bezrobotnych? Pan poseł Robert Kropiwnicki, klub Koalicja Obywatelska. Zastanawialiśmy się dzisiaj przez chwilę, po co to wotum, skąd ta nagła inicjatywa. No i teraz już wiemy: bo macie pożar w bunkrze. Pali się u was. No wszystko się wali. Ludzie się dowiedzieli, jaka jest prawda, i strach was obleciał. Sprawa się rypła. Ludzie widzą, że król został nagi, że po prostu zbankrutowaliście jako środowisko, że wasze kłamstwa zostały obnażone, bo wszystkie afery: Szumowskiego, Banasia, Kaczyńskiego, GetBacku, SKOK-ów i wielu innych - wszystko to jest niewyjaśnione. Prokuratura leży. Sądownictwo leży. Gdzie są te mieszkania? Naprawdę dziesiątki rzeczy obiecaliście i to wszystko zostało niezrobione. Banaś... ...bo wy zajmujecie się rodziną na swoim: urządzacie swoje siostry, wujków, ciotki, pociotki, bo to jest dla was najważniejsze, bo tak postrzegacie państwo. Powinniście odejść.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Moje pytanie będzie dotyczyć problemu umów śmieciowych, które raz wpuszczone do polskich przepisów regulujących zatrudnienie od lat, od lat przyczyniają się do pozbawiania milionów ludzi praw pracowniczych, tym samym systematycznie osłabiają polski Kodeks pracy, tworząc w nim kolejne wyłomy. Obiecywaliście zrobić porządek z umowami śmieciowymi, ale przypominam, że porządek miał polegać na ich usunięciu, a nie przejściu nad tym problemem do porządku dziennego. Efektem zaniedbań pańskiego rządu są dramaty polskich rodzin, Polek i Polaków, którzy z dnia na dzień stracili pracę bez okresu wypowiedzenia, bez odpraw, a często też bez możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych czy świadczeń z rządowej pomocy antykryzysowej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie przykryjecie afery Szumowskiego wnioskiem o wotum zaufania. Dziś Polska zobaczyła ten strach, strach przed utratą władzy. Szanowni Państwo! Kiedy i gdzie powstał ten szatański plan potraktowania pandemii komercyjnie? Kupilibyśmy maseczki nawet od diabła - mówił pan minister Szumowski. Tak, ten diabeł miał kask, gogle i narty. Szanowni Państwo! Kupuje za 137 tys. w hurtowni w Rzeszowie 7 tys. przyłbic, jedzie do Ministerstwa Zdrowia, sprzedaje za 340 tys. Ile zarabia? 200 tys.

Szanowny Panie Premierze! Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości w końcu weźmie się na serio za ochronę zdrowia? Ale nie tak, jak do tej pory. Od tego, że minister Szumowski klaszcze, a pan prezydent rapuje, nie zwiększają się nakłady na ochronę zdrowia. Przyjęliście ustawę, 6% PKB, i zapisaliście tam fałszywy sposób obliczeń. Liczycie PKB w stosunku do 2 lat wstecz, po to żeby oszukać pracowników ochrony zdrowia, ale też obywateli i obywatelki. Pytam się: Kiedy poprzecie ustawę Lewicy podnoszącą nakłady na ochronę zdrowia? Ale tak, jak trzeba, tak, jak jest liczone we wszystkich krajach europejskich. Nie oszukujecie opozycji, oszukujecie obywateli i tych, którym trzeba dzisiaj dziękować za całą pracę, którą wykonali w walce z pandemią, bo to nie jest wielki sukces Szumowskiego. To jest ogromna praca tysięcy pracowników ochrony zdrowia, od salowych przez lekarzy, przez pielęgniarki, którzy za psi grosz pracują, bo nie potraficie im zapłacić za tę pracę porządnie. Poseł Maria Małgorzata Janyska, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Farsa, którą pan dzisiaj odstawił w Sejmie, odbiła się szerokim echem w Polsce i Polacy pytają, czy nie jest panu wstyd, bo im jest wstyd, że mają premiera zakłamanego i aroganckiego. Na dowód przytoczę kilka wypowiedzi, nie da się oczywiście wszystkich: W trakcie przemówienia Morawieckiego wyłączyłam telewizor. Nie dało się tych oszczerstw słuchać. Słucham tego bełkotu i nie rozumiem. I teraz najlepsze, proszę państwa, na koniec, i prawdziwe, bo to był motyw tego dzisiejszego wotum: Trzaskowski jest nie do zatrzymania. Pozostał im paniczny strach. Polacy mówią: mamy dość. A przy okazji, panie premierze, sprowadzając pana z orbity kosmicznej na Ziemię. chcę zapytać: Gdzie jest obwodnica Piły, Ujścia, Obornik, gdzie jest „Kolej+”, gdzie są mosty+, gdzie są przystanki autobusowe i dowozy na wieś? Dzień dobry, panie premierze. Na początek gratulacje. Bardzo ładna PR-owska ustawka: pan mówi przez godzinę, my mówimy przez minutę, miejsca na poważną dyskusję nie ma. Udało się panu znowu uciec przed poważną dyskusją. Gratuluję. Ale tak czy inaczej chciałbym panu zadać proste pytanie. Bo mówił pan o tym, jak pan sobie świetnie radzi, walcząc z kryzysem, tylko nie wspomniał pan o tym czyim kosztem. Więc chciałbym, żeby pan powiedział Polkom i Polakom, ilu milionom pracowników już obniżono pensje i ilu pracownikom jeszcze planujecie państwo pensje obniżyć i ilu spośród nich w przyszłym roku wpadnie w ubóstwo. Bo to właśnie robicie. kosztem pracowników, dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy robił pan to ręka w rękę z Donaldem Tuskiem jako jego doradca. Czekam na odpowiedzi na te pytania, bo bała się na nie odpowiedzieć pani Maląg, bała się na nie odpowiedzieć pani Emilewicz i mnie, i związkom zawodowym, więc może pan zdobędzie się w końcu na odwagę cywilną i na te pytania odpowie. Ilu pracownikom już obcięliście pensje?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie o wiarygodność pana prezydenta i pana premiera. Jest trzaskanie obcasami, jest salwa honorowa, ale też jest petycja dotycząca obwodnicy Kargowej.

Dopiero po upomnieniu się samorządowców idzie to dalej. Dalej nic. Kolejna obietnica. Minister pana rządu pani Elżbieta Rafalska razem z wojewodą Dajczakiem składają obietnicę słubiczanom: będzie 1 mln zł na opracowanie dokumentacji wstępnej na obwodnicę Słubic. Nie ma nic. To wszystko jest bujda i tylko w kampanii wyborczej potraficie obiecywać. Obietnice to jest coś, co wam najlepiej wychodzi. Ale Polacy mają dość, dość obietnic, pustych obietnic polityków PiS-u. Dość. Panie Marszałku! Panie Premierze!

Po tych 2 latach nos rośnie panu nawet wtedy, kiedy pan siedzi i nic nie mówi. Bo o jakim dobrobycie pan mówi? O dobrobycie swoich kolegów i koleżanek, którzy dostają w spółkach Skarbu Państwa po 50 tys. za nic? O dobrobycie pana Szumowskiego? A może o dobrobycie biskupów i księży? O jakim szacunku pan mówi? Pan jest architektem rządu, który zieje nienawiścią, który zieje pogardą, który dzieli ludzi. Pan jest architektem rządu ludzi inteligentnych bezobjawowo. I mówiąc słowami Jarosława Kaczyńskiego: wara od naszych dzieci. Mówię to jako Polka i jako matka trójki dzieci.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chciałem panu serdecznie podziękować za pana exposé, ponieważ głównym bohaterem tego wystąpienia był wielki nieobecny na tej sali - Rafał Trzaskowski. Mało tego, był tak naprawdę powodem tego exposé, powodem tego punktu w Sejmie i powodem tej ustawki z panem prezydentem. To jest istota tego dzisiejszego posiedzenia. Rzadko się zdarza taka wielkoduszność w tak ostrym sporze politycznym, aby głównemu swojemu rywalowi oddać taką cześć i taką uwagę. Ale równocześnie chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj emocje na tej Izbie są bez znaczenia, bo dzisiaj prawdziwe emocje są w Gdańsku z Rafałem Trzaskowskim. I z całego kraju idzie szept: mamy dość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Tak się zastanawiam, po co z nas pan robi sobie jaja. Po co to? Czy jest aż tak źle, że musicie pokazać swoją prawicową, PiS-owską jedność? Czy chcecie przykryć przewały swoich ministrów? Co pan jeszcze nam zaproponuje, żeby zwrócić uwagę na PiS i na Dudę? Będziecie aresztowali właścicieli rowerów, zamkniecie niezależne media, ustawowo obniżycie ceny żywności czy to, co dla was jest najważniejsze, może zaczniecie układać listy przebojów? Proszę pana, jest pan takim samym cynikiem jak ja albo jeszcze większym. Natomiast ja nie jestem kłamczuchem. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Panie premierze, jak można zaufać rządowi, który jako jedyny blokuje Europejski Zielony Ład, który ryzykuje, naraża Polaków na utratę 64 mld euro z funduszu odbudowy? Rozmontowaliście państwo państwo prawa.

Jak można zaufać komuś, kto od 5 lat nie zrobił nic w kwestii suszy, dopuścił do 8,5 mld strat rocznie u rolników, a teraz ogłasza śmieszny plan małej retencji, stojąc przy zbiorniku dużej retencji. Od 2 dni śmieje się z tego, proszę państwa, cała Polska. Poseł Krzysztof Gawkowski, klub Lewicy. Panie Marszałku! Panie Premierze! Pan premier jest jednak spryciarzem. Przybył do Sejmu, poprosił o to, żebyśmy debatowali. Zrobił najtańszą konwencję wyborczą w dziejach III Rzeczypospolitej. Mam, panie premierze, jedno ważne pytanie do pana. Plotki są na mieście, że ostry cień mgły chce na Stadionie Narodowym zorganizować największe, centralne oczko wodne. Pytam o to nie bez przyczyny, panie premierze, dlatego że podobno Kazik zaczął pisać o tym piosenkę. W związku z tym lepiej o tym wiedzieć, żebyście jej później nie ocenzurowali. Pytam o to, panie premierze, bo pan chce tutaj poważnie, to my poważnie.

Poseł Mirosława Nykiel, klub Koalicja Obywatelska. Panie Premierze! Jaki trzeba mieć tupet, by uprawiać propagandę sukcesu w czasie, gdy kolejne firmy upadają, a Polacy tracą pracę? Jak trzeba się bać zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, by w ostatniej chwili zgłaszać wniosek o wotum zaufania, aby uprawiać propagandę sukcesu? W swoim krzykliwym i kłamliwym wystąpieniu powiedział pan, że 5 lat temu otworzyły się drzwi do dobrej zmiany.

To, co dla was i znajomych jest dobrą zmianą, dla milionów ciężko pracujących Polaków jest czasem poniżenia, wstydu, podwyżek cen i podatków. Pani poseł Anita Sowińska, klub Lewicy. Panie Premierze! To pan bezczelnie kłamie i mydli ludziom oczy, ale ludzie to widzą i nie dadzą się już nabrać na kolejne pana oszustwa. Mam do pana pytanie: Dlaczego w ustawie COVID-owej wykluczyliście Prawo zamówień publicznych? I nie mówię tu tylko o przetargach, ale również o zamówieniach z wolnej ręki i zapytaniach o cenę. Czy po to, aby tabuny Szumowskich mogły się uwłaszczać na kryzysie? O to wam chodzi? O bezkarność polityków i kolesi, którzy wydają nasze pieniądze i zbijają na tym majątki? Gdzie jest to prawo, które macie w nazwie, gdzie jest ta sprawiedliwość?

Panie Premierze! Mówił pan bardzo długo, oskarżał kłamliwie na prawo i na lewo, ale nie odpowiedział pan na istotne pytania, na te pytania, które dzisiaj zadają panu Polacy, o aferę Szumowskich, o aferę Kaczyńskiego i jego srebrnych wież, o aferę Banasia, o aferę Sasina. Nie powiedział pan dzisiaj nic na temat śmierci Igora Stachowiaka, szczególnie że pańska Policja tak brutalnie spacyfikowała przedsiębiorców na ulicach Warszawy. Gdzie milion mieszkań? Gdzie milion polskich aut elektrycznych? Pytania o pański majątek przepisany na żonę. Pytania o majątek pana ministra Szumowskiego przepisany na żonę. Ilu jeszcze pańskich współpracowników przepisało swój majątek na swoje żony i mężów?

Dziękuję. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Panie Marszałku! Mówi pan premier o tym, że Polki i Polacy potrzebują spokoju, wyważonych i rozsądnych działań polskiego rządu. Tymczasem wasz rząd na problem katastrofy klimatycznej zamyka oczy. Co robicie, co zamierzacie robić z problemem suszy? Co zamierzacie zrobić, aby zapobiec katastrofie, która najbardziej dotknie przyszłe pokolenia? Interesuje was władza i ta kadencja, nie przyszłość. Panie premierze, nie walczycie z suszą, nie podejmujecie działań w sprawie katastrofy klimatycznej, nie wspieracie rolników. Gdzie ustawa antysuszowa? Co robicie? Negujecie naukowe fakty. Betonujecie rzeki i osuszacie Polskę, budując np. Kaskadę Dolnej Wisły, stopnie wodne w Siarzewie czy Kanał Krakowski. To jest bilans waszych rządów dewastacja środowiska naturalnego i niszczenie przyszłości naszych dzieci. Dziękuję. Poseł Michał Krawczyk, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! Grunt się wam pali pod nogami. Wasze sondaże spadają, Polacy są wściekli i mówią: mamy dość. A wy co robicie? Rozpaczliwie próbujecie szukać ratunku w wotum zaufania dla rządu. Ogłasza pan plan Dudy, tylko problem polega na tym, że jednym z jego głównych elementów jest oczko wodne dla każdego.

Chwali pan Ministerstwo Aktywów Państwowych, to samo, które zmarnowało 70 mln zł z naszych podatków na wybory, których nie było. Marnuje pan prawie pół dnia polskiego parlamentu na ten polityczny spektakl.

Poseł Krzysztof Śmiszek, klub Lewicy. Panie Premierze! Opisywał pan rzekome sukcesy w negocjacjach finansowych. Nie wspomniał pan o jednym drobnym szczególiku, że to są na razie propozycje unijne. Skuteczność to będzie pan mógł dopiero pokazać w negocjacjach z Radą czy w Parlamencie Europejskim. Tam w sojuszu z takimi tuzami polityki europejskiej, jak Beata Kempa, Patryk Jaki czy Beata Szydło, będzie pan mógł się wykazać, jak te pieniądze pozyskiwać. Jak na razie to wasza polityka prowadzi do pozbawiania Polski środków unijnych. Za te wasze lokalne sojusze z fundamentalistami Komisja Europejska przed chwilą ogłosiła, że jest zagrożenie dla środków finansowych dla takich województw, jak małopolskie, świętokrzyskie czy podkarpackie - tam przecież rządzicie. Za rasizm, za homofobię, za nietolerancję. Zamiast włączać, wykluczacie. Zamiast łączyć, dzielicie. Zamiast sprawiedliwie dzielić, sami napychacie sobie kieszenie krociami.

Wysoka Izbo! Wystąpienie pana premiera to propaganda sukcesu. Jak te sukcesy mają się do sytuacji w służbie zdrowia i zadłużenia ponad 90% polskich szpitali na kwotę 14 300 mln? Na szpitale nie macie, ale Szumowskim dajecie. Jak te sukcesy mają się do obiecanych dopłat bezpośrednich dla rolników, dla 126 tys. polskich rolników? Jak te sukcesy mają się do zrównoważonego rozwoju kraju, który pan premier obiecywał, i najbiedniejszych regionów, jakim jest Lubelszczyzna, gdzie przyjeżdżacie przed wyborami, obiecujecie zamówienia rządowe, śmigłowce bojowe, których do dzisiaj nie ma? Pan premier to samochwała, a samochwała w kącie stała.

Panie Marszałku! W wystąpieniu pana premiera jednego zabrakło, zabrakło konkretów moim zdaniem. Chciałem panu premierowi pomóc. W tej propagandzie sukcesu, jak o tym mówiła moja przedmówczyni, zabrakło porównań. Pozwólcie państwo, że porównamy sytuację w Polsce nie z Europą Południową, nie z Francją, nie z Hiszpanią, a porównamy ją z sąsiadującą Słowacją. Zachorowalność w Polsce - 604 osoby na 1 mln, na Słowacji - 279 na 1 mln. Pan do perfekcji opanował sztukę prezentacji, nie tylko w PowerPoincie, jak widzimy, ale rzeczywistość skrzeczy. Poseł Jan Grabiec, klub Koalicji.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wszyscy się zastanawiamy, po co pan dzisiaj przyszedł do Sejmu prosić o wotum zaufania dla rządu w czasie, kiedy Polska walczy z epidemią, kiedy ludzie się zastanawiają, czy będą mieli pracę, czy firma przetrwa, jak wyjść z kryzysu gospodarczego. Pan chce, żebyśmy wszyscy zajmowali się pana rządem. Ale kiedy usłyszeliśmy w pana głosie strach, zrozumieliśmy, o co tutaj chodzi. Pan się po prostu boi.

I to wszystko się wyda pomimo tego dzisiejszego spektaklu, bo wiele rzeczy robicie w świetle dnia. 2 mld na propagandę w TVP wtedy, kiedy w Europie zaczyna się epidemia - to wasz pomysł, to Polacy zobaczyli.

Wysoka Izbo! Panie Premierze! Rozpływał się pan, jaki to mamy w Polsce dobrobyt. Panie premierze, ceny w Polsce w kwietniu tego roku w porównaniu do kwietnia ub.r. wzrosły przeciętnie o 4%, ceny usług - o 6,5%, żywności - prawie o 8%, mięsa - o 11%, pieczywa - o 9%, owoców - o 22%, wywozu śmieci - o 54%. Finansowanie służby zdrowia niestety pozostaje na poziomie 5%. Pana partia właśnie w tej chwili likwiduje porodówkę w Kraśniku. Pana partia chce sprywatyzować szpitale. Gdzie jest ten dobrobyt, panie premierze? Gdzie ta uczciwość wobec Polaków? A gdzie uczciwość pana prezydenta Dudy? Panie Marszałku! Pan tak obsesyjnie krytycznie cały czas mówi: za waszych czasów, za waszych czasów. Panie premierze, za naszych czasów to pan lubił Platformę Obywatelską. Pan był doradcą Donalda Tuska, ale też lubił pan się zabawić, bo nieźle pan balował w restauracji Sowa i Przyjaciele, o czym Polacy mogli usłyszeć. Wtedy kiedy pan lubił Platformę Obywatelską czy dzisiaj, kiedy pan lubi PiS? Ale ja panu powiem jedną ważną rzecz. Za naszych czasów, wtedy kiedy był kryzys, myśmy zwiększyli środki na inwestycje publiczne w relacji do PKB do 5%, co pozwoliło nam m.in. uchronić się przed recesją. A dzisiaj pan obniża poziom inwestycji publicznych, dlatego że wydajecie ledwo ponad 4% w relacji do PKB. Panie Premierze! Niech pan nie utożsamia walki z polską rodziną z pytaniami o dziwne fortuny niektórych polityków PiS-u. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zadam kolejne pytanie z serii tych o to, kiedy jest pan prawdziwy, panie premierze. Być może był pan prawdziwy wtedy, kiedy był pan doradcą premiera Donalda Tuska, który na Twitterze pisze - cytuję: Mateusz nie zawsze mija się z prawdą. mówił, że prezes nie ma pojęcia o współczesnym świecie i gospodarce. Mam pytanie, czy pan ma pojęcie o gospodarce i współczesnym świecie, bo wsłuchując się w pana wypowiedź, mam poważne dylematy, czy taką elementarną wiedzę pan posiada. Wtedy kiedy jest państwu wygodnie, to odwołuje się pan do budżetu Unii Europejskiej i mówi o swoich sukcesach. Wtedy kiedy Wspólnota Europejska domaga się ochrony partykularnego interesu państwa polskiego, walczy o to, aby polski rząd przestrzegał polskiej konstytucji, to wam jest nie na rękę. Pan poseł Cezary Grabarczyk, klub Koalicji Obywatelskiej.

Wysoka Izbo! Panie Premierze! Pan premier już wie, że to nie był dobry pomysł z wnioskiem o wotum zaufania, [[Oklaski]] ale autor tego pomysłu przyznał się publicznie i już opuścił Sejm. Rozpoczął pan pytaniem, czego dziś potrzebują Polacy. My słyszymy odpowiedź, bo gdy Polacy podpisują listy poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, opowiadają: chcemy uczciwego, moralnego państwa, a państwo PiS takie nie jest. Państwo PiS symbolizują dziś interesy instruktora narciarskiego i rodziny Szumowskich. Państwo PiS symbolizują dwie wieże i koperta Kaczyńskiego. Także pan jest symbolem państwa niemoralnego. Wie pan, co opowiadają dziś Polacy? Polacy mają dość i powiedzą to już niedługo w wyborach.

Panie Premierze! Pan mówi, że prowadzicie politykę dla ludzi? Chyba dla ludzi związanych z PiS. Setki milionów złotych dla firm związanych z rodziną ministra zdrowia, miliony złotych na felerne maseczki dla instruktora narciarstwa, setki tysięcy złotych na przyłbice od znajomego, który nie zajmował się handlem środkami ochrony zdrowia, tylko handlem oscypkami. Taka jest prawda o waszej polityce dla ludzi. Pan mówi, że prowadzicie politykę inwestycji. Gdzie jest 100 tys. mieszkań dla młodych, które pan obiecał? Gdzie są promy? Nie ma. Gdzie są elektryczne samochody? Nie ma. Gdyby Pinokio z tej mównicy wypowiadał słowa o pańskich obietnicach, to nosem wybiłby szybę w drzwiach na końcu tej sali. Pana rząd nie zasłużył na zaufanie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W swoim populistycznym wystąpieniu pan premier Morawiecki pytał, czego potrzebują Polacy, a potem sam sobie odpowiadał, że potrzebują skuteczności i sprawiedliwości. No to trochę o waszej skuteczności. Czy miarą pana skuteczności jest zakup maseczek bez atestu od kumpla z nart pana ministra Szumowskiego, czy może 70 mln wyrzucone w błoto przez pana Sasina?

W tym rzeczywiście jesteście najlepsi, w tym pan jest bardzo dobry. Całe państwo, którym pan teraz zarządza, zajmuje się jedną rzeczą: ukrywaniem afer PiS-u. To jest ta wasza skuteczność i o tej skuteczności pan mówił.

Polacy boją się tego, że trafią do szpitala, do którego Ministerstwo Zdrowia wysłało trefne maseczki kupione za 5 mln zł od instruktora narciarstwa, znajomego ministra waszego rządu. Polacy mają dość tego, że jeżeli nikt nie będzie patrzeć na ręce waszemu rządowi, to jeszcze więcej publicznych pieniędzy trafi do waszych rodzin, do waszych znajomych. Polacy mają dość tego, że wszystkie zapowiadane wielkie inwestycje oznaczają wielkie pieniądze dla waszych znajomych, dla waszych rodzin. Panie Premierze! Stawiając dzisiaj po rozmowie z Andrzejem Dudą wniosek o wotum zaufania, znowu zajmujecie się samymi sobą, czyli nie tym, za co płacą wam Polacy.

Wysoki Sejmie! Był pan dzisiaj w transie, ale przy ulubionym przez pana stole ping-pongowym nie wygrałby pan nawet jednego seta. Bo jest pan w nieustającym transie nienawiści, buty i pogardy, nieustającym transie dzielenia Polski i Polaków. Dzisiaj mówił pan: my i oni, lepszy i gorszy sort. A mądry premier powinien bardziej słuchać nie własnych klakierów, a właśnie opozycji. Dzisiaj potwierdził pan, że jest pan premierem partyjnym, nie jest pan premierem Polski. Dlaczego? Dlaczego właśnie dzisiaj, 4 czerwca, w tak ważnym dniu dla Polski, pan tę partyjność potwierdza? Pana wystąpienie to Niagara tępej propagandy, jak za najgorszych czasów. Musi panu brakować tlenu w czasie kampanii, a sejmowanie to nie wiecowanie. Dlatego ja przypomnę panu: mamy dość. A jeśli pan ma dość, to proszę poprzeć listę kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy do nas. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Jedna z waszych megalomańskich wizji dotyczy mojego regionu, mojej małej ojczyzny. Nazywa się „Program dla Śląska” Miał być wydarzeniem epokowym dla regionu, a jednak cicho o nim ostatnio. Miały być regularne raporty, które obiecywaliście państwo w odpowiedziach na moje interpelacje, a raportów brak. Miały być miliardy na inwestycje, a póki co skończyło się na stronie internetowej za kilkaset tysięcy złotych. Miał być doświadczalny poligon dla dronów, a był seksualny skandal w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i związane z nim odwołanie zarządu jednej ze spółek córek. Mam dość waszej propagandy. Czekam, aż pokażecie, co naprawdę zrobiliście dla Śląska. Poseł Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Jesteście już tak słabi, że dzisiaj chcecie pokazać, że macie poparcie Jarosława Gowina. Natomiast to jest dobry moment, żeby rozpocząć rozliczenie waszych rządów. Efektem waszych rządów jest dramatyczne obniżenie potencjału bojowego Sił Zbrojnych. Mieliśmy czarną serię lotnictwa, katastrofy, cztery samoloty bojowe zniszczone, jeszcze więcej śmigłowców.

Pan jako minister nie zawarł umowy na zakup śmigłowców, twierdząc, że offset był niewystarczający, ale pana rząd zawarł teraz umowę na zakup samolotów F-35 w ogóle bez offsetu. I jeszcze jedna sprawa wielkich inwestycji. Zawsze je rozpoczynacie w kampanii wyborczej. W 2015 r. obiecywaliście budowę bloku węglowego w Ostrołęce. Poseł Barbara Nowacka, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Premierze! Musiał pan tu przyjść pokrzyczeć, zapytać, czy koledzy pana popierają. Może pan pójdzie do TV PiS, może tam jeszcze pana pogłaszczą. Bo ludzie, ci ludzie spotkani na ulicach, już po prostu was nie chcą, bo widzą tę skalę obłudy i hipokryzji. Staliście się elitą, elitą władzy i arogancji, elitą pychy, a zapominacie o tych, którzy wam byli potrzebni tylko do wyborów. Chcecie budować wspólnotę, a dzielicie i wykluczacie. To nie jest patriotyzm, panie premierze - pokrzykiwanie. Patriotyzm to dbanie o biedniejszych. Mieliście budować mieszkania. Dzisiaj proponujecie oczka wodne w ogródku dla bogatszych. Popatrzcie, jak galopują ceny. Likwidujecie szpitale powiatowe. I to najbiedniejsze osoby za waszych rządów mają źle. I dlatego ci ludzie mówią wam: dość.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiejsze przedstawienie miało tak na dobrą sprawę przykryć aferę ministra Szumowskiego, ale nie przykryje. Otóż było dużo o pandemii, pan o tym mówił, ale jakoś dziwnym trafem nic pan nie wspomniał o dostawcy lewych maseczek, przyłbic, testów, nic pan nie wspomniał o największym chyba w historii konflikcie interesów ministra w rządzie, gdy przekazano spółkom powiązanym z nim prawie 200 mln zł.

Panie premierze, chcę panu powiedzieć tak. My w Polsce musimy jeszcze na ten czas poczekać. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Pan mówi o uczciwości. No to niech pan wreszcie w końcu tutaj stanie i wszystkim Polakom powie, jaki jest pana majątek. Bo wszyscy chcieliby znać tę odpowiedź. Jeszcze kilka miesięcy temu razem z pana pomocnikiem wicepremierem Sasinem co pan mówił wszystkim Polakom? Ceny prądu nie wzrosną. A o ile wzrosły? O kilkanaście procent. Kolejne kłamstwo. Mówiliście o tym, że tylko i wyłącznie będziemy zużywać polski węgiel. A jaka jest prawda? Pan mówił o kwestii dotyczącej młodych, jakie to jest ważne - perspektywa. Ile wybudowaliście mieszkań? A prawda jest jasna. Bo pan prawdę mówił tylko raz, w Sowie i Przyjaciołach. Co pan mówił o młodych? Co pan mówił o młodych? Trzeba obniżać ich oczekiwania, będą (...) za miskę ryżu.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ewidentnie macie problem z kandydaturą tak silnej osobowości, jaką jest Rafał Trzaskowski.

Może warto uwierzyć Polakom, którzy wiedzą, kogo mają wybrać, bo Polacy to mądrzy i rozsądni ludzie.

Poseł Agnieszka Hanajczyk, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po pana wystąpieniu przeczytałam w mediach społecznościowych taki wpis, że pan całkowicie odleciał. Może nie byłabym tak ostra w ocenie. Mnie się wydaje, że pan nieustająco ogląda filmy o Avengersach. Nawet więcej, panu się wydaje, że pan jest superbohaterem, [[Wesołość na sali]] że pan jest takim Kapitanem Ameryką. Nawet się nie chcę domyślać, kto jest kapitanem, Iron Manem. Nie przepadam za Kapitanem Marvelem, tak że nie chcę o tym myśleć. Ale muszę pana rozczarować, panie premierze. Pan mówi o imposybilizmie, a ja twierdzę, że dzisiaj w pana wystąpieniu było dużo infantylizmu. Mało tego, oni w ogóle nie żyją jak w filmie. Nie wiem, czy pan wie, jakie jest ubóstwo, o czym myślą dzisiaj przedsiębiorcy, [[Dzwonek]] o czym myślą dzisiaj pracownicy, jak wygląda służba zdrowia. Poseł Krzysztof Piątkowski, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie Premierze! Nie udał się panu ten dzisiejszy spektakl. To kiepski spektakl, a jego finał wszyscy znamy. Pana koledzy nie rozczarują, zagłosują tak, jak prezes zdecydował. Zachowacie swoje posady jeszcze przez chwilę, bo potraficie zadbać przede wszystkim o siebie. A tych, którzy was krytykują, którzy was nie cenią, którzy mają odwagę mówić prawdę, ośmieszacie, kpicie z nich, poniżacie za 2 mld zł podarowane publicznej telewizji. Zrobiliście to polskim nauczycielom, lekarzom, sędziom, a ostatnio obrońców nazwaliście mataczami. Powiem, za co dostaniecie dzisiaj wotum zaufania.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Naprawdę chcę zapytać zupełnie poważnie w imieniu osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, kiedy zrealizujecie, panie premierze, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., o który sami wnosiliście. Mija prawie 5 lat, a wy nie potraficie tego wyroku zrealizować. Nam udało się podnieść świadczenie pielęgnacyjne, tak żeby opiekunowie, rodzice dzieci niepełnosprawnych mieli dzisiaj ponad 1800 zł, ale opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych mają niecałe, ponad 600 zł. I wy tego drugiego kroku nie potraficie zrobić. Mało tego, miał powstać specjalny system orzecznictwa, pan podpisał się pod zarządzeniem, że to będzie do końca czerwca 2018 r. Nie ma go, a Fundusz Solidarnościowy, który stworzyliście na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, tak naprawdę im zabraliście. Poseł Monika Wielichowska, klub Koalicji Obywatelskiej.

Nie zauważył jednak, że to już nie działa, że Polki i Polacy mają dość. Zamiast bajdurzyć, lepiej pokazać zrealizowane obietnice, więc pytam: Kiedy oprowadzi pan prezydenta Dudę po 100 tys. wybudowanych mieszkań dla młodych? Kiedy zabierze pan prezydenta kandydata na przejażdżkę jednym z miliona elektrycznych samochodów? To może chociaż prototypem. Pojechalibyście wtedy po tych 100 wybudowanych mostach, przez te 100 nowych obwodnic, a podczas przejażdżki prezydent opowiedziałby panu, jak to chciał, ale nie podniósł kwoty wolnej od podatku, jak to chciał, ale nie zlikwidował umów śmieciowych, jak to chciał, ale nie obniżył podatku VAT, jak to chciał pomóc frankowiczom, ale ich zawiódł, jak to chciał dać dopłaty rolnikom, ale nie zdołał. Poseł Waldemar Andzel, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować na wstępie rządowi Prawa i Sprawiedliwości [[Wesołość na sali, oklaski]] i rządowi premiera Mateusza Morawieckiego za skuteczne rozwiązywanie problemów pandemii koronawirusa. Jak szybko działał polski rząd, wprowadzając ograniczenia związane z epidemią koronawirusa? Jak to wygląda na tle innych państw Europy Zachodniej, panie premierze? Totalna opozycja tylko tutaj przeszkadza i szkodzi Polsce. Mam pytanie także do pana premiera: Ile wynosi wartość pakietów pomocowych przygotowanych dla polskich przedsiębiorców i pracowników? Pan poseł Henryk Kowalczyk, klub Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! To jest kontekst radzenia sobie w czasach pandemii zarówno z chorobą, jak i gospodarczo. Ale też oceniamy dokonania ostatnich lat, kiedy to właśnie udało się temu rządowi przekazać środki finansowe polskiej rodzinie.

Ja wiem, że opozycja pewnie zagryza zęby z wściekłości, że nie ma tysięcy zarażonych, [[Wesołość na sali]] że nie ma tysięcy zmarłych. Nie ma nieszczęścia, ale to jest wszystko dzięki bardzo roztropnym decyzjom ministra Szumowskiego i premiera Morawieckiego. Tak, te roztropne decyzje Polacy doceniają [[Dzwonek]] i są za te decyzje wdzięczni. Ogłaszam 3 minuty przerwy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Notowałem tutaj większość pytań.

Niektóre z nich postarałem się pogrupować i niektóre mają charakter bardziej ogólny, więc pozwolę sobie również na kilka bardziej ogólnych komentarzy.

Otóż, szanowni państwo, przede wszystkim jeśli chodzi o zakup śmigłowców, to to, co przyświecało nam z panem ministrem obrony narodowej, z panem ministrem Błaszczakiem i wcześniej z panem ministrem Macierewiczem, to kwestia budowy potencjału polskiego tam, gdzie tylko można. Niestety nie mamy jeszcze takich zdolności produkcyjnych, kompetencji i technologii, żeby samoloty klasy F-35, F-16 w jakikolwiek sposób współkonstruować, w związku z tym rzeczywiście zakup w przypadku F-35 odbył się bez offsetu. Mówiliśmy o tym głośno po to, żeby jak najszybciej można było tego zakupu dokonać. Chyba rok czy 2 lata temu poseł Platformy Obywatelskiej pan Siemoniak mówił o tym, że Wojska Obrony Terytorialnej to weekendowcy w mundurach, a pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że trzeba Wojska Obrony Terytorialnej zlikwidować, bo nikomu nie służą.

Chcę zatem bardzo wszystkim żołnierzom, podobnie jak służbie zdrowia, ale właśnie żołnierzom i też żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej bardzo serdecznie podziękować za wasze wsparcie. Chcę bardzo konkretnie na nie odpowiedzieć. Otóż była mowa o dopłatach do materiału siewnego. Chcę podkreślić - być może pani poseł nie miała kompletnych informacji - że nastąpiła wypłata w pełni wszystkich, w całości wszystkich dopłat do materiału siewnego. Ubezpieczenia rolnicze. Tutaj również nie ma żadnych zaległości. Proszę sobie sprawdzić to w budżecie. My przeznaczamy znacząco większe kwoty niż państwo na ubezpieczenia rolnicze. Było pytanie również w obszarze rolnictwa o susze. Już odpowiadam. Jeśli chodzi o suszę, wypłaty nastąpiły dla 92% wszystkich rolników. Oprócz tego chcę podkreślić tę różnicę, bo naprawdę posłowie opozycji, którzy mówią o suszy, niech pro domo sua w tym przypadku, uderzą się we własną pierś i popatrzą, ile wy wypłacaliście przy podobnej suszy w 2015 r. Otóż wypłaty w przypadku Platformy Obywatelskiej i PSL wynosiły ok. 400 do 500 mln zł.

Teraz mówiliście państwo w kilku głosach o sprawach społecznych, o kwestiach osób bezrobotnych. To jest ten temat, który rządowi Zjednoczonej Prawicy leży bodaj, podkreślę to, najbardziej na sercu.

Otóż chcę to podkreślić, że przyrosty bezrobotnych to dla nas jest zawsze tragedia, zawsze to jest dramat ludzki, ale też trzeba pokazywać te przyrosty w zestawieniu z krajami Europy Zachodniej i krajami Europy Wschodniej. W tym przypadku widać, że tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa działa, że staramy się chronić miejsca pracy. Spójrzcie na statystyki ministerstwa rodziny, spójrzcie na statystyki Eurostatu, na przyrosty bezrobocia w krajach Europy Środkowej, chociażby w Bułgarii, w Rumunii w ostatnim czasie. Pytaliście mnie, pytaliście również o przykłady z Europy Wschodniej, więc je podaję. W Europie Zachodniej przyrost bezrobocia w Hiszpanii, we Włoszech czy Francji w tych obszarach. w tych krajach bardzo mocno rzeczywiście wystąpił. Cieszę się, że nasze programy przede wszystkim są ukierunkowane na obronę miejsc pracy i rzeczywiście to na razie się sprawdza. Będziemy robili wszystko, żeby w najbliższych miesiącach sprawdzało się jeszcze lepiej. W tym kontekście chcę też podziękować bardzo panu prezydentowi za pomysł i za propozycję legislacyjną dotyczącą dodatku solidarnościowego. Drodzy Państwo! Wysoka Izbo! Dla niektórych z państwa to jest ściema, a ja powiem, że to jest ratunek dla wielu osób. Dziękuję, panie prezydencie, za to, że dodatkowo zaproponował pan i, mam nadzieję, że Wysoka Izba to przegłosuje, dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł netto, bo będzie to pewne wsparcie dla osób, które zostaną dotknięte tragedią bezrobocia. Mam nadzieję, że przejściowego. Były pytania o ochronę zdrowia, o nakłady na ochronę zdrowia. Otóż, drodzy rodacy, Wysoka Izbo, niech to wybrzmi tutaj: między rokiem 2008 a 2014 na ochronę zdrowia koalicja Platformy i PSL wydawała w proporcji do PKB mniej. I to, szanowna pani poseł, tą samą miarą, która jest dzisiaj. Przecież gdybyśmy robili to w proporcji do PKB na ten rok, zakładając we wrześniu zeszłego roku, to pomylilibyśmy się bardzo, ponieważ był planowany wzrost 3,8%, a będzie prawdopodobnie spadek PKB, spadek najmniejszy wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, to warto podkreślać. W związku z tym, tak na to patrząc, dzisiaj trzeba podkreślić, że wydatki na służbę zdrowia przekroczą w tym roku 5%.

W naszym przypadku - ponad 5% w tym roku. Było pytanie o PROW, o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otóż tutaj już 70% środków zostało zakontraktowanych i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich korzystają coraz lepiej i coraz chętniej kolejni beneficjenci. Jestem przekonany, że zmieścimy się w terminie, zmieścimy się w budżecie.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo, a zwłaszcza szanowni państwo posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy bardzo mocno optowaliście za tym, ubiegaliście się o te dodatkowe dopłaty, odnieśliśmy, już dzisiaj mogę powiedzieć, wielki sukces, też dzięki naszemu komisarzowi panu Januszowi Wojciechowskiemu. Zaproponowaliśmy Unii Europejskiej większe wydatki na wspólną politykę rolną i te większe wydatki, o 24 mld euro, są ujęte w przyszłej perspektywie. To już powoduje, że te dopłaty, przyspieszanie wzrostu do średniej dopłat będzie na pewno dużo szybsze niż w przypadku rządów PSL - Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo! Było pytanie o osoby niepełnosprawne. Tutaj warto podkreślić ten dodatkowy, finansowy dodatek, który zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy. To jest realny dodatek. To jest dodatek 500 zł, który jest doceniany przez te środowiska. Miałem spotkanie z tymi środowiskami, z fundacjami, stowarzyszeniami. Zawsze ta pomoc jest za mała, ja się z tym zgadzam. Zawsze będziemy dążyć do tego, żeby najsłabsi członkowie naszej wspólnoty, naszej wspólnoty narodowej, dostawali więcej wsparcia ze strony państwa. były to wydatki wielkości 15 mld zł. Znacząca różnica.

Natomiast ponieważ tutaj mówiliście o różnych sprawach związanych z dzieleniem i pan Trzaskowski, pan Rafał Trzaskowski również coś takiego podniósł. Czy ci, którzy stosują taktykę opozycji totalnej, taktykę przeciwstawiania się wszystkiemu, co dobre, a potem, po latach zgadzają się, że coś było rzeczywiście dobre, i w panice zmieniają swoje zdanie, jak w stosunku do 500+ czy naszej polityki gospodarczej. Ja dzisiaj podawałem mnóstwo faktów, mnóstwo liczb. Nie odnieśliście się do tego. To jest wezwanie do rozmowy o faktach, do rozmowy o tym, co może stanowić dobry punkt startu do wspólnego mianownika w różnych sprawach. My jesteśmy otwarci na współpracę, również z opozycją, przez najbliższe 3,5 roku.

To poprzez totalne zaprzeczanie wszystkiemu, co dobre, poprzez manipulowanie, poprzez wysługiwanie się waszą propagandą, bo tak, to wy przede wszystkim posługujecie się propagandą waszych mediów. mediów niestety w większości po waszej stronie, bo tak wyglądała III Rzeczpospolita.

Szanowni Państwo! Teraz jedno pytanie. Ponieważ tutaj były również pytania o wynagrodzenia w administracji i w innych miejscach, to chcę zapytać o wynagrodzenia dyrektorów ratusza warszawskiego. Widzę, że próbujecie teraz w panice je zakrzyczeć, ale one są ważne. Drodzy rodacy, spójrzcie, ile zarabiają. nawzajem sobie różne synekury podsuwając, dyrektorzy ratusza warszawskiego. Uwypuklijmy to, bo wtedy może się okaże. CPK. ...że ministrowie rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zarabiają o wiele mniej niż dyrektorzy ratusza warszawskiego. W jednej kwestii chcę się zgodzić z panią posłanką, z panią poseł bodaj Scheuring-Wielgus, jeśli dobrze pamiętam, która powiedziała: wara od naszych dzieci. Tak, pani poseł, wara od naszych dzieci. Były też tutaj ataki na Policję, ataki oczywiście werbalne na Policję, na jej rolę. Otóż, szanowni państwo, chcę podziękować wszystkim policjantom, panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu za znakomite nadzorowanie pracy Policji, za bodaj, jeśli dobrze pamiętam, 7 mln. To właśnie jest też część sukcesu walki z koronawirusem. Pytaliście państwo o przedsiębiorców, pytaliście o to, ile osób otrzymuje wsparcie.

Bo owszem, ten kryzys jest absolutnie wyjątkowy. Nigdy wcześniej ekonomiści nie mierzyli się w teorii z takim kryzysem, nikt wcześniej nie przewidział takich możliwości. Jednocześnie też to szok popytowy, a w tym samym czasie też porwane linie dostaw, linie produkcji, a więc i szok podażowy. Spytajcie o to przedsiębiorców, bo zdaje się, że na antenie radia wasz poseł Krzysztof Truskolaski chwalił tę tarczę, jak również pan przewodniczący Budka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za takie pochwały. Myślę, że wypowiadane poza kamerami, jak pan sądził, są najszczersze. Ale najważniejsze dla mnie jest to, że te tarcze poprzez przedsiębiorców ratują miejsca pracy. Każda kolejna tarcza.

pozytywnie tutaj oceniła i przegłosowała, dziękuję, dziękuję za tę współpracę. Chciałbym, żeby ona była jak najczęstsza. Otóż, szanowni państwo, europejski fundusz odbudowy to kolejny sukces, który kłuje was w oczy, [[Oklaski]] to wielki sukces, bo próbowaliście coś mówić o europejskich pieniądzach wtedy, kiedy ich nie było. Naprawdę nie było żadnych nowych środków, po prostu było przesunięcie z poprzedniej perspektywy na ochronę zdrowia. Od kwietnia głośno mówiłem o ambitnym planie dla Europy, o planie Marshalla dla Europy. Przeczytajcie sobie w kilku gazetach zachodnich.

Owszem, z bardzo dobrej współpracy z Grupą Wyszehradzką w ramach Trójmorza, również z Rumunią, również z Bułgarią, z innymi państwami Europy Środkowej, a nie jedynie z możnymi tego świata. A więc europejski fundusz odbudowy, tak, będzie znakomitym, wielkim dodatkiem przez duże D do wieloletnich ram finansowych, do tego budżetu, który wynegocjujemy przez najbliższe kilka miesięcy. I wiecie, co, Wysoka Izbo, szanowni państwo? To będzie również bardzo dobry budżet dla Polski, ale najważniejsze jest to, że. Bo kiedy tarcza europejska wejdzie w życie? Orientujecie się państwo? Mniej więcej jesienią, może nawet na początku przyszłego roku. Tak się dzisiaj mówi. Jak by wyglądali polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy do zimy tego roku, do grudnia, gdyby nie było pomocy państwa polskiego, bezpośredniej pomocy z tarcz finansowej i antykryzysowej? Jak by wyglądali? Zadajcie sobie to pytanie i szczerze na nie odpowiedzcie. Powiem w ten sposób: w czasach Platformy Obywatelskiej i PSL-u odziedziczyliście dług w wysokości ok. 515 mld zł. jak dobrze pamiętam. Kiedy my przejmowaliśmy rządy, było to 888 mld, ale do tego trzeba dodać, żeby porównywać jabłka z jabłkami, 160 mld z OFE, które obiecywaliście, że nie zabierzecie ludziom, a zabraliście, Platforma Obywatelska zabrała środki z OFE ludziom.

Ale mam jeszcze dwie dobre wiadomości. Nie wiem, czy one was dzisiaj jeszcze interesują, ale powiem, bo myślę, że każdy patriota ucieszy się, a właśnie na to liczę, jak mówię o tym, że dzielenie na opozycję totalną czy dzielenie Polaków na tych lepszych i gorszych, które niestety przebija. Otóż potężnym zagrożeniem dla długofalowego, wieloletniego rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej było uzależnienie od długów w walutach i długu zagranicznego.

To się nazywa mądra polityka gospodarcza, to jest bufor, który broni nas przed różnymi wahaniami walutowymi. A wiec tutaj też mamy dobre wiadomości. Było pytanie o maltretowanie zwierząt, o zapisy. Szanowni państwo, odrzucamy jakiekolwiek zapisy.

Nie wolno tak się zachowywać. Było również pytanie o „Program dla Śląska”, o zaangażowanie środków w „Program dla Śląska” Otóż „Program dla Śląska”, który pierwotnie był programem zaplanowanym na 42 mld zł, dzisiaj został rozwinięty do 55 mld zł. Z tego zaangażowanych zostało 44,5 mld zł w łącznych projektach, czyli ogromna większość, a w już zaangażowanych środkach budżetowych są 24 mld zł. Czyli, szanowni państwo, jest konkret, są konkretne działania.

To jest projekt, który my zatwierdziliśmy i my realizujemy, podobnie jak liczne inne projekty infrastrukturalne. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za te merytoryczne pytania.

Wtedy bojkotowałem te wybory, ale po latach mogę i chcę przyznać, że trzeba było wejść w tę przestrzeń budowania demokracji. Potem trzeba było tę przestrzeń w ramach III Rzeczypospolitej poszerzać. I chcę podziękować wszystkim tym, którzy przez lata III Rzeczypospolitej przestrzeń demokracji, wolności, solidarności i sprawiedliwości poszerzali, [[Oklaski]] przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwości, ale też wszystkim innym ludziom dobrej woli, [[Wesołość na sali]] wszystkim ludziom ze wszystkich stron sceny politycznej, którzy się do takiego dziedzictwa, dziedzictwa „Solidarności” i wolnej Polski, przyznają. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy za chwilę.

Proszę państwa, przystąpimy do stwierdzenia kworum. W związku z tym bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu stwierdzenia kworum. Nie, nie tylko, pani poseł. Bardzo proszę o naciśnięcie dowolnego przycisku.

W związku z tym stwierdzam kworum. Proszę państwa, chciałabym tylko zapytać posłów, którzy zwracali się z wnioskami formalnymi, czy one są aktualne. Pan poseł Krzysztof Paszyk - wniosek formalny nieaktualny.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym złożyć wniosek formalny w imieniu klubu Lewica o przerwanie posiedzenia Sejmu, ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu w celu zmiany porządku obrad.

W naszej ocenie to kontynuacja tego, co dzisiaj o godz. 12.10 się zaczęło, a więc dalej kampania wyborcza i jest przedstawiany projekt prezydencki. W związku z tym chcielibyśmy, ażeby włączyć ten projekt do porządku obrad. żeby dyskutować, jeżeli już, o dwóch tych projektach, bo nie widzę żadnej podstawy, dlaczego projekt pana prezydenta ma być lepszy niż projekt Lewicy, tym bardziej że pan prezydent ten projekt złożył w dniu wczorajszym. Padł wniosek o przerwę, w związku z czym poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy, proszę o naciśnięcie przycisku.

się wstrzymał?

Czy wniosek pana posła Bogusława Sonika jest aktualny? Bardzo proszę, panie pośle.

Dzisiaj przypada kolejna rocznica wolnych wyborów, częściowo wolnych wyborów. To już 31 lat. Zarówno same wybory, jak i ich przygotowanie, a także wynik spowodowały niesłychany wręcz entuzjazm.

Dominowało poczucie beznadziei. Wybory 4 czerwca radykalnie to zmieniły. Polacy znowu poczuli, że coś od nich zależy. Okazało się, że ludzie gotowi są do ogromnych wysiłków, że wierzą w lepszą przyszłość, że obudziła się nowa nadzieja i nowy entuzjazm. I trudno przecenić siłę i znaczenie tego impulsu, jakim był 4 czerwca. Przykro mi bardzo. Dziękuję. Przepraszam, ale naprawdę, panie pośle, nie w tym miejscu. Proszę bardzo, czy pan poseł Grzegorz Braun podtrzymuje wniosek formalny? Proszę bardzo. Jesteśmy w tym punkcie. Za parę godzin minie 100 lat od podpisania aktu rozbiorowego ziem Korony Świętego Stefana, po południu, w pałacu Trianon w Wersalu 4 czerwca 1920 r. Wiele łączyło w historii Koronę Świętego Stefana z Koroną Królestwa Polskiego. Przedkładałem, pani marszałek, wcześniej projekt uchwały w tej sprawie. Pan podpisał się sam. Pani Marszałek! Ponieważ nie odczytam państwu tego projektu uchwały, a tym bardziej szerzej go nie uzasadnię, więc pomilczmy chwilę, pomilczmy chwilę nad tym faktem, że 100 lat temu dokonano rozbioru państwa (Dzwonek), które miało z nami wspólnych monarchów.

Przepraszam bardzo. Właściwa komisja przedstawiła opinię w sprawie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej sprawy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedłożył projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, druk nr 406. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Proponuję, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusjach nad dodanymi punktami porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. To jest pańska propozycja, panie pośle. Przystępujemy do przegłosowania sprzeciwu.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji wysłuchania 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm propozycję przyjął. Powracamy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów. Przechodzimy do głosowania. Przypominam, że zgodnie z art. 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o wyrażenie wotum zaufania Radzie Ministrów, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto się wstrzymał?

Dziękuję bardzo. Stwierdzam jeszcze raz, że Sejm wyraził wotum zaufania Radzie Ministrów. Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury o godz. 16.30. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (druk nr 406) Proszę zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Pawła Muchę.

Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Dudę projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Pan prezydent od początku pandemii aktywnie włącza się w walkę z nią, w szczególności z niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Przedstawiona inicjatywa stanowi uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Przedstawiony projekt został zapowiedziany przez pana prezydenta na początku maja. Jest także elementem umowy programowej zawartej w dniu 5 maja 2020 r. przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Omawiany projekt ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, projekt ustanawia wsparcie dla osób, które straciły pracę ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym epidemią COVID-19. Po drugie, projektowana ustawa na stałe podnosi wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Wysoka Izbo! Projektowana regulacja określa warunki nabywania, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie. Dodatek przysługiwał będzie osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i z którymi umowa o pracę została po dniu 31 marca 2020 r. rozwiązana albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni. Dodatek przysługiwał będzie osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są obywatelami polskimi, obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski. Dodatek nie będzie przysługiwał osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym mającym prawo do emerytury lub renty rolnikom. Projekt rozstrzyga sytuację, gdy osoba jest jednocześnie uprawniona do dodatku solidarnościowego i zasiłku dla bezrobotnych. W okresie pobierania dodatku solidarnościowego osobom uprawnionym nie będą wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz stypendia, jednak jeśli osobie bezrobotnej zostanie wypłacony zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ww. ustawie, wówczas dodatek solidarnościowy wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym dodatkiem solidarnościowym a zasiłkiem lub stypendium wypłaconym przez urząd pracy. Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie skracał okresu pobierania zasiłku bądź stypendium. Okres pobierania dodatku solidarnościowego będzie natomiast wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, oraz stażu pracy określonego w odrębnych przepisach wymaganego do wykonywania niektórych zawodów. Projekt, podobnie jak to czynią ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej, ustanawia także podstawę dla Rady Ministrów, aby w drodze rozporządzenia określiła dłuższy niż 3-miesięczny okres przysługiwania świadczenia solidarnościowego, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Proponuje się w szczególności dla szybkości postępowania, aby wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane były w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego będzie udostępniona na profilu informacyjnym osoby uprawnionej utworzonym w systemie teleinformatycznym ZUS. Odmowa przyznania dodatku solidarnościowego nastąpi w drodze decyzji, od której przysługiwać będzie prawo odwołania do właściwego sądu w terminie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne finansował będzie w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji. Oznacza to, że uprawniona osoba otrzyma całą kwotę 1400 zł. Jak wskazałem na początku, projekt zakłada również podwyższenie od 1 września 2020 r. zasiłku dla bezrobotnych. Prezydent proponuje, aby w okresie pierwszych 90 dni zasiłek wynosił 1200 zł, a następnie 942,30 zł. Ponadto projekt zakłada zaliczenie do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku tych osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmniejszono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Proponuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych, które wejdą w życie od dnia 1 września 2020 r. Przewidywany termin wejścia w życie ustawy nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego i jest uzasadniony szczególnie ważnym interesem społecznym. Wysoka Izbo! Szacunkowa liczba osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, które spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku solidarnościowego, wynosi ok. 307 tys. osób.

To można powiedzieć, że 200 tys. osób, które dzisiaj są pozbawione jakichkolwiek świadczeń, na podstawie tej ustawy będzie otrzymywać dodatek solidarnościowy w kwocie 1400 zł. Z drugiej strony ponad 300 tys. osób z ustalonym prawem do zasiłku dla bezrobotnych będzie to świadczenie otrzymywało w wysokości prawie 200% dotychczasowego świadczenia, bo to jest 1400 zł w porównaniu z obecną wysokością zasiłku. Poza tym mamy, tak jak powiedziałem, podwyższenie zasiłku dla wszystkich przewidywane od dnia 1 września. Chciałbym bardzo podziękować stronie społecznej - NSZZ „Solidarność” za prace nad tą ustawą, chciałbym bardzo podziękować za współpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za prace nad tą ustawą pani minister Marlenie Maląg, Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także ekspertom z ZUS, którzy nas wspierali w tych pracach. Jestem przekonany, że to jest bardzo ważna ustawa, bardzo istotna ustawa, która polepsza sytuację tych wszystkich osób, które dzisiaj wskutek COVID-19 mają absolutne poczucie niepewności czy nie mają możliwości zaspokajania podstawowych niekiedy swoich potrzeb życiowych, bo pozbawione zostały jakichkolwiek dochodów. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że zaproponowane przez pana prezydenta rozwiązania są potrzebne i oczekiwane społecznie. Uprzejmie proszę zatem panie i panów posłów o poparcie inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jak najszybsze nad nią procedowanie, aby dodatek solidarnościowy niezwłocznie mógł być wypłacony osobom, które utraciły pracę ze względu na pandemię COVID-19 i niewątpliwie oczekują na tę pomoc. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5- minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. W pierwszej kolejności usłyszymy stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Pan poseł Sylwester Tułajew. Dziękuję bardzo. 4 czerwca 1989 r. Polacy solidarnie zagłosowali za wolną Polską. Solidarność to wartość zawsze aktualna. Złożyłem projekt ustawy o dodatku solidarnościowym, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19. Będzie służył tym, którzy teraz potrzebują pomocy. Czyny, nie słowa. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To słowa pana prezydenta, który dzisiaj rano zamieścił odpowiedni tweet, właśnie pokazując całą swoją prezydenturę. Takim właśnie prezydentem jest pan prezydent Andrzej Duda - prezydentem wiarygodnym, prezydentem, który dotrzymuje obietnic. prezydentem, który skutecznie realizuje wszystkie swoje obietnice, które były złożone w 2015 r., jeszcze przed objęciem prezydentury... Frankowicze. ale przez te ostatnie 5 lat w sposób szczególny. Chciałbym podkreślić, że 1 maja pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział, zaproponował wprowadzenie dodatkowej formuły wsparcia dla każdego, kto stracił pracę w wyniku kryzysu spowodowanego wirusem COVID-19. Czyny, nie słowa. Kolejna rzecz, którą prezydent udowadnia, że jest prezydentem wiarygodnym, że jest prezydentem, który dotrzymuje słowa. Również 5 maja została podpisana stosowna deklaracja wspólnie ze związkiem zawodowym „Solidarność”

Czyny, nie słowa. Również 1 maja pan prezydent Andrzej Duda zaproponował i podkreślił potrzebę podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych, uzasadniając to koniecznością właśnie zmian w tym zakresie, bo zdawał sobie dokładnie sprawę, że nastąpi wzrost liczby osób tracących pracę na skutek COVID-19. Czyny, nie słowa. Po raz kolejny prezydent pokazał, że skutecznie realizuje swoje obietnice wyborcze. Chciałbym zwrócić uwagę, że ten projekt, bardzo dokładnie przedstawiony przez pana ministra, zakłada również szereg takich bardzo ważnych spraw. M.in. art. 6, gdzie mówi się, że wypłata dodatku będzie następować w terminie nie dłuższym niż 7 dni. To pokazuje, że właśnie chcemy działać szybko, że chcemy szybko pomagać, szybko wspierać osoby, które potrzebują pomocy. Co ważne, dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji. To bardzo ważne. Dzisiaj apeluję z tego miejsca, aby cała Wysoka Izba poparła projekt pana prezydenta, abyśmy właśnie w tym duchu solidarności poparli rozwiązania, które proponuje pan prezydent.

Dzisiaj pada również pytanie w tym szczególnym dniu o solidarność, o solidarność 2020, jak ją możemy pojmować. To niewątpliwie wsparcie potrzebujących pomocy i empatia społeczna. To inwestycje, które zapewnią przyszłość kolejnym pokoleniom. To drogi, które ułatwią poruszanie się. Taką właśnie misję realizuje prezydent Andrzej Duda. Apeluję o to i zgłaszam wniosek w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania bez odsyłania prezydenckiego projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 do komisji. Popieramy w pełni ten projekt ustawy i wnosimy o jak najszybsze uchwalenie tego projektu. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Borys Budka. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Panie Ministrze! Cieszę się, że pan prezydent Andrzej Duda kolejny raz sięgnął do dobrych rozwiązań, które Koalicja Obywatelska proponowała już kilkanaście tygodni temu. Cieszę się, że pan prezydent Andrzej Duda wreszcie stara się zrozumieć, co to jest prawdziwa solidarność, bo przez ostatnie 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy słowo „solidarność” zostało wypaczone. Pan prezydent Andrzej Duda przedstawiał się jako człowiek, który przychodzi po to, by wsłuchiwać się w głos suwerena, a jedynym głosem, w który on się wsłuchiwał, to był głos prezesa z Nowogrodzkiej. Dzisiaj, gdy panikuje w obliczu sondaży, w obliczu tego, że Polacy mówią wyraźnie: mamy tego dość, prezentuje projekt ustawy, który jak w soczewce obrazuje wielką porażkę rządu premiera Morawieckiego. To właśnie pan premier Morawiecki obiecywał z tej mównicy, że żadne miejsce pracy nie zostanie utracone. Pan prezydent Andrzej Duda musi ratować to, co pan zepsuł. Tak, solidarność jest potrzebna, ale potrzebna jest nowa solidarność w nowych wyzwaniach. To nie ma być tylko coś na potrzeby kampanii wyborczej. Skorzystał pan prezydent i rząd Prawa i Sprawiedliwości z pomysłu Koalicji Obywatelskiej: 500+ na każde dziecko. Skorzystaliście przed wyborami europejskimi z trzynastej emerytury, oczywiście robiąc to po swojemu i wypaczając ideę. Teraz korzystacie z dobrego pomysłu Koalicji Obywatelskiej, tylko znowu robicie to za późno i niestety robicie to w zły sposób. Otóż jedynym celem, który przyświeca tej ustawie, jest cel wyborczy. Kiedy mówimy o solidarności, należy zapytać pana prezydenta: Czy jest pan solidarny z panem Szumowskim i jego rodziną? Gdzie był pana głos, kiedy media informowały o tym, w jaki sposób rodzina Szumowskich bogaciła się na majątku Skarbu Państwa? Gdzie pan był, panie prezydencie, chyba solidarnie z panem Banasiem, kiedy zarzuty, poważne zarzuty nie spowodowały, że pan premier wprowadził plan B? Pan Banaś nadal zajmuje swoje stanowisko. Gdzie pan był, panie prezydencie, gdzie była ta solidarność, kiedy krok po kroku ten rząd niszczył kolejne elementy życia publicznego? Gdzie pan był, panie prezydencie, kiedy była potrzebna solidarność z opiekunami osób niepełnosprawnych? Gdzie pan był, panie prezydencie, kiedy potrzebna była solidarność z nauczycielami, z pedagogami, z lekarzami, z tymi wszystkimi, którzy byli przez ten rząd obrażani i niszczeni? I wreszcie gdzie pan był, panie prezydencie, kiedy potrzebna była solidarność z polskimi pacjentami? Jest pan niewiarygodny. Obiecał pan, że Jacek Kurski zniknie z polskiej telewizji. Obiecał pan 2 mld zł dla polskich pacjentów. Kurski wrócił do TVP, bo pan wie doskonale, że bez Kurskiego nie ma pan żadnych szans w tej kampanii wyborczej. Ale ja panu mówię z tego miejsca, że z Kurskim czy bez Kurskiego pan już te wybory przegrał. I szkoda, panie prezydencie, że nie ma pana dzisiaj z nami. Szkoda, panie prezydencie, że po tych 5 latach prezydentury niesamodzielnej, prezydentury pod dyktando jednego człowieka z Nowogrodzkiej nie przyszedł pan do Wysokiej Izby, żeby spojrzeć nam prosto w oczy i powiedzieć: przepraszam. Powinien pan przeprosić za swoich partyjnych kolegów, którzy z polskiego państwa zrobili Bizancjum, którzy w sposób haniebny dorabiają się na krzywdzie innych, którzy nawet w czasach pandemii potrafili bogacić się kosztem polskich podatników. Pan, panie prezydencie, jest twarzą tej złej zmiany. Pan, panie prezydencie, firmuje wszystko to, co najgorsze w tym rządzie. Dzisiaj ten rząd rękami pana premiera Morawieckiego rozpaczliwie próbuje ratować pana kampanię, ale ona jest nie do odratowania.

Mamy dość. Mamy dość słabej prezydentury. Chcemy silnego prezydenta dla wspólnej Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Słuchaliśmy tutaj pana premiera, który właśnie odkłada komórkę, który mówił o tym, żeby nie wracać do rządów Platformy Obywatelskiej, do czasów, kiedy nikt nie dbał o ludzi, którzy tracili pracę, kiedy nikt nie dbał o tych, którzy byli wypchnięci na śmieciówki, żeby nie wracać do tych czasów, kiedy płaciło się 3,50 za godzinę. I, panie premierze, ja się z panem zgadzam, do tego nie należy wracać. To są błędy, których nie wolno powtórzyć. Jak rozumiem, ta ustawa to miał być dowód, że wy jesteście inni. I nie ma co ukrywać, rozbudziliście spore oczekiwania. Ja tutaj jakiś czas temu rozmawiałem na korytarzu z jednym z posłów PiS-u, który mi się odgrażał, że pokażecie tak prospołeczną ustawę, że nam w Razem kapcie pospadają, jak to ujął. Miała być jakaś bomba, miał być wielki game changer. No i cóż? No i ustawa leży na stole. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, ten podstawowy, ten, który bezrobotny dostanie po 3 miesiącach? Bo zgodzicie się państwo, że za Platformy ten zasiłek był skandalicznie niski, bo wynosił ledwo 36% płacy minimalnej, i za te pieniądze nie dało się żyć, prawda. No to ile teraz, panie premierze, dostanie bezrobotny od tego podobno prospołecznego rządu? Otóż policzyłem. Po tych 3 miesiącach dostanie ni mniej, ni więcej tylko 36% płacy minimalnej. Dokładnie tak samo jak za rządów liberałów. Więc miała być bomba, a wyszedł trochę kapiszon, wyszła z tego po prostu zwykła, trochę zaległa waloryzacja zasiłku. I jak patrzę na to puste krzesło tam na górze, które pan prezydent opuścił, to myślę sobie, że może nie przypadkiem je opuścił. Te pieniądze to było za mało za Tuska, pana ówczesnego szefa, i te pieniądze to jest za mało teraz. Zbyt niski zasiłek dla osób, które tracą pracę, to jest skazywanie ludzi na to, że nie będą mieli za co zapłacić czynszu, że nie będą mieli za co zrobić zakupów. A komuś, kto stracił pracę, trzeba realnie pomóc stanąć na nogi, a nie wpychać go w długi u lichwiarza. A tym właśnie skończy się wyznaczenie poziomu zasiłku dla bezrobotnych na zbyt niskim poziomie. To można było i trzeba było zrobić inaczej. Pokazywaliśmy wam zresztą, jak to zrobić. Tam to macie bardzo prosto i jasno przygotowane - normalny, europejski system pomocy dla osób bezrobotnych, z prostą zasadą, że świadczenie to jest połowa ostatniej pensji, tak jak to działa w wielu krajach Europy Zachodniej. Szczerze mówiąc, myślałem, że trzymacie coś naprawdę dużego, jakiś hit, że dlatego przetrzymujecie naszą ustawę w zamrażarce, bo przyniesiecie nam tutaj coś naprawdę lepszego. A teraz już wiemy, jak jest, i trzeba powiedzieć to otwarcie: szału nie ma. A jak go przepisujecie, to nie przepisujcie po kawałku, tylko weźcie w całości, bo jak przepisywaliście po kawałku, to przepisaliście z dziurami, bo w tej waszej ustawie o dodatku solidarnościowym jest cała grupa osób, które nic nie dostaną. Kto nie dostanie tego waszego dodatku solidarnościowego? Ludzie, którzy pracowali na śmieciówkach, bo oczywiście nie mają stosunku pracy. Ludzie, którzy szukali nowej pracy akurat po wybuchu epidemii. Myślę, że bardzo wielu mieszkańców Szydłowca, bardzo wielu mieszkańców Braniewa, tych miejsc, gdzie jest cały czas wysoki poziom strukturalnego bezrobocia, serdecznie wam podziękuje, kiedy się zorientują, że to wsparcie jest, owszem, ale nie dla nich. Wreszcie nie dostaną pieniędzy ludzie, którzy są na wymuszonych umowach za tzw. porozumieniem stron, które teraz, w realiach kryzysu, wyglądają tak, że pracodawca mówi: albo porozumienie, albo dostaniesz dyscyplinarkę. Więc ci ludzie nie dostaną, bo pan premier z panem prezydentem postanowili pobawić się w centusiów, chociaż to naprawdę nie jest czas na to, żeby mówić: ten bezrobotny zasługuje na pomoc, ten nie zasługuje, i nie wolno ludzi w ten sposób teraz tak traktować. To jest bardzo ciekawa część uzasadnienia tej ustawy, bo jak pan się zresztą wielokrotnie chwalił, panie premierze, bardzo szybko przeznaczyliście dziesiątki miliardów złotych na pomoc dla pana przyjaciół z sektora finansowego i dla wielkiego biznesu, a tutaj zasiłki dla bezrobotnych - po 3 miesiącach, ponaglani przez Lewicę, z wiszącym poselskim projektem ustawy, ostatecznie wyskrobaliście na ten cel, jak piszecie, 490 mln zł. Pani minister się ze zdziwieniem przypatruje uzasadnieniu, które wyszło, jak rozumiem, z jej ministerstwa, zanim podpisał je pan prezydent. Tyle właśnie przeznaczacie na zasiłki. No to są naprawdę nieporównywalne pieniądze z tymi, które przeznaczyliście na pomoc dla biznesu. Szanowni Państwo! Koalicyjny klub Lewicy poprze oczywiście każdą podwyżkę świadczeń dla osób, które tracą dziś pracę, ale chcę powiedzieć jasno: ta ustawa nie rozwiązuje tych problemów. Jeżeli bezrobocie będzie rosnąć tak, jak mówią prognozy, to jesienią, panie ministrze Kowalczyk, sami się o tym przekonacie. będziecie musieli jesienią wrócić do projektu ustawy przedstawionego przez Lewicę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Panie Ministrze!

Panie Ministrze! Panie Premierze! Państwo Posłowie! Ujmując rzecz precyzyjnie, bardziej precyzyjnie, one straciły pracę na skutek decyzji podjętej przez rząd w dwóch albo nawet i trzech, bo była jeszcze nowelizacja, zarządzeniach wydanych przez ministra zdrowia, za zgodą całego rządu, ogłaszanych wspólnie z premierem, z 13 i 20 marca, o ograniczeniu albo wręcz zakazie prowadzenia konkretnych działalności gospodarczych. Nie twierdzę z tego miejsca, że te decyzje były bezzasadne, ale to była bezpośrednia przyczyna, dla której ci ludzie tracili zatrudnienie, dotychczasowe zatrudnienie, dotychczasowe miejsca pracy, ponieważ ich pracodawcy, ich przedsiębiorstwa nie miały możliwości operacyjnego działania albo było one ograniczone do minimum decyzją rządu. Dlaczego przywołuję tę okoliczność?

Czy naprawdę tak nisko traktujecie Polaków, że uważacie, iż wtedy kiedy tracili pracę, to nawet nie zarabiali minimalnej pensji? To znaczy, że wielka nieufność i wielki brak szacunku dla pracodawców i pracowników przebija z waszych wystąpień, z waszej polityki i z waszych projektów. Ci ludzie zarabiali, gwarantuję wam, co najmniej minimalną pensję, a pewnie więcej. A więc ogłaszana z takim przytupem propozycja dodatku solidarnościowego jest niczym więcej jak tylko jałmużną i do tego jałmużną, która budzi oburzenie również z tego powodu, ile czasu zajęło przygotowanie dosyć prostego projektu ustawy panu prezydentowi, jak rozumiem, we współpracy z rządem. W tym czasie przygotowano cztery wersje tarczy antykryzysowej. Rząd w tych tarczach zdążył zadbać o zwolnienie z odpowiedzialności karnej urzędników państwowych kupujących maseczki albo przyłbice od znajomych, ewentualnie firm kogucik, ale zawsze po wyższej cenie. Rząd zdążył zapewnić czy ograniczyć kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w organizacji uczciwych, transparentnych wyborów prezydenckich, ale przez te prawie 3 miesiące o bezrobotnych, nowych bezrobotnych, którzy stracili pracę na skutek rządowych decyzji, jakoś nie pamiętał. A przecież 1 maja, 5 tygodni temu, pan prezydent Duda również z przytupem ogłaszał ten dodatek na swojej tzw. konwencji programowej. Co się stało, że ten projekt wpływa dopiero teraz, na początku czerwca, mimo że był z takim hukiem ogłaszany 1 maja? Wiemy, co się stało. Przesunięto termin wyborów prezydenckich. A więc z tego miejsca oskarżam również prezydenta Andrzeja Dudę, że grał strachem, stresem i niepokojem osób, które straciły pracę już w połowie marca albo najpóźniej z dniem 1 kwietnia i które stanęły wobec ryzyka braku możliwości spłaty kredytów albo nawet opłaty czynszu mieszkalnego, zwyczajnie rzecz biorąc, być może zakupu w

Ale nasz klub mimo wszystkich zastrzeżeń będzie za dalszymi pracami nad tym projektem, bo jest tam kilka rozwiązań sensownych, w tym również rozwiązanie mówiące o tym, że dodatek solidarnościowy będzie wypłacany bez potrącania podatków. Otóż to jest droga, którą od dawna proponujemy. Emerytura bez podatku, panie premierze, emerytura bez podatku, panie ministrze Kancelarii Prezydenta. Śmiało, skoro robicie już pierwszy krok, ażeby naprawdę zwolnić obywateli w potrzebie, polskich obywateli będących w potrzebie, w tym również emerytów, to idźcie dalej, przyjmijcie nasz projekt (Dzwonek), który powtórnie w tej kadencji był złożony do laski marszałkowskiej i czeka na waszą pozytywną decyzję. Dziękuję bardzo. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Jakub Kulesza. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Nie ma? Szkoda, bo mam dla pana prezydenta cytat: Amerykańska demokracja przetrwa do czasu, kiedy Kongres odkryje, że można przekupić społeczeństwo za publiczne pieniądze. Kilka dni przed wyborami samorządowymi w 2018 r. została wypłacona wyprawka+, kilka dni przed wyborami europarlamentarnymi w 2019 r. została wypłacona trzynasta emerytura, kilka dni przed wyborami parlamentarnymi - majstersztyk, kumulacja, 1500 zł zaległych za 3 miesiące 500+ na pierwsze dziecko.

Zastanawiałem się, co będzie kolejne. Pan, panie prezydencie, doskonale wie, że rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko pieniądze zagrabione kolejnymi podatkami, ale wymyślił pan dodatek solidarnościowy właśnie po to, żeby, tak jak na targu w Garwolinie kilka dni temu, mógł pan kłamać, że to pan sam daje trzynastą emeryturę, 500+, wyprawkę, dodatek, a te ustawy o opłatach za śmieci, te 34 podwyżki podatków to nie pan - oczywiście pan te ustawy podpisał - tylko to opozycja. To jest dodatek do dalszej likwidacji miejsc pracy, którą zafundował nam pana kolega z nart - minister „nie nosić maseczek” Szumowski. Ten dodatek tak naprawdę tylko pogłębi problem bezrobocia. Panie prezydencie, ta propozycja to jest moim zdaniem dyletanctwo ekonomiczne. Pan nie rozumie, jak działa gospodarka i skąd się biorą publiczne pieniądze. Jeśli chce pan, żeby w osłabionej waszymi restrykcjami gospodarce pracodawcom opłacało się zatrudniać, a pracownikom opłacało się pracować, to proszę zrealizować swoją obietnicę sprzed 5 lat i podnieść kwotę wolną od podatku, np. tak jak proponuje Konfederacja, do 30 tys. zł rocznie albo najlepiej do dwunastokrotności pensji minimalnej. Natomiast ten dodatek solidarnościowy to zachęta do kolejnych zwolnień i do przechodzenia do pracy na czarno. Na przykład wiele podmiotów na rynku działa w powiązanych kapitałowo grupach i osobowych grupach i w takiej grupie nie ma problemu, by w jednej spółce zwolnić pracownika, a w drugiej go zatrudnić i na odwrót. Co więcej, to jest świadczenie 1400 zł przez 3 miesiące. Dotyczy nie tylko zwolnionych, ale tych, którym po prostu wygasła umowa o pracę po 31 marca. Wiele osób ma niezależną od COVID-19 pracę sezonową i taki urlop akurat, np. na uczelniach, im wypada. Jeśli w jakiejś rodzinnej firmie pracodawca zastanawiał się, nie chciał zwalniać pracownika, to ten dodatek właśnie go do tego zachęci. Chciałbym, panie prezydencie, żeby pan sobie wpoił inny cytat, tym razem Miltona Friedmana: Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują, a każecie im płacić podatki, gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jeśli dopłacamy do fotowoltaiki albo wiatraków, to w jakim celu to robimy? Weźmy taki właśnie przykład. Domyślam się, że robimy to w tym celu, że spodziewamy się, że dzięki temu będzie więcej wiatraków i więcej paneli słonecznych. Niezależnie, czy to jest słuszna decyzja czy nie, ale taka jest zapewne intencja takich działań. No to w jakim celu dopłacamy teraz do bezrobocia? Rozumiem, że chcemy mieć więcej bezrobocia, tak?

W dodatku podnosimy te zasiłki w sytuacji, kiedy szczególnie nas na nie nie stać, kiedy wielu osobom obniżono pensję itd. W tej sytuacji tym bardziej nie będzie opłacało się znajdywać pracy, bo ten, kto znajdzie pracę, przeskoczy jednym susem do grona tych, którzy będą musieli płacić na pozostałych. Więc wydajecie miliardy w ramach różnych programów pomocowych na promocję zatrudnienia, a teraz robicie coś dokładnie odwrotnego.

Solidarność jest wtedy, kiedy ktoś się dobrowolnie solidaryzuje, a kiedy przystawiamy komuś pistolet do głowy i mówimy: teraz ty, burżuju, [[Dzwonek]] solidaryzuj mi się natychmiast z tym drugim, biednym - to to nie jest żadna solidarność, tylko to jest rabunek i napaść. bo będziemy utrzymywać tutaj cudzoziemców.

Wyznaczam czas - 1 minuta. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! 5 lat, panie prezydencie, miał pan 5 lat na to, żeby zrealizować swoje obietnice wyborcze. Zrobił pan to? Gdzie jest pomoc dla frankowiczów? Nie ma. Gdzie jest 100 tys. tanich mieszkań? Nie ma. Gdzie jest emerytura bez podatku? Nie ma. Gdzie są zamówienia dla PZL Świdnik, które pan obiecywał, będąc na Lubelszczyźnie? Nie ma. A teraz, 3 tygodnie przed wyborami, składa pan projekt ustawy, którą się obecnie zajmujemy. Składa go pan w dniu, w którym marszałek Sejmu ogłasza i zarządza wybory prezydenckie. Liczy pan na to, że w ostatniej chwili uratuje pan swoją prezydenturę. Zamiast zaproponować projekt ustawy, który by w sposób długofalowy rozwiązywał problemy osób zwalnianych z pracy, proponuje pan 1400 zł, ale tylko do zakończenia swojej kadencji. Im nie proponuje pan nic. Proszę nie liczyć na to, że przekupi pan. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Zastanówmy się, czy te 1400 zł, które dostaną zwolnieni z pracy, nie obróci się przeciwko nim, dlatego że pracodawcy mogą nie mieć już motywacji do walki o zachowanie miejsc pracy. Pomyślmy, czy tak wysokie zasiłki paradoksalnie nie utrwalą bezrobocia. A z drugiej strony te 1400 zł jest tylko na 3 miesiące, dziwnym trafem do końca kadencji obecnego prezydenta. A co będzie później? Może oprócz zasiłku państwo powinno tworzyć nowe miejsca pracy? Bo przecież po koronawirusie nic już nie będzie takie samo i trzeba będzie jakoś się w tym nowym świecie odnaleźć. Pomyślmy o tym. Bardzo proszę. Panie i Panowie Posłowie! Pani Marszałek! Ani dodatek, ani solidarnościowy. Nie jest to dodatek, bo jest to zamiast zasiłku dla bezrobotnych. Oczywiście my też postulowaliśmy to, że wobec pandemii należałoby zwiększyć trochę zasiłek dla bezrobotnych, bo jest dramatycznie niski. Natomiast zauważmy jedną rzecz. Osoba, która dostanie ten zasiłek, który nazwaliście dodatkiem, nie dostanie podstawowego zasiłku. W związku z tym nazwa „dodatek” jest zwykłym oszustwem. Jedyna solidarność, którą ja tu widzę, to solidarność z panem prezydentem Andrzejem Dudą, w tym znaczeniu, że rozumiem, że rząd powiedział tak: Nie mogę zwiększyć kwoty wolnej, którą obiecałeś - trudno. Nie możemy przewalutować kredytów dla frankowiczów - nie da się. To zrobimy dodatek solidarnościowy na 3 miesiące, nazwiemy zasiłek dla bezrobotnych dodatkiem solidarnościowym i powiemy, że to twoja inicjatywa. No i to jest takie właśnie dokładnie oszustwo wyborcze. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja myślę sobie, że taką największą hipokryzją i oszustwem tej ustawy to jest nazywanie zastąpienia dodatku czy zasiłku dla bezrobotnych jakimś rodzajem solidarności z tymi, którzy mają trudności. Panie prezydencie, a może by pan pomyślał o solidarności z obywatelami w jakiś inny sposób? Od początku pana prezydentury rosną niesamowicie wydatki na pańską kancelarię. W tej chwili wysokość utrzymania pana i pańskiego dworu jest równa utrzymaniu dworu brytyjskiego. Tyle tylko, że jak porównują to media, statystyczny Brytyjczyk na swój dwór wydaje dwa razy mniej niż Polak. Nie mówiąc już o tym, że dwór hiszpański kosztuje pięć razy mniej niż pański dwór. Może by wykazać się solidarnością (Dzwonek) w ten sposób, żeby zrezygnować ze złotych piór. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Prezydencie! Pańska ustawa nie powinna nazywać się ustawą solidarnościową, tylko ustawą wyborczą. Gdzie pan był przez ostatnich 5 lat? Gdzie są rezultaty pańskich obietnic? Gdzie jest kwota wolna od podatku w wysokości 8 tys. zł? Nie ma. Gdzie jest pomoc dla frankowiczów? Nie ma. Gdzie są mieszkania, te 100 tys. mieszkań dla młodych Polaków, które obiecaliście? Pamiętam, jak w Szczecinie, obok stoczni mówił pan, że będą budowane statki, a Polska będzie światową potęgą. Niech pan pojedzie do stoczni i zobaczy, jak rdzewieje stępka. Nie ma żadnych efektów pańskich działań. Natomiast co jest? Propozycja programu oczko wodne+. Panie Prezydencie! Młodzi Polacy mają dzisiaj inne oczekiwania i inne problemy. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pana prezydenta nie ma, ale może pan przekaże. Słowo „solidarność”, odmieniane dzisiaj przez wiele przypadków, jest potrzebne panu prezydentowi, rozumiem, na potrzeby kampanii wyborczej. Chcę zapytać o jedno.

Pytam: Do kiedy słowo „solidarność” będzie przez państwa tak wykorzystywane? Kiedy jest kampania wyborcza? Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie zada pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Nie ma. A więc pani poseł Magdalena Biejat, Lewica. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Trzeba mieć dzisiaj nie lada szczęście, żeby zakwalifikować się do zasiłku dla bezrobotnych. W tej chwili pobiera go mniej niż 20% osób przebywających na bezrobociu. Ale te absurdalne kryteria, które trzeba spełnić, żeby zyskać ten zasiłek, to jest nic w porównaniu z kryteriami, które należy spełnić, żeby zyskać dodatek solidarnościowy. Ten dodatek będzie przysługiwać tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, tylko osobom, które zatrudnione były na tę umowę o pracę przez minimum 90 dni w 2020 r., i tylko tym osobom, które straciły pracę po 31 marca 2020 r. To nie jest żaden dodatek solidarnościowy, tylko mechanizm segregowania pracowników w samym środku najgorszego kryzysu od lat. Jeśli to jest wizytówka prezydentury Andrzeja Dudy, to nie najlepiej to świadczy o tej prezydenturze. Dlatego mam pytanie do pana ministra Muchy, bo brak jest pana prezydenta: Dlaczego dzielicie pracowników na lepszych i gorszych? Dziękuję. Bardzo proszę. Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Do tej pory, mimo że w wyniku epidemii pracę już teraz tracą tysiące osób, władze konsekwentnie odrzucały propozycję pomocy bezrobotnym. W kolejnych tarczach antykryzysowych nie pojawiało się nawet słowo „bezrobotny” Czy wszystko tylko po to, żeby w trakcie kampanii prezydenckiej prezydent Andrzej Duda mógł przedstawić swoją propozycję? Po pierwsze, jest to robione z olbrzymim opóźnieniem. Po drugie, z wielkich obietnic prezydenta został nam wzrost bazowego zasiłku o 200 zł. Oczywiście lepsze to niż nic, ale to ciągle zdecydowanie za mało, chyba że czekamy na rozwój kampanii i na kolejne prezydenckie dodatki. Jeżeli tak, to w Sejmie już od dawna czeka gotowy projekt Lewicy, który zakłada to, o czym mówi prezydent: prawdziwą podwyżkę zasiłku na stałe oraz specjalne świadczenie dla tych, którzy dziś przez epidemię nawet nie mają szansy szukać pracy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Monika Falej, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dopiero pan premier mówił, jak świetnie sobie rząd poradził z epidemią, a tu taka niespodzianka, prezydent składa projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, który z dnia na dzień jest procedowany. Projekt Lewicy leży od kilku tygodni i niestety nie ma takiej możliwości ani takiego szczęścia. Rozumiem zatem, że rząd jednak sobie nie poradził i stąd taka wrzutka. Tylko pytanie: Pomocna dłoń dla obywateli, dla rządu czy dla kandydata Dudy? Bo sam dodatek ma być świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące i tylko na okres od 1 czerwca do końca sierpnia. Mógłby pan wyjaśnić, skąd te ograniczenia? Ograniczenie czerwiec-sierpień spowoduje, że duża liczba osób pozostających bez pracy z tego dodatku nie skorzysta, skorzysta natomiast pan prezydent. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Anita Sowińska, klub Lewica. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! Ta ustawa to jest nieudolna próba naśladownictwa propozycji Lewicy. Panie prezydencie, ośmiesza się pan tą ustawą, po raz kolejny zresztą. To tak, jakby zamiast jabłka, które zaproponowała Lewica, pan dawał ludziom ogryzek. Żałuję, że nie ma pana tutaj z nami, ponieważ chciałam powiedzieć panu prosto w oczy, że jest pan najgorszym prezydentem w ciągu ostatnich 30 lat. Przez ostatnie 5 lat nie dał pan żadnej wartości dodanej Polkom i Polakom. Podpisywał pan wszystko, co panu podsunęli. Nie potrafił pan podejmować samodzielnych decyzji. Nawet nie stać pana było na własne zdanie i powtarzał pan tylko PiS-owskie przekazy dnia. Szkoda naszego czasu. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan prezydent zafundował sobie dzisiaj na koszt podatników kampanię wyborczą w Sejmie. Ale, jak rozumiem, prezydent ma takie prawo i zawsze może, nawet tuż przed wyborami, z tego prawa skorzystać.

Przyznam trochę ironicznie, że pan prezydent zamierza bardzo tanim kosztem kupić sobie głosy w przeddzień wyborów. Przecież wiadomo, że koronawirus nie zniknie za pomocą czarodziejskiej różdżki 31 sierpnia, a zakłady pracy nie podniosą się do tego czasu. Moim zdaniem, i myślę, że zdaniem wielu Polaków, jest to bardzo populistyczne, wyborcze manipulowanie Polakami. Mam pytanie: Czy na tym kończy się pana pomoc dla ofiar COVID-19 i czy już zapomniał pan o tym, że na jesieni (Dzwonek) przewidywana jest kolejna fala zachorowań? Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pan premier zadał dzisiaj pytanie, czyja będzie Polska. A ja chciałbym zadać pytanie, jaka będzie Polska i z kim będzie solidarna. Czy będzie solidarna z najsłabszymi, z tymi, którzy potrzebują podania pomocnej dłoni, czy będzie solidarna z rodziną Szumowskich, tak jak to ma miejsce od 4 lat?

Szanowni Państwo! Kolejna sprawa to jest sprawa zakupów Ministerstwa Zdrowia. Z tej opcji nie skorzystano. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek Czcigodna! Wysoka Pustawa Izbo!

Z drugiej strony to jest tak jawnie korupcyjny projekt, to jest tak jawne szalbierstwo, bardzo dobrze wypunktowane przez szanowne koleżanki i kolegów, moich przedmówców. No i rozdarci między tymi dwoma skrzydłami zdecydowaliśmy, że nie będziemy wnioskowali o odrzucenie tego projektu, żeby się nad nim jeszcze poznęcać w następnych czytaniach. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja, łączy się zdalnie. Szanowna Pani Marszałek! Panie Prezydencie! Nie ulega wątpliwości, że pan prezydent Duda będzie obiecywał, będzie sypał z worka i twierdził, że to on dał Polakom pieniądze, co jak wiemy - nie jest prawdą. Byłbym nawet w stanie zgodzić się z samą zasadnością tego projektu, ponieważ jest on skierowany do osób, które często niezależnie od swojej winy zostały pokrzywdzone. Natomiast chciałbym się też już bardziej konkretnie odnieść do jednej rzeczy.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na początku maja podczas konwencji wyborczej pan prezydent Andrzej Duda ogłosił pomoc dla tracących pracę przez pandemię. Pracował nad tą ustawą przeszło miesiąc. Ale wtedy powiedział, cytuję: zasiłek dla bezrobotnych musi zostać podniesiony do 1300 zł i być przeznaczony dla wszystkich, którzy stracili pracę z powodu koronawirusa. Ale musi być jeszcze dodatkowa formuła wsparcia, coś, co nazywam dodatkiem solidarnościowym. Ten dodatek to 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę w wyniku kryzysu spowodowanego koronawirusem. Panie Ministrze! To jak? To gdzie jest... 1300 zł i 1200 zł to jest 2500 zł przez 3 miesiące.

Bardzo proszę.

Chciałem zwrócić się do pani minister z pytaniem, czy istnieje możliwość prolongaty wypłaty z tego funduszu poza ten 3-miesięczny okres, bo wtedy jest zapowiedź zwiększenia wysokości zasiłku.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szkoda, że nie ma dzisiaj z nami pana prezydenta.

Ale już podchodząc poważnie. Panie ministrze, lepiej późno niż wcale, tylko gdzie był pan, panie prezydencie, kiedy. Pewnie pan wiedział, że te zwolnienia się rozpoczną. Myślę, że to jest przede wszystkim inicjatywa spóźniona. Tutaj ponownie, jak mój kolega klubowy, zaapeluję, bo jednak 3 miesiące to chyba jest za krótki czas i chyba jedynie pan prezydent wie, że kryzys w Polsce się skończy. I życzyłbym sobie, żeby tak było, ale nie wiem, czy tak będzie. Panie premierze, obawiam się, że pan prezydent obnaży dziury w pana tarczy. Jeżeli chodzi o skutki finansowe dla budżetu, panie ministrze, wydaje mi się, chciałbym podać.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym rozpocząć od apelu, bo przecież wiemy, że trwa kampania wyborcza i wszyscy tutaj, na tej sali, i po prawej, i po lewej stronie, mamy przeświadczenie, że ten projekt ustawy jest elementem tejże kampanii. Mam apel do pana ministra, którego znam tyle lat, o to, żeby jednak podyskutować poważnie nad tym projektem i żeby rzeczywiście pochylić się nad projektem Lewicy, czyli nad tym dokumentem, projektem ustawy o świadczeniu kryzysowym, bo być może będzie pole do tego, ażeby podyskutować o grupie osób, których ma dotyczyć to świadczenie, żeby podyskutować o terminie wypłacania tego świadczenia, żeby podyskutować o rzeczach i problemach, które tu są, bo oprócz kampanii kluczem jest to, żebyśmy pomogli ludziom. Czy macie państwo te koszty wyliczone?

Zapraszam. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Myślę, że nie wszyscy doczytali tę ustawę, bo tak naprawdę drugą częścią tej ustawy jest podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł - i to jest permanentny, można by powiedzieć, dodatek solidarnościowy, troszeczkę mniejszy, o 200 zł. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście bezrobocie w Polsce rośnie bardzo powoli. To jest ogromna zasługa bardzo skutecznej tarczy finansowej, różnego rodzaju działań: ZUS-u, pożyczek z Funduszu Pracy - 5 tys., tarczy realizowanej przez PFR. Ale jednak zdarzają się przypadki zwolnień i to właśnie te przypadki zwolnień, utraty pracy zauważa pan prezydent - i wielka chwała, i wielkie podziękowania za to. Natomiast ja mam takie pytanie do pani minister Maląg i wnioskodawców, pana ministra Muchy.

Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na postawione pytania w pierwszej kolejności odpowie minister rodziny, pracy i polityki społecznej pani Marlena Maląg. Zapraszam.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ostatnie 5 lat to dobry czas dla Polski i ten dobry czas dla Polski i dla polskich rodzin rozpoczął nie kto inny, tylko pan prezydent Andrzej Duda. Działania wprowadzone przez pana prezydenta, zapoczątkowanie Polski+, świadczenie „Rodzina 500+”, „Dobry start”, trzynasta emerytura, obniżenie wieku emerytalnego, waloryzacja świadczeń emerytalnych na godziwym poziomie to właśnie troska o polskie rodziny. I w tym momencie, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, również pan prezydent, właśnie we współpracy z rządem, zapowiada i wprowadza konkretne rozwiązania, to, co pan prezydent pokazał właśnie w swojej 5-letniej kadencji. Ja przypomnę, bo państwo tutaj wielokrotnie powtarzacie słowa o ochronie miejsc pracy, o tym, jak pracownicy nie są chronieni. Od 1 kwietnia, teraz są to 2 miesiące - podsumowujemy działanie tarcz, które zostały wdrożone - realne pieniądze, które zostały przekazane dla pracodawców i pracowników na ochronę ich miejsc pracy, a więc na wypłaty wynagrodzeń, bo pracodawcy i pracownicy to jest jedna całość, to jest naczynie powiązane, to ponad 73,5 mld zł. Odnosząc się do ustawy, którą dzisiaj zaproponował pan prezydent, a zapowiedział ją 1 maja tego roku: tak naprawdę wszystkie mechanizmy, wszystkie instrumenty, które były wprowadzane przez rząd, przede wszystkim służą i służyć będą ochronie miejsc pracy. Cały czas zapowiadaliśmy, że analizujemy sytuację na rynku pracy, pokazujemy, jak ta sytuacja wygląda, i pan prezydent zaproponował dobrą ustawę. Natomiast dobrze byłoby, żebyście państwo tę ustawę dobrze przeczytali.

A więc o nikim nie zapomniano, każda grupa została zabezpieczona. Szanowni państwo, dodatek solidarnościowy 1400 zł to chyba jest więcej niż połowa płacy minimalnej. Ale pan prezydent pamięta także o tym, że od września zasiłek dla bezrobotnych proponuje w wysokości 1200 zł.

Odniosę się do ustawy, która została przedstawiona przez klub Lewicy. Szanowni państwo, państwo proponujecie, żeby realizowały to powiatowe urzędy pracy. Mechanizm jest tak skomplikowany, że kiedy świadczenie byłoby rzeczywiście wypłacone, trudno powiedzieć.

Warto powtarzać, pokazać, jak sprawnie działa ZUS. Dzisiaj świadczenia postojowe, a także zawieszenie składki ZUS-owskiej jest realizowane na poziomie 98%. Natomiast niektóre powiatowe urzędy pracy. Myślę, że warto wspomnieć, że również powiatowy urząd pracy nadzorowany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego na wczoraj miał wykonanie 32%. Średnia z wszystkich mechanizmów, z których (Dzwonek) wsparcie jest przekazywane przede wszystkim na ochronę miejsc pracy, jest ok. 80%. ZUS jest też gwarantem tego, że osoby, które tego świadczenia potrzebują, to świadczenie będą miały jak najszybciej wypłacone. Dlatego też ustawa, która została zaproponowana przez pana prezydenta, jest głęboko przemyślana, jest łatwym instrumentem do wdrożenia i właśnie pokazania, że w ciągu kilku dni od wejścia w życie ustawy osoby objęte tym wsparciem będą miały świadczenie wypłacone.

Zawsze powtarzamy, że analizujemy sytuację.

Dlatego też, szanowni państwo, właśnie dobra współpraca rządu z panem prezydentem, panem prezydentem Andrzejem Dudą, pokazuje skuteczność działania, pokazuje wsparcie, które szerokim strumieniem. My jesteśmy w trudnej sytuacji, w której staramy się przede wszystkim jak najbardziej łagodzić skutki, aby rodziny. Również ta ustawa zabezpiecza polskie rodziny. Dziękuję bardzo, pani minister. Pół minuty, panie pośle. Pani minister powiedziała, że osoby na śmieciówkach zostały objęte postojowym. W odległości 3 m od pani siedzi pan minister Szwed, który na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych potwierdził, że to, co mówią Lewica i związki zawodowe o ludziach, którzy teoretycznie mają to uprawnienie, ale nie dostają go, bo uniemożliwiliście im bezpośrednie składanie samodzielnie wniosków, jest realnym problemem. Więc proszę nie mówić, że ludzie mają dostęp do postojowego. Proszę posłuchać związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego. Złożyliśmy poprawkę w tej sprawie.

Dziękuję, panie pośle. Na pytania odpowie również w imieniu wnioskodawców zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan minister Paweł Mucha. Dziękuję bardzo zarówno za wypowiedzi państwa posłów zawarte w oświadczeniach złożonych w imieniu klubów i koła poselskiego, jak i za zapytania, które państwo zgłosiliście do tej dyskusji. Warto przede wszystkim mówić o tym, że ta ustawa dzisiaj poprawia sytuację prawną tych wszystkich, którzy nie mają świadczenia, a uzyskują 1400 zł netto. Wbrew temu, co tutaj padało w wypowiedziach, te 1400 zł netto jest kierowane także do tych, którzy są dzisiaj uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Tak jak mówiłem, w ogromnej większości to są też osoby, które dzisiaj tego wsparcia od Wysokiej Izby oczekują, i te pieniądze trafiają z uwagi na to, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej taki projekt przedkłada, a państwo, mam nadzieję, sprawnie nad nim będziecie procedować. A w perspektywie jest podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1200 zł, więc nie możemy mówić o tym, że ta pomoc nie jest pomocą adekwatną, nie jest pomocą na czasie, ona jest dzisiaj bardzo potrzebna i jest taką pomocą, która wynika z pogłębionej analizy. To jest dobra ustawa, to jest ustawa, nad którą trwały prace ekspertów, to jest ustawa, która była konsultowana ze środowiskiem społecznym. Najlepszym podsumowaniem jest to, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w tych pracach uczestniczył, poparł tę ustawę.

Tu strona społeczna wypowiedziała się za siebie i dla mnie nie ulega wątpliwości, że te rozwiązania są trafne. Dziękuję bardzo za wypowiedź: czyny nie słowa. Pan prezydent Andrzej Duda wykonuje swój urząd. Pan prezydent Andrzej Duda jest urzędującym prezydentem, który podejmuje problemy związane ze zdrowiem publicznym, współpracując z rządem pana premiera Mateusza Morawieckiego, współpracując z Ministerstwem Zdrowia, z głównym inspektorem sanitarnym. Pan prezydent Andrzej Duda skupia się na kwestiach konsekwencji społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. To są chociażby tego rodzaju rozwiązania jak wypracowane wspólnie z rządem zwolnienie z ZUS-u dla przedsiębiorców. To są sytuacje związane z wakacjami kredytowymi, to są rozwiązania dotyczące objęcia pomocą także rolników, którzy są w systemie KRUS-u. I naprawdę trzeba mieć bardzo dużo złej woli, żeby stwierdzić, że ten projekt jest projektem kampanijnym. Dzisiaj zadaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie swoich obowiązków w warunkach światowej pandemii, w warunkach takich, kiedy walczymy z COVID-19. Prezydent podejmuje te wyzwania i stąd przedkłada tego rodzaju rozwiązania prawne, które mają służyć pomocą 0,5 mln Polaków.

Dzisiaj miliony Polaków popierają jego program, bo to jest autentyczna bliskość ludzi, to jest ta wrażliwość, która sprawia, że prezydent umie rozmawiać z ludźmi, i z tej rozmowy z ludźmi rodzą się też tego rodzaju projekty, jak to rozwiązanie szczególne. Mam poczucie niedosytu po wystąpieniu pana przewodniczącego Budki, który wykrzyczał, jakby jednoosobowo był suwerenem, że pan prezydent czy przegrał, czy wygrał wybory. Chciałbym powiedzieć panu przewodniczącemu Budce bardzo wyraźnie: to naród decyduje, wyborcy rozstrzygają w wyborach powszechnych i będzie to rozstrzygniecie, natomiast nie jednoosobowo pan przewodniczący Budka, który nie jest zainteresowany, jak widzę, dyskusją w tej sprawie. Bardzo ubolewam nad tym, że jeden z posłów mieniących się liderem opozycji nie chce rozmawiać merytorycznie, tylko wygłosił w tej sprawie bardzo polityczne stanowisko. Ja wskażę, że świadczenie postojowe to jest rozwiązanie prawne, które zostało tu zgłoszone. Państwo macie też świadomość co do swojego projektu, krytycznej opinii Związku Powiatów Polskich, bardzo wyraźnie wyrażonej, i macie też świadomość tego, że szereg rozwiązań prawnych, które zostały przyjęte w toku tarczy antykryzysowych, skonsumowało część tych propozycji.

Takie wypowiedzi nie powinny mieć miejsca - i mówię to, patrząc w oczy pana przewodniczącego Zandberga. Rozmawiajmy ze sobą merytorycznie, a wypowiedzi tego rodzaju, jak jedna z tych, które tu miały miejsce, są urągające wszelkim standardom. Jeżeli chodzi o kwestie zwolnienia z podatku, mówiłem o tym, przedstawiając projekt. Absolutnie nie zgadzam się z tymi głosami, które padły ze strony posłów Konfederacji, które mówią o negatywnych skutkach tej ustawy.

Co do pytań szczegółowych, w tym przypadku merytorycznych nie było zbyt wiele, pojawiła się zupełnie fałszywa teza, jakoby rząd odpowiadał za COVID-19 albo pan prezydent odpowiadał za COVID-19. Szanowni państwo, COVID-19 jest zjawiskiem obiektywnym, jest pandemią światową i z tymi konsekwencjami COVID-u, które występują, walczymy, minimalizując negatywne skutki COVID-u, a wiemy, że tym wyzwaniem poza zdrowiem publicznym są także konsekwencje gospodarcze. Więc miejsca pracy w Polsce, które zostały stracone, są dzisiaj stracone przez COVID, a nie przez działania rządu. Odwrotnie: działania rządu powodują, że ten ubytek miejsc pracy nie jest tak wielki, jak można było się spodziewać wtedy, kiedy pandemia się rozwijała i kiedy wszyscy byliśmy pełni obaw. Pani minister mówiła też o tym bardzo wyraźnie, że głównym zadaniem, które stawiają sobie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i polski rząd, jest właśnie ochrona miejsc pracy, jest wsparcie polskich przedsiębiorców, są środki dla polskich przedsiębiorców. To jest dostrzeżenie pewnej obiektywnej potrzeby. Z jednej strony robimy wszystko, żeby miejsc pracy bronić, żeby wspierać polskich przedsiębiorców, ale mamy też świadomość obiektywnej sytuacji, tych miejsc pracy, które zostały zlikwidowane, tych osób, które są bez prawa do zasiłku, i tych osób, które są bezrobotne. I stąd zgłoszenie tej ustawy, nad którą prace trwały około miesiąca i były to prace merytoryczne. No, szanowni państwo, bardzo długo mógłbym mówić o tym, jak wiele dobrego udało się zrobić w ciągu ostatnich 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy, dzięki dobrej współpracy większości parlamentarnej, rządów pani premier Beaty Szydło i pana premiera Mateusza Morawieckiego, który dzisiaj uzyskał wotum zaufania ze strony Wysokiej Izby, właśnie przez to, że jest ta szczególna wrażliwość społeczna.

Oczywiście, że mamy wsparcie dla kredytobiorców.

W ogóle dokonano wielu zmian w podatkach, wielokrotnie mówili o tym przedstawiciele rządu. Do pana posła Marchewki, który też nie jest zainteresowany, jak widzę, odpowiedzią na pytanie, które zadał. Była tutaj mowa o Pomorzu Zachodnim. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wspierał inwestycje takie jak rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, takie inwestycje jak budowa tunelu pod Świną, takie inwestycje jak bloki gazowe, największa dzisiaj tego typu inwestycja w Europie, w Zespole Elektrowni Dolna Odra. To jest prezydent, który dotrzymuje słowa, który dba o zrównoważony rozwój całej Polski, i to jest prezydent, który dostrzega także Pomorze Zachodnie, angażuje się w procesy inwestycyjne, wspiera te procesy na bieżąco. Tak więc tyle odpowiedzi na to pytanie. Była mowa o tym, mówiła też już o tym pani minister, czy wobec sytuacji na rynku pracy istnieje możliwość przedłużenia wypłacania dodatku solidarnościowego. Tak, wprost o tym stanowi przepis art. 4 ust. 5 ustawy, że Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres przysługiwania dodatku solidarnościowego. Mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie. Jestem przekonany, że te działania, które są podejmowane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i rząd Prawa i Sprawiedliwości, służą temu, żebyśmy jak najszybciej wyszli z kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19.

Bardzo się cieszę z tego, że tutaj padł taki głos, bo to było oczekiwanie Kancelarii Prezydenta i rozmawialiśmy o tym z panem przewodniczącym Henrykiem Kowalczykiem i z panią minister, że oczywiście chcielibyśmy, żeby świadczenie trafiło do jak najszerszego kręgu odbiorców. Oczywiście że stanowisko Kancelarii Prezydenta w tym zakresie jest pozytywne. Mamy świadomość tego, że po ujawnieniu pierwszego przypadku COVID na początku marca, od połowy marca te skutki w niektórych zakładach pracy już występowały, w szczególności myślę o branży turystycznej, a także innych sferach, gdzie mogło dojść do tego rodzaju sytuacji, że rozwiązanie umowy o pracę odbyło niejako z dnia na dzień. Znamy też, i państwo z interwencji poselskich, i pan prezydent z korespondencji, która jest kierowana z prośbą o wsparcie, o pomoc, tego rodzaju tragiczne sytuacje, kiedy przedsiębiorca podejmował działania niejako natychmiast, wtedy kiedy były procedowane rozwiązania prawne, które dzisiaj służą polskim przedsiębiorcom.

Dodatek solidarnościowy jest nazwą adekwatną do świadczenia, o którym rozmawiamy. To jest i dodatek, i solidarnościowy, w obu tych wymiarach ta nazwa jest adekwatna. Solidarnościowy, dlatego że to jest kwestia elementu takiego pojmowania Rzeczypospolitej, jak zresztą definiuje to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, takiego państwa, które dba o słabszych, takiego państwa, które działa w ramach zasady sprawiedliwości społecznej. Czerwiec, lipiec, sierpień. Jeszcze w tym miesiącu mogłoby to trafić do beneficjentów pomocy. Pojawiło się też pytanie o formułę elektroniczną. To jest taka formuła, która zapewnia prawidłowość, jeżeli chodzi o obsługę tych wniosków. To jest też tak, że ZUS, wskazujemy na to w uzasadnieniu, jest przygotowany, żeby przez dodatkowych pracowników i szczegółowe porady uruchamiać taką możliwość, żeby - jeżeli zgłasza się osoba, która może skorzystać z rozwiązań prawnych zawartych w tej ustawie - była pomoc w założeniu tego profilu, było wskazanie, że ten wniosek jest poprawny.

Wysoka Izbo! Wnoszę oczywiście o to, żeby poprzeć ten projekt prezydencki z uwzględnieniem zapowiadanej już poprawki, bo tego dzisiaj oczekują obywatele, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji z przyczyn przez siebie niezawinionych, z przyczyn spowodowanych utratą pracy z powodu światowej pandemii COVID-19. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Zwracam się z takim postulatem, jeśli będzie do tego potrzebna przerwa, pani marszałek, to będzie to wniosek o przerwę. Chodzi mi o to, żeby mimo wszystko traktować jednakowo wszystkich występujących, jeśli chodzi o limit czasu.

Druga kwestia to jednak pouczenie występujących o tym, żeby się trzymali swojej roli. Pani minister nie odpowiada na pytanie i tak naprawdę wchodzi w rolę wnioskodawcy. I mówimy tu o takich historycznych kwestiach. Nie był to wniosek formalny, umówmy się. A odpowiadając na pani wątpliwości: ja przestrzegam czasu i niezależnie od przynależności klubowej skracałam czy pilnowałam czasu zadania pytania. Natomiast pan minister ściśle trzymał się odpowiadania na postawione pytania w Wysokiej Izbie i trudno było ograniczać wystąpienie ministra, szczególnie że reprezentował po prostu wnioskodawców. Rząd ma prawo odnieść się tak naprawdę do każdego projektu ustawy i akurat reprezentantem. Zamykam dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania ustawy. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciw.

Wznawiam obrady. Proszę państwa, padł wniosek, który będziemy musieli przegłosować, w związku z tym pierwsze głosowanie to jest potwierdzenie kworum. Dlatego proszę państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu stwierdzenia kworum. Wniosek formalny, panie pośle, po stwierdzeniu kworum. Bardzo proszę, jest pan niezawodny w zgłaszaniu wniosków formalnych. Proszę państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu stwierdzenia kworum. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum. Proszę.

Wniosek o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji i głosowania. Mój projekt uchwały skierowanej do braci Węgrów dostarczyłem przecież zawczasu do biura pani marszałek - mam tu prezentatę - z pismem przewodnim, w którym zastrzegałem, że liczę na to, że pani marszałek sama, doceniając znaczenie tego faktu, tej sprawy, zechce. bo ma takie regulaminowe uprawnienia, przedstawić Wysokiej Izbie ten tekst, do którego ja nie roszczę sobie praw autorskich. Ale ponieważ sprawa spełzła na niczym, a stadny rechot z państwa strony. świadczył o tym, że w ogóle nie macie bladego pojęcia, o co chodzi. 100 lat temu rozebrane zostało królestwo Węgrów. Chwila ciszy po królestwie Węgrów. Przypominam panu raz jeszcze: to nie jest moje uprawnienie. 15 posłów musi się podpisać pod projektem uchwały. Panie pośle, pan napisał to indywidualnie. Proszę zebrać 15 podpisów. Proszę raczej zapoznać się z regulaminem w tej sprawie. Proszę państwa. Już się przyzwyczaiłam. Nie trzeba. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Wobec propozycji przejścia do drugiego czytania projektu ustawy zgłoszono sprzeciw. Pod głosowanie poddam propozycję przystąpienia do drugiego czytania tego projektu ustawy. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za propozycją przystąpienia do drugiego czytania projektu ustawy zawartego w druku nr 406, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek przyjął, a tym samym wyraził zgodę na przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy. Przystępujemy do drugiego czytania projektu ustawy. Otwieram dyskusję. Proponuję, aby Sejm w dyskusji w drugim czytaniu projektu ustawy wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Byłabym zdziwiona, gdyby go nie było. Proszę państwa, wobec sprzeciwu.

W związku z tym przystępujemy do drugiego czytania. Proponuję, aby Sejm w dyskusji w drugim czytaniu projektu ustawy wysłuchał 4-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam ogromny zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w drugim czytaniu projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Raz jeszcze chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość podziękować panu prezydentowi za aktywność, za to, że tak aktywnie realizuje swoją prezydenturę, za to, że po raz kolejny występuje do Wysokiej Izby ze swoim prezydenckim projektem ustawy. To bardzo ważne, że dzisiaj dyskutujemy na ten temat, że pochylamy się nad tymi, którzy dzisiaj potrzebują naszej pomocy, którzy dzisiaj potrzebują naszego wsparcia, którzy dzisiaj potrzebują naszej solidarności. Kolejny raz apeluję, aby Wysoka Izba przyjęła te rozwiązania na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Raz jeszcze chciałbym również podkreślić, że prezydentura pana prezydenta Andrzeja Dudy jest prezydenturą bardzo aktywną. Pan prezydent wielokrotnie pokazał, że jest politykiem wiarygodnym, jeżeli chodzi o to, co obiecuje w trakcie kampanii wyborczej, co obiecuje w trakcie realizowania swojej misji. W czasie kryzysu pan prezydent nie ucieka na zwolnienie lekarskie, nie ucieka na L4, ale rzeczywiście w sposób bardzo dojrzały, w sposób bardzo dobry, skuteczny uzgadnia, reaguje na konkretne problemy, dyskutuje z panem premierem, wielokrotnie spotyka się z ministrem zdrowia. Trzeba jasno powiedzieć, że po raz kolejny obywatele, Polacy nie zawiedli się na swoim prezydencie. I dzisiaj warto również powiedzieć, że są w Polsce tacy politycy, którzy naśmiewają się z programów społecznych, którzy uznają np. program 500+ za rozdawnictwo. Z drugiej strony na szczęście mamy pana prezydenta Andrzeja Dudę, na szczęście mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który nie zgadza się z takim podejściem, który pokazuje, że skutecznie można realizować swoje obietnice, te, które były składane. I w sposób skuteczny patrzy na tych, którzy potrzebują naszej pomocy, którzy potrzebują naszego wsparcia. Są tacy politycy, którzy nie dotrzymują słowa, którzy nie dotrzymują obietnic, którzy to, co mówili w trakcie kampanii, później puszczają mimochodem, i mamy takich, którzy realizują, dobrze realizują swoje obietnice. Są znowu tacy politycy, którzy proponują drastyczne podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste, którzy proponują niezrozumiałe podwyżki opłat za wywóz śmieci, i z drugiej strony mamy postawę prezydenta Andrzeja Dudy, mamy postawę rządu Prawa i Sprawiedliwości, tej bardzo dobrej współpracy pomiędzy prezydentem a premierem.

Na szczęście jest pan prezydent Andrzej Duda, na szczęście jest większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości, która skutecznie przy współudziale, przy znaczącym współudziale pana prezydenta Andrzeja Dudy wspiera seniorów, choćby poprzez program „Emerytura+” To bardzo ważne, że dzisiaj możemy jasno powiedzieć, że 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy to był bardzo dobry czas, że to był czas bardzo aktywny. I dzisiaj mamy kolejne potwierdzenie, kolejny projekt prezydencki. Bardzo proszę w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (Dzwonek), abyśmy mogli szybko go przyjąć.

Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Ja myślę, że po wystąpieniu mojego przedmówcy już nikt nie ma wątpliwości, że ten projekt był po to wniesiony jeszcze w tym momencie, z tą datą, żeby chwalić urzędującego prezydenta. Ileż trzeba mieć w sobie obłudy i hipokryzji, żeby w ogóle tak robić? Przecież państwo, gdybyście naprawdę chcieli pomóc osobom potrzebującym, to w momencie kiedy zaczęliśmy mieć do czynienia z pandemią, powinniście zaproponować kompleksowy, powszechny system wsparcia dla osób potrzebujących, a wy po trochu nam dawkujecie poszczególne tarcze i poszczególne rozwiązania. Ale jedno z rozwiązań zarezerwowaliście dla prezydenta Dudy, żeby w czasie kampanii wyborczej mógł się tym rozwiązaniem pochwalić. Tymczasem to rozwiązanie, owszem, pomaga pewnej grupie ludzi, ale jednak pomaga tylko tej grupie, która jest w mniejszości. Dlaczego państwo nie pomyśleliście o tym, żeby przyznać wyższe zasiłki osobom bezrobotnym, tak jak proponowaliśmy? Do tarczy 3.0 taką poprawkę składaliśmy, żeby ten zasiłek wynosił 1800 zł brutto, ale państwo tę poprawkę odrzuciliście. Senat 13 maja też taką propozycję złożył. Już 14 maja wy tę propozycję odrzuciliście.

Szanowni państwo, popatrzmy zatem na naszych zagranicznych sąsiadów. Tylko w Czechach, jeżeli ktoś traci pracę, to zasiłek dla niego wynosi 65% jego ostatniej pensji. W Niemczech ten zasiłek wynosi 60% ostatniej pensji. A w Polsce ile wynosi? Od 25 do 36% najniższego wynagrodzenia. Tak to wygląda. Mówicie państwo: dodatek solidarnościowy. Dla ilu tak naprawdę? Dlaczego?

Mało tego, ten dodatek solidarnościowy będzie dotyczył również osób, które mają prawo do zasiłku, i będzie ich ponad 300 tys. Więc tak naprawdę niewiele wydacie na rzecz tych osób, które tracą pracę. Natomiast jak słyszę panią minister, że ZUS daje radę, bo ten dodatek solidarnościowy będzie wypłacał ZUS. Pani minister, naprawdę, proszę zejść na ziemię i nie opowiadać tych bzdur. Przecież ZUS nawet rodzinom, które złożyły wnioski o wypłatę zasiłku opiekuńczego za marzec i kwiecień, jeszcze w maju ich nie wypłacił. I niech pani nie mówi, że nie ma takich przypadków, bo osobiście do pani napiszę o tych rodzinach, bo one do mnie piszą, bo ja je znam, i pani udowodnię, że ZUS nie daje rady z wypłatą zasiłków opiekuńczych, a jeszcze teraz państwo im dokładacie wypłatę tego dodatku solidarnościowego. Stworzyliście państwo taką hybrydę w całym systemie pomocy i w ogóle nie macie pomysłu, żeby ten system był powszechny, żeby te rozwiązania były naprawdę systemowe, tylko wszystko jest tak zdawkowe, pojedyncze, pod potrzeby kampanii wyborczej, bez patrzenia na tych, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Oczywiście, jeżeli państwo nie potrafiliście poprzeć dobrego rozwiązania, my to rozwiązanie oczywiście poprzemy, ale nie jest to rozwiązanie idealne, nie jest to rozwiązanie ani powszechne, ani systemowe. Będzie pomagało tylko określonej grupie osób, ale przede wszystkim, tak jak powiedział przedmówca, ma służyć panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie w ramach trwającej kampanii wyborczej. Przykra to prawda, ale niestety tak to wygląda. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! W dynamicznym tempie kłusujemy przez kolejne czytania. Ja chciałbym zacząć od odniesienia się do słów pani minister. Pani powiedziała, że to nie jest prawda, kiedy mówię o tym, że to jest 36% płacy minimalnej.

I to tyle, jeśli chodzi o wersję prezydencką, chyba że odnosi się pani do tego, jak pani poprzednio podniosła zasiłek. Proszę państwa, my w tym drugim czytaniu złożymy poprawki do tej ustawy, poprawki, które naprawiają te dziury, o których wspominałem w poprzednim wystąpieniu. Po pierwsze, chcemy, żeby chociaż część osób pracujących na śmieciówkach mogła skorzystać z tego świadczenia. Jest coś dziwnego w tym, że świadczenie dla pracowników jest niższe niż świadczenie dla przedsiębiorców, więc składamy poprawkę, żeby ta wysokość dodatku solidarnościowego wynosiła jednak 2080 zł na rękę, bo pracownicy nie są gorszą grupą niż samozatrudnieni i z tego musi dać się wyżyć. Trzecia sprawa to jest ten system dotyczący wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Proponujemy skromne rozwiązanie: 50% ostatniego wynagrodzenia. To jest dużo, dużo mniej niż choćby w Danii czy w innych krajach skandynawskich, ale to jakkolwiek zabezpieczy ludzi. To, co wy proponujecie w tym momencie, to jest wysokość zasiłku, która cały czas nie spełnia norm zalecanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. To cały czas jest dla wielu rodzin poniżej granicy przetrwania. Niechże ten zasiłek jak w każdym normalnym europejskim kraju przysługuje przez 720 dni, tym bardziej że wiemy wszyscy, jak tutaj siedzimy na tej sali, że problem z kryzysem ekonomicznym nie skończy się jutro, nie skończy się pojutrze, on będzie trwać długo. Znaczna część tych ludzi, którzy stracą pracę, będzie długo uzależniona od wsparcia państwa, w związku z czym przedłużmy to do normalnych ram, do europejskich norm.

Składamy te poprawki, tak żeby tę ustawę naprawić, tak żeby zabezpieczyć ludzi, którzy będą tracili pracę. I zwracamy się do państwa, żebyście te poprawki na serio rozpatrzyli, także te mniejsze, także te techniczne, takie jak ta, żeby pozwolić ludziom na skorzystanie z tego świadczenia, jeżeli mają 30 opłaconych dni składkowych.

Zachęcam państwa do tego, żeby te poprawki przyjąć, i zachęcam państwa do tego, żeby w końcu przełamać się i poddać pod głosowanie ustawę przygotowaną przez koalicyjny klub Lewicy. Rozumiem, że nie chcecie jej poddać pod głosowanie teraz, przed wyborami. Pewnie będziecie musieli poddać ją pod głosowanie jesienią, kiedy bezrobocie (Dzwonek) wzrośnie i będzie ona naprawdę bardzo, bardzo potrzebna, ale im szybciej, tym lepiej.

Nie ma pana posła Brauna. Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. O, wyjątkowa sytuacja. Oczywiście. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Słyszeliśmy tutaj z ust pana posła, jak to wspaniałomyślnie pan prezydent spełnia wszystkie obietnice. Gdyby tak było, to nie trzeba byłoby wprowadzać tego szkodliwego projektu. Gdyby pan prezydent złożył skutecznie, tak jak to teraz skutecznie zostało złożone, że - uwaga - bez komisji drugie czytanie, zaraz będzie trzecie i myk do podpisu, ustawę dotyczącą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł dla wszystkich, tak jak obiecywał, to wówczas byłoby mniejsze opodatkowanie pracy i pracodawcom bardziej opłacałoby się zatrudniać, a pracownikom bardziej opłacałoby się pracować. To rozwiązanie, które dzisiaj zaprezentował pan prezydent Andrzej Duda, jest podwójnie szkodliwe.

Państwo wyślą tysiące urzędników, żeby kontrolować? Jak teraz wszyscy przeszli na pracę zdalną, to jak państwo to skontrolują? Efekt tego będzie taki, że bezrobocie wzrośnie, a państwo jeszcze za to zapłacą. Proszę bardzo. Tak jest, coraz częściej przypomina się ten dowcip z czasów mojej PRL-owskiej młodości: Czy to prawda, że na placu Czerwonym rozdają pobiedy? Przypominam posłom młodszego pokolenia, że pobieda to był taki samochód czy samochodopodobna konstrukcja sowiecka. A więc czy to prawda, że na placu Czerwonym rozdają pobiedy? Radio Erewań odpowiada: tak, w zasadzie prawda, tyle tylko, że nie na placu Czerwonym, a Maneżowym, nie pobiedy, a rowery, i nie rozdają, tylko kradną. Wiele szumnych, niestety szalbierczych obietnic, wiele zapowiedzi, za które oczywiście przyjdzie zapłacić rodakom, Polakom, rzecz jasna nie tym, którzy będą obsługiwać te transfery wagonów pieniędzy, bo to wagonami one tutaj się przetaczają, prawda, przez tę Wysoką Izbę. Państwo tymi wagonami wieziecie te pieniądze na lotnisko, z którego startuje pani premier Emilewicz swoim wielkim helikopterem, rozsypuje je po Polsce.

Po prostu te pieniądze są coraz mniej warte. To, na co zwraca uwagę koło Konfederacja, przewodniczący naszego koła pan poseł Jakub Kulesza: jeżeli tworzymy popyt, to będzie podaż, jeżeli zachęcamy pracodawców do tego, żeby mieli mniejsze wyrzuty sumienia, zwalniając tego czy owego, jeśli zachęcamy pracobiorców do tego, żeby nie lękali się zmienić stanu zatrudnienia, gdyż będzie to jakoś amortyzowane przez władzę, to pod pozorem wielkich dobrodziejstw [[Dzwonek]] uruchamiamy spory ruch w szarej strefie. Zamykam listę posłów zapisanych do zadania pytania. Bardzo proszę. Jest pan poseł Michał Szczerba? W takim razie pan poseł Dobromir Sośnierz. Nie? Dobrze. Proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Tak zastanawiam się, jak to się stało i za jaką przyczyną.

I jak to się stało, że jednak nie poczekał do Matki Boskiej Królowej Polski, której święto w tym roku przypada następnego dnia?

Pan poseł Krzysztof Gawkowski, klub Lewicy. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ta ustawa to plagiat, plagiat, ale nieudany, plagiat, który jest kopią ustawy Lewicy o świadczeniu kryzysowym. Po pierwsze, późno, po drugie, źle. Pani minister, panie ministrze, panie prezydencie, bo to też do pana, 1 maja Lewica zgłosiła pakiet pracowniczy, szereg ustaw, które mają dawać więcej pieniędzy bezrobotnym, które mają dawać większe prawa osobom na umowy śmieciowe, które mają gwarantować prawa tym, których chcecie zwalniać przez e-maile. Dzisiaj mówimy jasno: chcemy nad tym pracować, chcemy tę ustawę przyjąć, ale na Boga, nie ośmieszajmy się, niech to nie będzie 1400, tylko 2 tys. zł. Z tym wnioskiem, z taką propozycją Lewica dzisiaj zwraca się do pani minister, do pana ministra i przede wszystkim do pana prezydenta.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! To bardzo dobrze, że pan prezydent zatroszczył się o bezrobotnych, ale powinniście się państwo wstydzić, że troszczy się o nich wtedy, kiedy zbliżają się wybory, i że po prostu proponuje kiełbasę wyborczą zamiast systemowego rozwiązania. dla tych wszystkich, którzy tracą pracę nie ze swojej winy: albo w wyniku recesji, albo w wyniku restrukturyzacji, albo w wyniku epidemii.

Szumnie zapowiadany prezydencki dodatek solidarnościowy nie jest nim. No właśnie nie jest dodatkiem do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych, to dodatek ma być pomniejszony o kwotę zasiłku.

I dodatkowy warunek, czyli w 2020 r. trzeba było wypracować co najmniej 90 dni, mieć stosunek pracy. Przykładowo, jeżeli byłam na śmieciówce, to co wtedy?

Więc w tym momencie jak to wygląda w rzeczywistości? Lewica w przypadku świadczenia kryzysowego założyła 3,6 mld zł (Dzwonek), ale na miesiąc. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Bezpośrednio po studiach pod koniec lat 90. sam byłem bezrobotnym i stałem w kolejce do rejestracji w urzędzie pracy. Co prawda nigdy zasiłku nie otrzymałem, ale jednak poznałem gorycz tego, że nie ma się pracy, a bardzo chce się pracować. W ciągu ostatniego miesiąca przybyło ponad 55 tys. bezrobotnych, ale tym wszystkim bezrobotnym potrzebna jest pomoc państwa w kreowaniu miejsc pracy, zwolnienie z podatków dla przedsiębiorców, którzy takie miejsca tworzą, a nie chwyt wyborczy sponsorowany nie z kieszeni funduszu PiS, tylko z podatków wszystkich Polek i Polaków. Dlaczego pan prezydent nie przychylił się do apelu pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem? Medycy apelowali o to, aby otrzymać 1000 zł dodatku. Na te głosy pan prezydent jest głuchy. Jednocześnie chciałbym zaapelować o rozwagę w wykorzystywaniu tytułu wielkiego przywódcy, którym w odniesieniu do prezydenta Dudy posłużył się premier Morawiecki. Pani poseł Wanda Nowicka, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od kilku miesięcy walczymy z pandemią koronawirusa, tysiące ludzi straciło pracę.

Dobrze. My chcemy pracować i Lewica mówi: sprawdzam.

Mam nadzieję, że ludzie mają świadomość, że to wszystko jest tak naprawdę kampanią przedwyborczą pana prezydenta, i nie dadzą się na to nabrać. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, klub Lewicy. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak mówią dane GUS. Duża część pokrzywdzonych tą ustawą to właśnie ludzie, którzy pracują na umowach śmieciowych. A duża część z nich to artyści, ludzie kultury i pracownicy kultury. I chciałam zapytać: W jaki sposób tarcza dla kultury, który to system w tej chwili nie działa - i to jest zgłaszane nam ze wszystkich stron, piszą do nas ludzie kultury.

Pani poseł Barbara Bartuś, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Państwo Ministrowie!

Państwo, wychodząc na mównicę, cały czas straszycie Polaków, ale żeby tylko: straszycie - wy kłamiecie. I tutaj mam pytanie do pani minister: Czy z trzynastej emerytury są dokonywane jakiekolwiek potrącenia egzekucyjne?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Bardzo dziękuję. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość składa poprawkę w tym zakresie.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Ten projekt ustawy doskonale potwierdza to, o czym dzisiaj mówiłam. Kolejny raz rządzący, tym razem w osobie prezydenta, nie zwracają uwagi na osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, których nie bójmy się nazywać śmieciowymi. Co z osobami zatrudnionymi w takiej formie? Jeżeli już nie potrafią państwo zrobić porządku z tego rodzaju umowami, tak żeby pracownicy mieli wszystkie zabezpieczenia, zgodnie z Kodeksem pracy, to chyba warto pomóc osobom pracującym na śmieciówkach teraz, w czasie kryzysu. Przymiotnik „solidarnościowy” zobowiązuje. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zadzwonił do mnie znajomy, który pracuje w biurze tłumaczeń, z prośbą o poradę podatkową. Jest zatrudniony na umowę o pracę. Całkowite koszty pracodawcy to 5 tys. zł, 40% opodatkowanie, więc ma 3 tys. na rękę.

Fajnie. Naprawdę, fajny system podatkowy tworzycie. Dzięki temu Polacy nie będą płacić tylu podatków. Niestety, posłanki Lewicy nazywają takie umowy śmieciowymi. Śmieciowa to jest Lewica, która karze ciężką pracę 40-procentowym opodatkowaniem. Te umowy cywilnoprawne pozwalają tylko na 9-procentowe opodatkowanie i to jest właśnie rozum i godność człowieka. Dziękuję bardzo. Pani poseł Mirosława Nykiel, klub Koalicji Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałabym - kieruję pytanie do pani minister Marleny Maląg - zapytać o to, czy pani zna problem z wypłacaniem zasiłków chorobowych dla mikroprzedsiębiorstw przez ZUS, bo jak pani wie, od marca problem jest bardzo wielki, są horrendalne zatory. Niestety ZUS sobie nie radzi, bo 15 tys. wniosków wpływało, a są przygotowani na 1 tys. Słyszałam, jak pani bardzo chwaliła panią prezes ZUS-u, i nie mam nic przeciwko temu, jeśli rzeczywiście było za co chwalić, ale musi pani zrozumieć tych pracowników, którzy od marca nie dostają zasiłków i mają pretensje do przedsiębiorców, że być może nie opłacają składek, tworzą się konflikty. Proszę popatrzeć oczyma tych małych przedsiębiorców, którzy siedzą w tym domu w czasie epidemii i nie dostają nawet tego zasiłku. Pan poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałoby się powiedzieć: lepiej późno niż wcale, że pan prezydent pewne działania podejmuje, ale widać, że te działania są podejmowane, bo widać strach w Kancelarii Prezydenta, widać, jak ludzie poznali się na was, że niestety nie dotrzymujecie słowa. Ale chciałem też zapytać, bo pan prezydent często mówi o dotrzymywaniu słowa, pytają o to frankowicze, kiedy wreszcie pojawi się ta ustawa, o której mówił pan prezydent równo 5 lat temu, że jednak pomoże frankowiczom i przewalutuje kredyt frankowy po cenie z dnia jego zaciągnięcia. Chciałem zapytać pana ministra Muchę, czy nie jest panu wstyd, może też panu prezydentowi, za słowa, które powiedział pod Pałacem Prezydenckim: Ojczyznę dojną racz nam wrócić, Panie. A później pani Sadurska, wiceszefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeszła do PZU i zarobiła przez 2,5 roku ponad 3 mln zł. Czy właśnie o tę dojną ojczyznę chodziło? Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym zapytać dlaczego, dlaczego partia rządząca nie skorzystała z już gotowego projektu Lewicy, który leżał już długi czas i nie doczekał się nawet numeru druku - dopiero teraz mamy nadany numer druku - pomimo że macie państwo gotowy projekt. Pytam: Dlaczego ten projekt dodatku solidarnościowego pojawia się tak późno, skoro mieli państwo gotowy projekt dodatku, świadczenia kryzysowego? Chciałam też zapytać, dlaczego nie trafił on do komisji. Czy dlatego, że jest tak dobry i nie chcą państwo nad nim pracować? Na szczęście mamy poprawki. Mam nadzieję, że zostaną uwzględnione. Dlaczego jest tak krótki okres wypłacania tego świadczenia, od czerwca do sierpnia tego roku? Czy dlatego, że będzie już po drugiej turze wyborów? Dziękuję. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan prezydent w swoim majowym wystąpieniu obiecał jednocześnie dodatek i zasiłek dla bezrobotnych, tymczasem zgodnie z tą ustawą mamy albo zasiłek, albo dodatek. W związku z tym, że pani poseł mówiła, że pan prezydent dotrzymuje swoich obietnic, liczę na to, że z jednej strony klub PiS-u, a z drugiej strony pan prezydent zmienicie tak zapisy tej ustawy, aby można było jednocześnie pobierać dodatek i zasiłek. Jeśli osobie bezrobotnej zostanie wypłacony zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, o którym mowa w ustawie, wówczas dodatek solidarnościowy wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym dodatkiem solidarnościowym a zasiłkiem lub stypendium wypłacanym przez urząd pracy. Zatem jeśli dotrzymujecie słowa, to dotrzymajcie tego, o czym mówił pan prezydent. Pan poseł Michał Szczerba, klub Koalicji Obywatelskiej. Niecodziennie mamy ministra z Kancelarii Prezydenta - pana ministra Muchę, więc skorzystam z tej okazji i zapytam o fundusz medyczny. Z wielką pompą 8 marca pan prezydent razem z panem ministrem Szumowskim ogłaszali powstanie funduszu medycznego. Nic z tego nie wyszło: funduszu medycznego jak nie było, tak nie ma. Chcielibyśmy na to pytanie znać odpowiedź. I wreszcie taka sprawa: Czy pan prezydent uważa, że sytuacja związana z konfliktem interesów pana ministra Szumowskiego jest rzeczą właściwą? Czy w tej sprawie pan prezydent jednak nie powinien zabrać głosu? Minister, premier, rodziny polityków powinni być poza wszelkimi podejrzeniami. Mam wrażenie, że państwo przymykacie oczy na tę sytuację, która jest (Dzwonek) sytuacją negatywną. Teraz o głos poprosił wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego pan Piotr Gliński. Wysoki Sejmie! Ja w charakterze ministra kultury, pani poseł, do pani. Pani poseł, z pani strony się nie spodziewałem tego. Jest ok. 30 różnych form wsparcia dla artystów w czasie epidemii. Jeżeli chodzi o osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, to nie tylko artyści, ale także każda inna osoba może otrzymać postojowe w wysokości 2080 zł miesięcznie, razy trzy to jest 6240 - każdy może dostać. Niezależnie od tego jest system zapomóg w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który powiększyliśmy wielokrotnie, ja nawet wczoraj jakieś decyzje finansowe podejmowałem w ramach naszego budżetu, 4 tys. osób już dostało zapomogę w wysokości 1800 zł.

Zwiększyliśmy także do 6,5 mln pulę stypendiów ministra, żeby także wesprzeć osoby z obszaru kultury, które są w złej sytuacji.

Tak więc wychodzenie tutaj i publiczne mówienie nieprawdy, że ludzie kultury zostali pozostawieni sami sobie, że nie ma form wsparcia. Tak to powiedzmy. Ale warto zauważyć, że faktycznie ludzie kultury zostali pozbawieni wsparcia, np. w przypadku samorządu warszawskiego.

A z tarcz antykryzysowych, z tego, co przedstawiliśmy, i co jest cały czas uzupełniane, bo tam też są specjalne rozwiązania dotyczące pomników historii wsparcia, filmowców itd.... Kazika Staszewskiego. nie będę o tym mówić, idą kolejne miliony i miliardy, bo ludzie zatrudnieni na tzw. śmieciówkach, jak państwo mówicie, na umowach cywilno-prawnych otrzymują przede wszystkim postojowe, ale także jest dla nich w tej chwili wiele innych możliwości wsparcia. Ja np. w swoim resorcie miałem 20% ludzi zatrudnionych na śmieciówkach. W tej chwili to są incydentalne, losowe przypadki wynikające z tego, że ktoś po prostu na chwilę tylko służy pracą dla resortu. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli zadekretować w Polsce uniemożliwienie ludziom zawierania umów cywilno-prawnych dotyczących dzieła czy zleconych. Ale generalnie sytuacja jest zupełnie nieporównywalna do tego, co zastaliśmy po naszych kolegach turboliberałach, którzy niewielką do tego wagę przywiązywali. Tak jest, panie pośle, jest duża zmiana w tym kierunku. Teraz głos zabierze minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Nie, nie, teraz nie jest czas na dyskusję. Bardzo proszę. Szanowni Państwo! Jeszcze raz odniosę się do tego, że to dobra współpraca rządu z panem prezydentem Andrzejem Dudą, a od początku wygrana pana prezydenta Andrzeja Dudy w 2015 r., spowodowała dobry czas dla Polski, budowanie Polski+, wsparcie dla polskich rodzin i wszystkich programów: 500+, „Dobry start”, trzynasta emerytura, obniżenie wieku emerytalnego, który państwo zabraliście. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią i jasne, czytelne, proste instrumenty przygotowane przez rząd dla ochrony miejsc pracy, dla zachowania płynności naszych przedsiębiorców i aby pracownicy dostali wynagrodzenia, to właśnie działanie naszych tarcz, które podsumowujemy. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że ponad 73 mld zł trafiło na to, aby przede wszystkim ochronić miejsca pracy, aby trafiły środki na wynagrodzenia pracowników. Cały czas mówimy, że analizujemy przedstawione instrumenty, i właśnie ta dobra współpraca z panem prezydentem, za co dziękujemy, za złożoną wczoraj ustawę. A więc dodatek solidarnościowy, który jest przewidziany w ustawie, przede wszystkim jest szerokim wsparciem.

Szanowni Państwo!

ZUS, jeżeli chodzi o instrumenty.

Padło pytanie o zasiłki chorobowe.

Szanowni Państwo! Przygotowana przez pana prezydenta ustawa przede wszystkim jest kolejnym instrumentem, który ma wspierać Polki i Polaków. Cały czas pracujemy nad tym, aby przede wszystkim ochronić miejsca pracy, bo to jest priorytet. I dlatego w tym momencie, we właściwym momencie zostaje wprowadzona ta ustawa. Dziękuję bardzo. Głos zabierze zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan Paweł Mucha. Wysoka Izbo! Dziękuję za te głosy w dyskusji, bo one odzwierciedlają to, że ta ustawa jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie społeczne.

Te głosy, które negują potrzebę tej pomocy, są naprawdę głęboko nieprzemyślane. Co do kwestii kwotowych. To jest tak, że jeżeli odnosimy minimalne wynagrodzenie do kwoty dodatku solidarnościowego, to mamy ponad 50%, bo mamy, patrząc na kwoty nawet brutto, netto, 1400 zł dodatku solidarnościowego i wynagrodzenie minimalne w wysokości 2600 brutto niespełna. Druga rzecz. W wypowiedzi pana przewodniczącego brakuje cały czas informacji o tym, że zasiłek dla bezrobotnych w tym okresie pierwszych 3 miesięcy wynosi 1200 zł. I pan przewodniczący podaje kwotę już po upływie tych 3 miesięcy, a my mówimy o tym, że zasiłek dla wszystkich bezrobotnych będzie podniesiony od 1 września. To jest zmiana oczekiwana od dawna, to jest zmiana postulowana także przez Lewicę, ale realizowana przez inicjatywę pana prezydenta. Trafnie tutaj mówił pan premier Piotr Gliński o świadczeniu postojowym, o tych elementach, które zostały przecież wprowadzone w ramach prac rządu. Od dawien dawna już funkcjonują i beneficjenci tych świadczeń te świadczenia otrzymują.

Czyli państwo chcieliście nałożyć pewien obowiązek prawny na samorząd powiatowy.

Nie sposób się zgodzić ze stwierdzeniem, że mówimy o jakimkolwiek plagiacie. Mamy takie przekonanie, że państwo mieliście intencje czy macie te intencje, które powinny odzwierciedlać to, że będziecie tę ustawę pana prezydenta popierać. Bardzo niepokojący mnie głos wskazywał, że to są rozwiązania prawne, które uzależniają wyborców. Zupełnie nie mogę zaakceptować takiego stwierdzenia jednego z państwa posłów, bo to jest taki głos, który się powtarza od czasu wprowadzenia programu 500+, takiej swoistej pychy, arogancji wobec Polaków, którzy mają niższe dochody, albo wobec tego 0,5 mln osób, które dzisiaj są uprawnione do tego świadczenia. To nie jest żadne uzależnianie wyborców od kogokolwiek. To jest pomoc państwa dla tych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji z przyczyn, tak jak mówiłem, od siebie niezawinionych, z przyczyn obiektywnych, z przyczyn związanych z występowaniem epidemii COVID-19.

W tym zakresie ta ustawa wypełnia tę rzeczywistą potrzebę, jeżeli chodzi o wsparcie tych osób, które w takiej trudnej sytuacji życiowej się znalazły.

Ona obejmuje zarówno tych, którzy mają kredyty złotowe, jak i tych, którzy mają kredyty indeksowane, denominowane. Nie różnicuje tych, którzy mają kredyty odnoszone do franka, i tych, którzy mają kredyty złotowe. Ta ustawa w tym roku także znajduje zastosowanie, jest bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! W trybie sprostowania. Jak by pan tego nie wykręcał, jak by pan tego nie obracał, to prawda jest brutalna: cały czas to jest 36%. Wszyscy eksperci mówią, że ten poziom świadczenia dla bezrobotnych jest zbyt niski. Wystarczy porównać się z naszymi sąsiadami. Wystarczy też poczytać opracowania Międzynarodowej Organizacji Pracy. W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy po doręczeniu paniom i panom posłom zestawienia poprawek. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Ogłaszam 10 minut przerwy.

Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu stwierdzenia kworum. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 390-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawiam dodatkowe sprawozdanie komisji odnośnie do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W czasie drugiego czytania na sali plenarnej w dniu 28 maja zostały zgłoszone 144 poprawki.

Z pozostałych poprawek 28 komisja rekomenduje przyjąć, resztę komisja rekomenduje odrzucić. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości, a także - w dodatkowym sprawozdaniu - poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wymienionych poprawek, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawki przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawki odrzucił. W 7. poprawce wnioskodawcy proponują zmiany do art. 27 pkt 2 projektu ustawy. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 9. i 12., zechce

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość 2. wniosku mniejszości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 18. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 75. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 77. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek

Sejm poprawki odrzucił. W 79. poprawce wnioskodawcy proponują dodać pkt 24a. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 79. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy.

Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę przyjął. Odrzucił?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 86. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 85. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Przystępujemy do głosowania.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 87. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. W 88. poprawce wnioskodawcy proponują dodać pkt 29a.

Sejm poprawkę odrzucił. Nad nimi będziemy głosować łącznie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 89. i 119., zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 93. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 95. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 96. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 99. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 100. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosowało 451 posłów. Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 102. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił.

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 105. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 106. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 108. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przyjęcie tych poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 110. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 109. i 114., zechce

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o jej odrzucenie.

Sejm poprawkę odrzucił. W 111. poprawce wnioskodawcy proponują dodać pkt 50a. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 111. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. W 112. poprawce wnioskodawcy proponują dodać pkt 51a. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 112. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 113. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 115. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 390, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Powracamy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Sejm przeprowadził pierwsze czytanie oraz podjął decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy. Zestawienie zgłoszonych w trakcie drugiego czytania poprawek zostało paniom i panom posłom doręczone. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość 2. poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do głosowania.

431 - za, 10 - przeciw, wstrzymało się 5. Sejm poprawkę przyjął.

Sejm poprawkę odrzucił.

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. W 8. poprawce wnioskodawcy proponują zmianę redakcyjną. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Poprawki 9. i 10. zostały zgłoszone do art. 15 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 406, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ogłaszam 3 minuty technicznej przerwy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (druki nr 398 i 403)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o wotum nieufności wobec ministra Łukasza Szumowskiego - chyba największego zawodu ostatnich miesięcy, człowieka, który udawał nadzieję, a kiedy opadły maski, zobaczyliśmy twarz, prawdziwą twarz rządu PiS. Twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa. Nie dał pan rady. Kolejki do lekarzy - nadal długie. Brak pielęgniarek, salowych i położnych. Kryzys lekowy - kolejne pana fiasko. A polski Internet aż huczy od zbiórek na dzieci, na chorych ludzi, na sprzęt medyczny. To również pana wina. Nie przygotował pan kraju na pandemię. Brak środków ochrony zarówno dla personelu medycznego, jak i dla chorych w szpitalach. Brak przemyślanego procesu zamrażania i brak strategii rozmrażania.

W milczeniu patrzył pan, jak miliardy szły na telewizję publiczną, i nie przeszkadzało panu, że te pieniądze mogły trafić do chorych na raka, a nie trafią. Głosował pan przeciwko zwiększeniu testowania lekarzy i pracowników służby zdrowia - jako jeden z nich czy jako zdrajca tej grupy zawodowej? Ale klaskał pan, kneblując usta lekarzom, kneblując usta epidemiologom, zwalniając ludzi za mówienie prawdy, w tym np. pielęgniarki, które mówiły, jak wygląda sytuacja w szpitalach. To, że w Polsce jest tak nisko krzywa zachorowań, że się wypłaszcza, to wcale nie jest zasługa pana ani pańskiego rządu. Niech pan sobie nie przypisuje zasług obywateli. To, co się wydarzyło, to wielka zasługa Polek i Polaków. To oni pomogli ludziom.

Panie marszałku, inaczej wyglądała kiedyś powaga Sejmu.

Panie Marszałku! Zanim zacznę mówić, chciałam powiedzieć, że lepsizm pana prezesa słyszałam już parę razy. Wtedy kiedy wchodził na ten cmentarz, na który ja wejść nie mogłam, bo wtedy jego ból był większy od mojego. Na ten sam cmentarz, na którym leży moja matka, ofiara katastrofy smoleńskiej, on wszedł składać kwiaty swojej matce i swojemu bratu, a inni nie mogli. Pani poseł, proszę przejść do tematu.

Po raz kolejny widzimy to, czym jest PiS. Nowa solidarność buduje się wśród ludzi, tych obrażanych i poniżanych, tych, którzy wspierali chorych, tych, którzy szyli maseczki. A PiS zaprezentował nam po raz kolejny swoją dojną zmianę. Arogancja, którą widzieliśmy tutaj na sali, korupcja, nepotyzm - to są wasze imiona, nowa elito z PiS. Chcecie przykładów? Pan minister Szumowski, reprezentant tej elity, Agencja Badań Medycznych.

To jest konflikt interesów.

A teraz jakie są tego efekty? W jednym z wniosków czytamy: Wdrożenie wyników projektu nastąpi poprzez sprzedaż licencji globalnej firmie farmaceutycznej. Przedsiębiorczy pan minister, zgodnie zresztą z instrukcjami koleżanki z rządu, uznał, że pandemia to czas na dorobienie się dla przedsiębiorców. Ale najpierw zabezpieczył ich, zabezpieczył ich kodeksowo, tak żeby urzędnicy nie ponosili kary. I poszło: respiratory, dziwne zakupy, zawyżone ceny. Narciarze i sprzedawcy oscypków zarobili 220 tys. na pośrednictwie między hurtownią w Rzeszowie a Ministerstwem Zdrowia. Ministerstwo mogło dokonywać tych zakupów samo. Czemuś zarabiali znajomi ministra. Ale ona, w przeciwieństwie do pana Szumowskiego, stanęła na wysokości zadania. Ooo!... ...i nie kupiła wadliwych szczepionek, choć chcieliście ją straszyć prokuraturą, [[Oklaski]] a w każdym województwie było sztuczne płuco. Ile wtedy firm padło? Ilu narciarzy się dorobiło? Na szczęście żaden narciarz. Mówimy: mamy dość. I Polacy, i Polki mają dość tego, co uprawiacie, tych konfliktów interesów, które kryjecie i które będziecie firmować, korupcji, nepotyzmu, tej waszej dojnej zmiany. Ja wiem, że dziś obronicie pana Szumowskiego, ale jego grzechy spadają na was, jego niedopatrzenia, konflikty interesów. Ludzie widzą, że go kryjecie. I ludzie was rozliczą szybciej, niż wam się to wydaje. I to jest twarde zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej. Nie śmiejcie się. O, przepraszam, przepraszam. Poproszę teraz pana posła Tomasza Latosa o przedstawienie opinii komisji. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chciałbym przedstawić sprawozdanie komisji co do druków nr 398 i 403 dotyczących wotum nieufności dla ministra zdrowia. Komisja po długiej, wnikliwej debacie rekomenduje odrzucenie, negatywne zaopiniowanie wniosku o wotum nieufności dla ministra. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy pan poseł Przemysław Czarnek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam wyjątkowy zaszczyt i honor. Ha, ha, ha! ...w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość [[Oklaski]] przedstawić stanowisko. w sprawie wotum nieufności, wniosku o wotum nieufności dla najlepszego ministra zdrowia w historii Rzeczypospolitej Polskiej. Byłoby to stanowisko wobec wniosku o wotum nieufności, gdyby nie fakt, że to, co państwo tutaj napisaliście, i to, co zostało potwierdzone przez moją przedmówczynię, przez panią poseł w sposób skandaliczny, obelżywy i chamski. To nie jest wniosek o wotum nieufności, to jest klasyczny paszkwil. Fundament numer jeden.

Pan poseł Rutnicki - ostrzegam pana po raz drugi. Fundament numer jeden. Pan minister Łukasz Szumowski nie przygotował Polski na pandemię - szereg zaległości, szereg złych decyzji, które doprowadziły do tego, jak tutaj piszecie, że naraziło to Polaków na zagrożenie, na masowe choroby spowodowane koronawirusem. To jest paszkwil, o którym wszyscy Polacy już wiedzą. Wam to po prostu wszystko nie pasuje do faktów i do rzeczywistości. A rzeczywistość jest absolutnie jednoznaczna i fakty są jednoznaczne. Dzięki pracy Łukasza Szumowskiego w Polsce uratowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich. Nie tylko to poczęte. Nie zauważacie, że w Polsce mamy tysiąc ofiar koronawirusa. To jest o tysiąc za dużo. Każdej ofiary szkoda. Ubolewamy i składamy kondolencje rodzinom wszystkich ofiar. Ale 1 tys. to nie jest trzydzieści parę tysięcy jak we Włoszech, to nie jest 27 tys. jak w Hiszpanii, to nie jest ponad 4,5 tys. jak w Szwecji, do której odwoływali się niektórzy koledzy z Konfederacji. Wiecie, dlaczego w Polsce jest mniej? Bo Łukasz Szumowski to jest lekarz z prawdziwego powołania, z krwi i kości, lekarz oddany pacjentom, świetny kardiolog. Ale przede wszystkim Łukasz Szumowski to jest człowiek wychowany na wartościach chrześcijańskich, to jest człowiek, który zasuwał do szpitali, kiedy brakowało lekarzy, i zawsze pracował tam za darmo. Tego nie dostrzegacie. Co najważniejsze, Łukasz Szumowski oprócz wychowania przez swoich rodziców i wzrastania wśród swojej znakomitej rodziny był wolontariuszem razem ze swoją żoną, którą też obrzucacie błotem bezczelnie i chamsko. był wolontariuszem, który pracował u boku św. matki Teresy z Kalkuty i ratował ludzi w Indiach za darmo. jest właśnie Łukasz Szumowski, ale wam to wszystko nie pasuje, bo wy byście chcieli, żeby w Polsce było 30 tys. ofiar, żeby w Polsce koronawirus był wcześniej. Wam to nie pasuje do teorii spiskowej, wam to nie pasuje do waszych haseł do dzisiaj forsowanych. Stan klęski żywiołowej. Nie ma klęski. Nie pasuje wam to do waszych tez.

które są wiodące, jeśli chodzi o rynek biotechnologiczny, i które mają świetne wyniki w badaniach. Wiecie, nad czym? Nad lekami na choroby nowotworowe dla Polaków, tańszymi i skuteczniejszymi. Z wielkimi osiągnięciami. Ale uderzacie w niego, fałszywie i obelżywie mówiąc w mediach. Są tutaj ci posłowie, widzę ich na sali: pan poseł Kowal, pan poseł Urbaniak, którzy mówią, że Łukasz Szumowski zarobił na pandemii 140 mln zł. To jest kompletne pomieszanie wszelkich kłamstw, jakie rzucaliście. Nie powiecie Polakom, że w OncoArendi udział Marcina Szumowskiego, brata pana Łukasza Szumowskiego, jest tylko 9-procentowy. Nie powiecie o tym, że za czasów waszych rządów OncoArendi uzyskiwało osiem dofinansowań z NCBR-u na osiem złożonych, a od kiedy Łukasz Szumowski jest ministrem, w czterech przypadkach tego dofinansowania nie było. Nie powiecie, że zatrudnionych w tej firmie jest 90 osób, [[Dzwonek]] że 80 to są naukowcy. Tego nie powiecie, bo to wam nie pasuje do waszej fałszywej tezy. Ostatnia rzecz. Chcecie oskarżyć Łukasza Szumowskiego o to, że jest uwikłany z jakimś Danielem O. Łukasz Szumowski jest jednym z tych, którzy padli ofiarą nierzetelności człowieka, który spowodował, że zespół lekarzy pracował za darmo i bez efektów - przez rzetelność człowieka, który później został o coś innego oskarżony - i przez to chcecie go usunąć z Ministerstwa Zdrowia, najlepszego ministra. Wstyd i hańba. To są obłudne i absolutnie niewiarygodne rzeczy, to, co robicie z Łukaszem Szumowskim. Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chcę panu złożyć naprawdę wielkie wyrazy uznania i wdzięczności. Chcę panu powiedzieć, że robimy to nie sami, tylko w imieniu milionów Polaków, którzy modlą się za pana i za pana rodzinę obrzucaną błotem.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Czy ma być TKM, czy ma być otwarta dla każdego Polaka? Przynajmniej niech pan zachowa szacunek dla tych cytatów, które w tej chwili przytoczyłem, bo pan nie wie, kogo ja cytuję. Chciałbym, po pierwsze, zwrócić się do panów dżentelmenów. Jestem tym oburzony. Powiedzcie zwykłe „przepraszam” za to, że w momencie kiedy na tej sali mówiła. Jeśli pan minister Gliński żąda szacunku dla urzędu ministra, to, panie ministrze, panie premierze, niech pan pierwszy pokaże, że ma pan szacunek dla posłanki Rzeczypospolitej, niech pan zmieni te standardy, niech pan nie stoi tyłem, kiedy ona mówi. Proszę do mnie teraz nie mówić. Pan będzie miał swój czas. To są retoryczne pytania do pana, żeby się pan zaczerwienił.

Myśmy w panu widzieli lekarza, a pan szukał sposobu, jak przeprowadzić głosowanie zamiast wyborów. Gdy myśleliśmy, że naprawdę chodzi o szukanie dobrych rozwiązań na czas epidemii, rząd witał chińskie maseczki i ośmieszał Polskę na arenie międzynarodowej - premier i najważniejsze osoby na lotnisku, przed samolotem z maseczkami, które okazały się wadliwe. To było niepotrzebne. Gdy w rządzie trwała wielotygodniowa debata, jak przedłużyć władzę obecnego prezydenta, gdy Wojska Obrony Terytorialnej dostawały zniżkę na Orlenie, ktoś zapomniał o lekarzach i pielęgniarkach, a ich najwięcej było poszkodowanych w tej pandemii. Ja doskonale rozumiem, co to znaczy domniemanie niewinności. Ale też my wszyscy na tej sali rozumiemy, co to znaczy konflikt interesów. i wiemy, jak dzisiaj Polacy bardzo potrzebują, żeby władza była czysta jak łza. I to nie chodzi o to, żeby pan nam coś wyjaśniał. Nie chodzi o to, żeby państwo posłowie teraz na mnie krzyczeli. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć na każdą wątpliwość każdemu obywatelowi i żeby wreszcie coś w Polsce powiedzieć na poważnie. A więc władza, panie premierze, musi być czysta jak łza i ludzie muszą mieć pewność, że w trudnych czasach nikt nie zarabia nieuczciwie. Pan wie, co to znaczy w 1 dzień zarobić 4 mln na czysto? Przecież Polacy to słyszą.

zamknięte uszy. Są one symbolem zepsucia, są symbolem grzechu, są symbolem samowoli władzy. Kiedyś do was dotrze to, że w momencie kiedy stawialiśmy te pytania, to stawialiśmy pytania w interesie, żeby każdy mógł wyjść potem na ulice Warszawy i każdego miasta i patrzeć spokojnie w oczy obywatelom.

W grze, panie pośle, jest dzisiaj obraz Polski. W grze jest obraz Polski, jaka ona ma być, czyja ma być ta Polska. Ona nie ma być jednej partii, ona nie ma być TKM. I teraz te dwa słowa do Polaków. Nie przejmujcie się tym, co się tutaj dzieje, drodzy, kochani obywatele. Jeszcze będzie normalnie, będzie jeszcze inna Polska.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W Polsce nie jest zabronione być milionerem i zajmować stanowisko ministra jednocześnie. Zabronione jest natomiast wykorzystywanie stanowiska ministra, żeby zostać milionerem. I tak właśnie postrzegany jest dzisiaj pan minister Szumowski. To są te dowody.

To jest tupet. Jakby tego było mało, pan minister robił jeszcze inne interesy na boku. Zapomnieliście o tym? Były też respiratory od handlarza nielegalną bronią. Bezużyteczny szmelc, którego nie dało się wykorzystać, a który kosztował setki tysięcy złotych. Ciekawe, czy pan minister takie zakupy robi też, jak kupuje warzywa. Chodzi do sklepu z narzędziami? A może chleb kupuje u wulkanizatora? Może to w PiS-e jest normalność? Z panem Szumowskim miało być inaczej. Przez chwilę nawet wszystkim wydawało się, że jest inny. Ja również w to uwierzyłem. Dałem się przekonać, że minister z PiS-u będzie pracował, nie będzie interesował się władzą, pieniędzmi. Byłem przekonany, że po nocach, kiedy te worki pod oczami rosną, to jest praca przeciwko temu wszystkiemu, co niesie epidemia. Okazało się jednak, że te worki pod oczami pan minister miał dlatego, że były to worki wypełnione pieniędzmi. Szybko zaczęło wychodzić na jaw, ile tak naprawdę warta była praca pana ministra Szumowskiego.

Brak waszych kryteriów organizacji, brak kompetencji - to jest wasza, państwa PiS-u, kompromitacja. Nie zapewnił pan, panie ministrze, szpitalom odpowiedniego sprzętu, maseczek, kombinezonów, rękawiczek. Maseczki do szpitali musiały sobie pielęgniarki szyć same albo pomagali im obywatelki i obywatele. Mieliśmy przez to kilka razy więcej zachorowań wśród personelu medycznego niż w Unii i pan to doskonale wie. Zamykaliście całe oddziały. Narażaliście ludzi, którzy tam pracują i którzy tam się leczą. Gdy medycy adaptowali maski do nurkowania chałupniczym sposobem albo robili sobie przyłbice z ręczniczków papierowych, Agencja Rezerw Materiałowych sprzedała ponad 60 tys. profesjonalnych masek po zaniżonych cenach. To nie może być zapomniane. Taka była sytuacja i taka jest prawda. To jest wasza nieudolność. A o tym, jak nadchodziła epidemia, w styczniu z tej mównicy mówiła Lewica. Co mówił? Panikujecie. Z tej mównicy pan minister. I kto miał rację, panie ministrze? Może warto dzisiaj przeprosić i uderzyć się w pierś, bo w styczniu nam pan minister mówił: Nie macie racji. To jednak nie wszystko. decyzje, tarcze, brak kontroli nad rynkiem wyrobów medycznych. Pan minister dostał nawet specjalne kompetencje, które upoważniały go do tego, żeby reglamentować leki. Co zrobiliście? Jedno takie rozporządzenie. Reszta obrotu - na żywioł. To jest prawda o waszych rządach. Musicie. Dlaczego? Jak nie było klientów, nie trzeba było nosić masek. Jak znaleźli się klienci, to trzeba było zakładać maski. Wszyscy się o tym dowiedzieli. Więcej pieniędzy na sprzęt, płace dla pielęgniarek, więcej miejsc na uczelniach wyższych, żeby kształcić lekarzy. Przynajmniej 7% PKB na zdrowie. A co z tym robi PiS? Wiem, że was to męczy. Żadnej pomocy dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych. Szpitale pozostawione same sobie, a pacjenci skazywani na śmierć. Maska pana ministra Szumowskiego opadła, i to na dobre. Lewica będzie głosowała za odwołaniem pana ministra.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku chciałbym się upomnieć o szacunek dla pani posłanki Barbary Nowackiej. Z panią Barbarą Nowacką mamy w wielu sprawach bardzo różne poglądy, natomiast to, jak się państwo wobec tej posłanki zachowali, jest niegodne. Szanowni Państwo! Zaufanie to jest sprawa dla wielu ludzi święta, najważniejsza na całym świecie. Zaufanie, szczególnie do lekarza, to jest rzecz niezwykle ważna. Dlatego byłem niezwykle zdziwiony, kiedy przeczytałem w Internecie, że ludzie pisali prośby o porady lekarskie do doktora House’a, który jest aktorem. Pan miał obiecujący początek, pan mógł być podczas tej epidemii polskim doktorem House’em. ale niestety pan zawiódł i zmarnował tę szansę. Dzisiaj taki list o poradę do pana może co najwyżej napisać fan serialu „Szpital na Ale dlaczego tak się stało z tym pana zaufaniem? Pierwsza sprawa: bagatelizowanie problemu. Na początku pana wypowiedzi na temat maseczek, czy są potrzebne, czy niepotrzebne.

Nie zrobiliście tego. Później braki w przygotowaniu do epidemii, mimo że pan jeszcze 28 lutego w Telewizji Polskiej mówił, że jesteśmy przygotowani, że są zakupione testy, że są uruchomione rezerwy materiałowe, że stworzyliście państwo instrukcje, które zostały wysłane przez NFZ do każdego szpitala. Jak przyszedł koronawirus, pojawił się chaos we wszystkich placówkach. Dyrektorzy nerwowo szukali respiratorów, a sprzęt ochrony osobistej najczęściej docierał do szpitala poprzez stowarzyszenia i osoby dobrej woli. Podjęliście państwo bardzo wiele złych decyzji o charakterze strategicznym. Myślę tu chociażby o wyznaczeniu szpitali jednoimiennych na Podlasiu czy w Małopolsce.

To samo, jeżeli chodzi o Małopolskę. Mieliście do wyboru wiele szpitali w Krakowie. Wybraliście ten najważniejszy, najsilniejszy w Krakowie, blokując jego bardzo wielkie możliwości. Nie mieliście żadnego pomysłu, jak w czasie pandemii wykorzystać niepubliczny sektor ochrony zdrowia, farmaceutów i ich apteki. To były błędy strategiczne, ale to, co chyba dotknęło ludzi najbardziej, to niekonsekwencja. Maseczek nie ma? Są niepotrzebne. Maseczki przyjechały? Wszyscy mają obowiązkowo je nosić, wszędzie mają obowiązkowo je nosić. Wybory? Nie. W normalnym trybie bezpieczne będą tylko za 2 lata, a najlepiej po wynalezieniu szczepionki. Najbardziej w tej postawie boli mnie to, że pan minister Szumowski ponad swoją ogromną wiedzę medyczną, ponad swoją profesurę postawił te nakazy, które dostaje z Nowogrodzkiej. Później wszystko zaczęło się kręcić dookoła polityki.

Jeżeli to się sprawdzi, a uważam, że powinny zbadać to odpowiednie instytucje, będzie to wielki kłopot nie tylko dla pana, ale i pana obozu. Natomiast ja wyciągnąłem z tego jeszcze inny wniosek. Tak naprawdę pan się marnuje na funkcji ministra zdrowia.

Uważam, że do tej sprawy powinniśmy podejść rzetelnie, z całym szacunkiem do dorobku pana ministra Szumowskiego.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Oczywiście wypada przy tej okazji wyrazić głębokie zażenowanie, szanowni państwo.